Panie i Panowie Posłowie!

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Grzegorz Braun, koło Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle. Szczęść Boże! Wniosek formalny o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów i przeprowadzenia dyskusji zmierzającej do wniosku praktycznego, jakim byłoby zaprzestanie reglamentacji dostępu do tej sali, dostępu, który jest ograniczany arbitralnie, nieregulaminowo, nieustawowo, z naszego punktu widzenia bezprawnie, albowiem reglamentacja dostępu do tej Izby jest w jaskrawy sposób sprzeczna z obowiązkami posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Zatem każdy, kto takie regulacje wydaje, i każdy, kto je egzekwuje, godzi w obowiązek i prawo posła do wykonywania jego mandatu. Koło Poselskie Konfederacja jest w tej Izbie bardzo konsekwentnie przez Prezydium Sejmu sekowane.

Bardzo proszę, skończcie państwo z tą szopką, skończcie państwo z tą praktyką, która parlamentaryzm w Polsce redukuje do fasady, dekoracji. Zarządźcie przerwę i czym prędzej wycofajcie się z tych złych, szkodliwych i bezprawnych rozwiązań. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Proszę o zadanie pytania panią poseł Dorotę Niedzielę. Bardzo proszę. Tu, na tej sali, 3 kwietnia 2019 r. podczas debaty nad wotum nieufności wobec ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego obiecałam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będę broniła stadniny koni w Janowie Podlaskim przed nieudacznikami, którzy czego się nie dotkną, to zniszczą. I po 15 miesiącach znowu muszę stanąć w obronie Janowa Podlaskiego, bo zapaść finansowa spółki się pogłębia, a warunki higieniczne w stadninie, w jakich przebywają zwierzęta, wołają o pomstę do nieba. Widziałam to na własne oczy podczas wizyty interwencyjnej 19 maja. Zaraz minister Ardanowski powie mi, że nie wiem, co widziałam, i będzie mówił, że wszystko jest w porządku.

Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę podziękować za to pytanie, oczywiście z tezą, ponieważ to pozwoli chociaż krótko wytłumaczyć stan stadniny i - pani może w to i tak nie uwierzy - przedstawić pewną obiektywną ocenę jej stanu. W Polsce kochamy konie - to jest nasza duma narodowa - szczególnie konie arabskie. Historycznie dzięki Polsce, polskim magnatom zostały te konie uratowane, dlatego troska o stadniny zajmujące się końmi arabskimi jest absolutnie uzasadniona. Ja nie będę odpowiadał pani moimi ocenami, ponieważ, jak już pani stwierdziła, one będą subiektywne, bo pani wie lepiej. Przeczytam kilka dokumentów, które inni, niezwiązani ze mną ludzie, osoby, instytucje przedstawili. Przewodniczący Przyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Janowie, jako żywo ze mną niezwiązany, pisze: W przestrzeni ostatnich dni wszystkie główne media krajowe, jak i zagraniczne, nie tylko prasę branżową, obiegła wiadomość, iż w Stadninie Koni Janów Podlaski wystąpiła sytuacja „skrajnego zaniedbania zwierząt” Według pań posłanek Doroty Niedzieli i Joanny Kluzik-Rostkowskiej konie, jak i krowy, są skrajnie zaniedbane. My jako organizacja związkowa musimy zdementować te informacje. To nie moje sformułowanie. Pokazywanie negatywnych wydarzeń w stadninie koni w ciągu ostatnich lat jest wykorzystywane do zwalczania się partyjnych ugrupowań. Zawsze na wiosnę konie wyglądają gorzej. Faktem jest, że część zebranego siana była złej jakości. Jezus Maria... ...a słaby odrost traw na pastwiskach z powodu zimnych dni i suszy spowodował przedłużające się przebywanie koni w stajniach i konieczność dłuższego karmienia ich sianem, co odbiło się na ich kondycji. Także kłopoty z powodu braku własnego podkuwacza i brak możliwości, z przyczyny koronawirusa, zatrudnienia podkuwaczy z zewnątrz poskutkowały brakiem bieżącej pielęgnacji kopyt u części koni. Fakty te skrzętnie zostały wykorzystane przez polityków do pokazania stadniny w złym świetle. Apelujemy do opozycji i mediów o opamiętanie się i nieniszczenie ludzi, w tym przypadku ciężko pracującej załogi stadniny koni w Janowie Podlaskim, a wszelkiej maści politykom - myślę, że to jest do pań posłanek - przypominamy, że żyją z ciężkiej pracy robotników rolnych. Teraz, proszę państwa. Pani poseł, możemy się przekrzykiwać, ale to nie ze mną. To nie ze mną. Teraz mit o znakomitym prowadzeniu stadniny w minionych latach przez odwołanego przez Krzysztofa Jurgiela poprzednika. Powinno mieć dobre wyniki, chociaż hodowla koni nie jest w Polsce działaniem dochodowym, szczególnie w wydaniu państwowym, gdzie trzeba zachowywać zasób genetyczny, a nie patrzeć tylko na sprzedaż koni.

To były lata, kiedy przysługiwały podwyższone dopłaty zabrane przez ministra Sawickiego. Chociaż takie były przepisy unijne i capping był w całej Europie stosowany, Polska mogła, nie musiała się do tego przyłożyć. Czyli te wyniki były w czasach, kiedy były dużo wyższe dopłaty bezpośrednie. Słynny 2015 r., euforia, znakomity wynik finansowy.

Jednej polskiej klaczy. Sprzedażą, która nosi znamiona wręcz hodowlanej głupoty, bo nie sprzedaje się najlepszych koni. Nie sprzedaje się najlepszych koni. Sprzedaje się córki, a nie matki. Sprzedaż Pepity w tym roku uratowała wynik finansowy, bo 2015 r., przypomnę, był trudnym rokiem z powodu suszy, wspominaliśmy o tym wielokrotnie, i wyniki finansowe dramatycznie się w stadninie pogorszyły, również ze względu na zabranie dopłat bezpośrednich. W związku z tym o jakich tu wielkich sukcesach pana Treli możemy mówić? Wynik finansowy w 2019 r. - państwo już wiecie, bo się nim posługujecie, jakieś miliony wymyślacie - został poprawiony w stosunku do roku poprzedniego o 2700 tys. zł. Więc chcę tu powiedzieć: te wszystkie zarzuty, nie chcę złych słów używać. Panie marszałku, jeszcze zdanie. te wszystkie zarzuty, które są stawiane, są wyssane z palca. To są zarzuty nieprawdziwe. Na początek czerwca zapraszam wszystkich dziennikarzy na konferencję prasową, gdzie zostaną przedstawione szczegółowe dokumenty.

Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. Ja tutaj mam pismo z ubiegłego roku, z maja. KOWR już wtedy pisał, że jeżeli chodzi o hodowlę bydła, w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta, ściany są wilgotne, zabrudzone odchodami. Odchody zwierząt nie są usuwane odpowiednio często. Zabrudzone odchodami są zwierzęta w różnym wieku. Rok temu, w maju, sytuacja w Janowie już była bardzo trudna. Może pan oczywiście tutaj nas czarować.

Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Najwyższa Izba Kontroli pod rządami pana Kwiatkowskiego, chyba nie sojusznika Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadziła analizę w spółce w 2019 r. i w zaleceniach pokontrolnych stwierdzono: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie - czyli dotyczącym tych zwierząt - nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec braku stwierdzonych nieprawidłowości odstępuje się od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Stadnina jest tak dramatycznie zła, że ci, którzy ją nagradzają, nie wiedzą, co czynią?

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje w mediach polskich i zagranicznych przedstawiają bardzo krytycznie obraz hodowli koni arabskich w Polsce, a co za tym idzie - mają wpływ na ich wartość na rynkach światowych. Podejrzewamy, że pośrednicy zajmujący się sprzedażą naszych koni są zainteresowani obniżeniem ich wartości i poprzez zaangażowanie w ten atak w efekcie są w stanie uzyskać znacząco większe zyski ze swojej działalności handlowej. Hejterzy, przedstawiając w bardzo krytyczny sposób obraz hodowli koni arabskich w Polsce, mają negatywny wpływ na ich wizerunek, a co za tym idzie - na wartość i ceny koni pochodzących z polskiego programu hodowli koni arabskich. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Dorota Niedziela. Znany jest pan z tego, że nie umie pan mówić prawdy. Kłamał pan, kłamie i będzie pan kłamał.

Przeczytam panu: W poidle dla krów dojnych woda wymieszana z odchodami, w nawiasie: gnojówka, brak zapasów pasz objętościowych, sianokiszonka w silosie organoleptycznie przypomina obornik. Czy to jest według pana dobrze prowadzone gospodarstwo bydła? Może panu pokażę. Cielęta mają biegunkę, kaszlą i są chore, są zaniedbane. Dziękuję bardzo. Przedstawię bardzo precyzyjne dane, również odnośnie do zdjęć, które panie tam wykonywały. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Marek Polak zada pytanie w sprawie skali przemocy domowej w Polsce i rozwiązań wprowadzonych przez ustawę antyprzemocową. Pytanie jest skierowane do ministra sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Blisko miesiąc temu Sejm niemal jednogłośnie przyjął przygotowaną przez resort sprawiedliwości ustawę pozwalającą na zobligowanie sprawcy przemocy domowej do natychmiastowego, przymusowego opuszczenia mieszkania. To odpowiedź m.in. na nierzadką potrzebę niezwłocznego przerwania przemocy przez odizolowanie ofiary od sprawcy. Myślę, że to bardzo dobra ustawa, bo w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia ofiary daje możliwość udzielenia jej realnej pomocy już w chwili interwencji Policji, zapewniając jednocześnie godne życie w czasie oczekiwania na rozpatrzenie tej decyzji przez sąd. Ale ja chciałbym zapytać pana ministra: Jaka jest skala osób dotkniętych przemocą w Polsce i ile osób według szacunków ministerstwa będzie mogło skorzystać z szybkiej i skutecznej pomocy na mocy tej ustawy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania, które mają na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania sprawcy przemocy od ofiary przemocy właśnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia dla życia lub zdrowia domownika. To jest właśnie jeden z nowych instrumentów w polskim porządku prawnym, tzn. nowe uprawnienie dla Policji, również odpowiednio dla Żandarmerii Wojskowej, uprawnienie do wydania wobec osoby stosującej przemoc natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego najbliższego otoczenia. To oznacza, że to właśnie sprawca przemocy będzie musiał natychmiast opuścić mieszkanie, a nie ofiara, jak to miało miejsce dotychczas i wcześniej, oraz nie będzie już sytuacji, w których ofiara przemocy będzie musiała pozostawać pod jednym dachem ze sprawcą.

Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące „Niebieskich kart”, to w 2019 r. mieliśmy do czynienia z nieco ponad 88 tys. osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, z czego 65 tys. to kobiety, 12 tys. to osoby małoletnie, nieco ponad 10 tys. - mężczyźni. Jeżeli chodzi o pewne szacunki, bo oczywiście nie mamy tutaj żadnych twardych danych, zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem pogotowia „Niebieska linia”, to określa się, że ok. 10% wszystkich zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie wymagało pilnej interwencji służb, m.in. ze względu na zagrożenie życia.

Jeżeli chodzi o twarde dane, to najwcześniej po pół roku, po roku od wejścia w życie ustawy będziemy mieli miarodajne dane odnośnie do liczby osób dotkniętych przemocą i korzystających z rozwiązania w postaci natychmiastowego nakazu policyjnego.

Jesteśmy również w stałym kontakcie z odpowiednimi jednostkami Komendy Głównej Policji oraz Żandarmerii Wojskowej, tak aby te statystyki były ze sobą skorelowane. Istotne też jest stosowanie dotychczasowych narzędzi izolacji sprawcy od ofiary, narzędzi cywilnych i karnych.

Na marginesie mogę dodać, że średnio jedną sprawę sąd rozpatrywał 134 dni. To też jest ważna informacja, bo w tej nowelizacji, która został podpisana przez pana prezydenta, wprowadzamy również rozwiązanie, które to postępowanie cywilne usprawni, tak żeby w jednej instancji postępowanie trwało maksymalnie 30 dni. W 2018 r. było łącznie nieco ponad 2600 takich postanowień.

To jest realne działanie, dzięki któremu Polska dołącza do krajów, w których ochrona ofiar przemocy jest najskuteczniejsza. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Bardzo dziękuję za te szczegółowe statystyki i dane. Jak już powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, to bardzo dobra ustawa. Choć to potrzebna regulacja, pojawia się jednak pytanie: Czy tak daleko idące uprawnienie dla poszczególnych organów nie będzie nadużywane? Mam tu na myśli skutek powstały w wyniku ewentualnych fałszywych oskarżeń o przemoc domową w celu łatwego pozbycia się niechcianego domownika. I w związku z tym chciałbym zapytać: Czy w takich sytuacjach osoby eksmitowane będą musiały dochodzić swoich praw w sposób zwyczajowy, przed sądem, co - jak wiadomo - może trwać nawet kilka miesięcy, czy też będą mogły skorzystać z przyspieszonego, określonego trybu rozpatrzenia tych ewentualnych zażaleń? Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! To rzeczywiście jest ważne zagadnienie, nad którym bardzo szczegółowo się pochylaliśmy w trakcie prac nad projektem przedmiotowej ustawy.

A więc powtarzam: to jest bardzo krótki termin, sąd będzie zobowiązany w ciągu 3 dni rozpatrzyć zażalenie, które może być złożone przez osobę, w stosunku do której wydano nakaz policyjny. Tutaj mówimy o nakazie opuszczenia mieszkania, który na podstawie nakazu policyjnego albo Żandarmerii Wojskowej będzie obowiązywał tylko przez 14 dni, a przedłużenie może być dokonane tylko i wyłącznie na drodze sądowej, właśnie w ramach odrębnego postępowania cywilnego, które również w tej ustawie zostało szczegółowo unormowane z wszelkimi gwarancjami. Oczywiście w momencie interwencji Policja będzie dokonywać bardzo szczegółowych ustaleń, jeżeli chodzi o ustalenia faktyczne.

Jeżeli chodzi o postępowanie zażaleniowe, to w przypadku stwierdzenia przez sąd nielegalności lub bezzasadności zastosowania natychmiastowego nakazu policyjnego będzie obowiązek poinformowania bezpośredniego zwierzchnika służbowego tego funkcjonariusza, który ten środek zastosował. Jest również realne zabezpieczenie w postaci ewentualnego postępowania dyscyplinarnego. Osoby, które stosują przemoc, te związki, w których ta przemoc ma miejsce, są bardzo często dobrze znane Policji.

Będziemy wspólnie te kompetencje wzmacniać, przygotowując i przeprowadzając siłami Ministerstwa Sprawiedliwości szkolenia dla Policji, dla Żandarmerii Wojskowej, które będą dedykowane specjalnie w celu wdrożenia i podniesienia kompetencji Policji w zakresie stosowania natychmiastowego nakazu policyjnego. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie będzie dotyczyło zagrożeń dla wolności twórczości, powrotu cenzury i ręcznego sterowania przekazami w mediach publicznych, m.in. w kontekście wydarzeń w Programie 3 Polskiego Radia oraz milczenia pana ministra w sytuacji represji wobec ludzi kultury. To pytanie skierowane jest do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pytanie zada pani marszałek, przepraszam bardzo, pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Bardzo proszę. Panie Marszałku!

Zatem zacznę od pytania: Gdzie pan jest, panie ministrze? Ostatni raz pana widziałam na tej sali, jak pan bronił swojego kolegi ministra Szumowskiego. Czy może pan nie miał czasu przyjść tutaj dzisiaj, by odpowiedzieć na nasze pytania, bo pan szuka dowodów niewinności swojego kolegi ministra Szumowskiego? Kiedy chcemy rozmawiać o kulturze, pana nie ma. Kiedy chcemy rozmawiać o mediach, pana nie ma. Pan, zdaje mi się, w ogóle milczy, gdy chcemy rozmawiać z panem o kulturze. Pan milczał, gdy Policja atakowała słuchaczy oburzonych tym, co tam jest.

Nie wiem, czy pan nie wie, kto to był Kantor. Milczenie pana jest wymowne, bo pan nie znosi kultury i nie znosi ludzi kultury. Chcę tylko powiedzieć, że pan odpowiedzialności za to, co się dzieje, nie uniknie. Jeśli chodzi o media, proszę pana, to te wszystkie ustawy rodziły się pod pana ręką, te medialne ustawy potworkowe. To spod pana ręki wyszedł pana ówczesny zastępca Krzysztof Czabański, który dzisiaj jako szef Rady Mediów Narodowych dokonuje tych roszad personalnych. Pan będzie odpowiadał i za Jacka Kurskiego, i za Agnieszkę Kamińską. Pan będzie za nich odpowiadał, pan tej odpowiedzialności nie uniknie. Pan jest walnym zgromadzeniem tych spółek medialnych i pan działa na szkodę tych spółek. Dziękuję bardzo za zadanie pytania.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowne panie posłanki zadające pytania! Kilka uwag wstępnych. Pierwsza uwaga wstępna jest taka, skoro została poruszona kwestia tego, że premier Gliński jest walnym zgromadzeniem tej spółki, że ja też jestem walnym zgromadzeniem tej spółki, też mam uprawnienie do tego, żeby to walne zgromadzenie przeprowadzać. Dlatego informuję o uregulowaniach prawnych, jakie odnoszą się do walnego zgromadzenia. Kodeks spółek handlowych zakazuje wydawania jakichkolwiek wiążących poleceń radzie nadzorczej czy tez zarządowi. Zarząd jest autonomiczny i sam kształtuje politykę funkcjonowania spółki w każdym zakresie, program funkcjonowania spółki, to, jak spółka działa.

Dlatego minister kultury i dziedzictwa narodowego rzadko wypowiada się pozytywnie czy negatywnie o mediach, żeby nikt nie mógł pomyśleć, że w jakiś sposób chce wpływać na te media. Niemniej o sytuacji Trójki pan premier Gliński już kilka godzin po ujawnieniu tej informacji wypowiedział się w mediach.

To chyba jakaś prowokacja. Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i minister kultury nie musi się zgadzać ze wszystkimi decyzjami władz publicznego radia. I w tym miejscu chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeden ważny szczegół, że pan premier Gliński zareagował bardzo stanowczo na tę sprawę, która miała miejsce.

Chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że nie reagowaliście państwo tak ostro, kiedy na cmentarzu umawiano się z szefem jednej z redakcji, żeby wyrzucić dziennikarzy, którzy pisali nie w smak władzy.

Zdepenalizowaliśmy np. kwestie dotyczące autoryzacji, w tym momencie każdy dziennikarz może dosłownie przytoczyć każdą wypowiedź i nie potrzebuje do tego autoryzacji. Działamy na rzecz wolności słowa i na rzecz wolności artystycznej, czego przykładem jest szereg rozwiązań, które wprowadziliśmy m.in. w tarczy antykryzysowej, żeby pozwolić artystom przeżyć ten trudny czas. Ze wszystkimi szczegółami tej tarczy możecie państwo zapoznać się na stronie internetowej ministerstwa kultury. Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, to oczywiście służę. Dziękuję bardzo. To prawda, też bym chciała, żeby wicepremier Gliński odpowiedział na to pytanie, bo minister kultury powinien nie tylko stać na straży wolności kultury, ale także dbać o kondycję polskiej kultury, polskich artystów i twórców kultury. Odmrażamy gospodarkę, z czego jestem bardzo zadowolona, bardzo się z tego cieszę, ale dlaczego nie ma dialogu, dlaczego nie rozmawia się ze środowiskami. Słyszymy, że mają być otwarte kina, jestem jak najbardziej za, ale środowiska te martwią się, jak te kina mają być odmrażane. Nikt z nimi nie ustalił zasad, jak to ma funkcjonować. Przecież to jest bardzo ważne, bo to kiniarze będą potem ponosili odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków. Za kilka dni ma to się stać, a oni nadal nie wiedzą, jak to ma wyglądać. Druga sprawa. Tak, rozpisano program wsparcia dla artystów, którzy utracili możliwość [[Dzwonek]] funkcjonowania. Może trzeba uczciwie ludziom powiedzieć: kochani, nie ma pieniędzy, możemy wam pomagać tylko przez 3 miesiące - ale trzeba wyjść i to powiedzieć, bo niedomówienia są najbardziej szkodliwe. Proszę bardzo, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Otóż nieprawdą jest, że nie wprowadzamy w konsultacji z ludźmi kultury naszych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących odmrożenia gospodarki. Działa zespół antykryzysowy ds. kultury, który spotyka się średnio co tydzień. Biorą w nim udział w zasadzie przedstawiciele każdej branży. W związku z tym na podstawie także pracy tego zespołu przygotowaliśmy instrukcję, która została zaopiniowana albo jest w trakcie opiniowania przez GIS, Główny Inspektorat Sanitarny. To jest instrukcja, która została. Tak samo w przypadku teatrów.

Ostatnio tak szybko odpowiedzieliśmy na postulaty np. kinematografii, wprowadzając 1,5% opłaty od VOD, tak jak odpowiadamy na postulaty instytucji kultury, które działają w formie stowarzyszeń czy fundacji, dając im takie uprawnienia jak normalnym pracodawcom, żeby mogli korzystać z FGŚP, czy tworząc podobne rozwiązania dla innych typów organizacji, m.in. instytucji samorządowych, żeby częściowo partycypować w wynagrodzeniach dla pracowników tych instytucji, także z FGŚP. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze nie odchodzić, panie ministrze, bo ze sprostowaniem zgłosiła się pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Panie Ministrze! Bardzo się cieszę, że pan mówi o tej tarczy, bo już dwie interpelacje składałyśmy do pana ministra, żeby nam dokładnie powiedziano, co niby w tej tarczy takiego genialnego jest i ile już instytucji z tego skorzystało, ilu twórców. To tyle, jeśli chodzi o tarczę. Natomiast jeśli chodzi o cenzurę, panie ministrze, powiedziałam bardzo wyraźnie: ustawy medialne doprowadzają do takiej sytuacji, że Rada Mediów Narodowych, która się składa z trójki waszych partyjnych przyjaciół i kolegów, podejmuje takie, a nie inne decyzje kadrowe. Jeszcze raz powtarzam: cenzurowanie przez kierownictwo Polskiego Radia jest regułą, proszę zapytać dziennikarzy wyrzucanych na bruk, proszę zapytać Radę Programową. Z tego słynie pani prezes Agnieszka Kamińska, także jako szefowa Jedynki. Tak więc proszę mi nie opowiadać, że minister milczy, żeby nie cenzurować.

Panie Marszałku! Chciałem tego uniknąć, żeby nie przedłużać, nie zabierać czasu innym posłom na zadawanie pytań, ale skoro pani przewodnicząca zapytała, to dobrze. Kwotę 80 mln zł w programie „Kultura w sieci”, który składa się z dwóch części: stypendia i dotacje.

Wnioski są rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników odbyło się 8 maja. Pieniądze są właśnie wypłacane. 50 mln zł to jest wstępnie planowany budżet uruchomienia programu rekompensującego straty w kulturze po zakończeniu epidemii. Ponadto wystąpiliśmy o zerową stawkę VAT na książki drukowane, kontynuujemy prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, umożliwiliśmy dyrektorom instytucji kultury wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę zastępczą, przygotowujemy nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności, zmieniliśmy definicję dzieła filmowego, tak by umożliwić otrzymywanie dotacji z PISF również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych, zawiesiliśmy raportowanie danych przez kina, uelastyczniliśmy terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Ale to jeszcze nie koniec. Ale dlaczego na 3 miesiące, a nie na pół roku, jak miało być? Policzymy to na koniec epidemii.

Wyliczyliśmy, że ok. 1,7% wszystkich przedsiębiorców to są właśnie przedsiębiorcy w sektorze kultury. I mniej więcej odpowiednio taką kwotę lub nieco wyższą, oprócz tych kwot, które tutaj wymieniliśmy, oni otrzymają. Dziękuję bardzo. Panowie posłowie Jarosław Rzepa, Jan Łopata i Dariusz Klimczak z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 skierują pytania do ministra zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej polskich szpitali, zagrażającej utratą płynności finansowej. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Jarosław Rzepa. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od chwili, kiedy w Polsce ogłoszono stan zagrożenia, a potem epidemii, zamroziliśmy nie tylko gospodarkę, ale bardzo mocno ograniczyliśmy również to, co się dzieje w polskich szpitalach. Wynikało to oczywiście z przyjętych przez nas wszystkich zaleceń, ale spowodowało, szanowni państwo, to, że w wielu szpitalach z dnia na dzień ograniczono w bardzo drastyczny sposób ilość wykonywanych operacji, zabiegów, porad. W kwietniu znowelizowano wprawdzie rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, wskazując, że szpitale mogą dostać 1/12 ryczałtu - bo, jak państwo wiecie, szpitale w większości właśnie z tej formy korzystają, jeżeli chodzi o finansowanie - jako formę zaliczki, ale wszyscy, szanowni państwo, zdają sobie z tego sprawę, że dzisiaj mamy ogromne zagrożenie tym, że te zaliczki być może trzeba będzie zwracać. Chciałbym tutaj, panie ministrze, wyraźnie usłyszeć odpowiedź od pana, w jaki sposób zostanie naliczony ryczałt dla szpitali, które dzisiaj są szpitalami jednoimiennymi, oraz czy pozostałe jednostki służby zdrowia, w tym szczególnie szpitale powiatowe, które nie wykonywały ryczałtu za względu na ograniczenia, mogą liczyć na wypłatę naliczonych wcześniej kwot. Czy ministerstwo rozważa przedłużenie terminów rozliczania ryczałtów? Szanowni Państwo! Dzisiaj polskim szpitalom należy się pomoc. Chciałbym usłyszeć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia tę sprawę też zamierza rozpatrzeć. Odpowiedzi na pytanie udzieli pan Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ kondycja polskich szpitali to jest bardzo istotna sprawa i to, że, jak wszyscy wiemy, one funkcjonują teraz w zupełnie wyjątkowych okolicznościach, nie może zmienić faktu, że musimy o te jednostki zadbać i musimy zadbać o to, aby one utrzymały swój potencjał i były gotowe na to, by wrócić do normalnego funkcjonowania tak szybko, jak to będzie możliwe. Mówię: normalnego, ale ono na pewno będzie inne, ono będzie różne od tego, jakie znamy z lat ubiegłych, jeszcze przez kilka miesięcy, może nawet dłużej. Natomiast od samego początku Ministerstwo Zdrowia działało na rzecz tego, żeby zapewnić niezależne źródło finansowania dodatkowych świadczeń w ramach walki z COVID. Jeżeli przyjrzymy się finansom szpitali jednoimiennych, to widzimy jednoznacznie, że za marzec i kwiecień te szpitale otrzymały dodatkowo, w zależności od podmiotu, kilkadziesiąt, nawet do 80% więcej niż dostawały w standardowych miesiącach, ponieważ otrzymywały równocześnie ryczałt i środki przeznaczone na utrzymanie w ramach walki z COVID, środki, przypomnę, wypłacane niezależnie od standardowej zasady, która przewiduje, że płacimy za wykonane świadczenia, a nie za zgłaszaną gotowość. Tutaj zaproponowaliśmy 100 zł dziennie za każde łóżko gotowe i dodatkowo 200 zł za każde łóżko respiratorowe - za każdy dzień utrzymania takiej gotowości.

Na pewno będziemy chcieli to wydłużyć o pół roku, do połowy przyszłego roku, kiedy kończy się pierwszy cykl funkcjonowania sieci szpitali. Natomiast elastycznie podchodzimy do tej sprawy i wiemy, że może być taka sytuacja, że będzie to wymagało jeszcze dalszego wydłużenia. Jest absolutnie zrozumiałe, że teraz nie było możliwości pełnego wykonywania ryczałtów. Odpowiednie rozwiązania będą przygotowane zgodnie z naszymi deklaracjami. Jutro jest posiedzenie zespołu programowania prac rządu i mam nadzieję, że w ramach tego zespołu zostanie przyjęte odpowiednie rozwiązanie legislacyjne. Chciałbym też przypomnieć, że pomimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej, która dotyczy wszystkich instytucji publicznych, zgodnie z porozumieniem, które zawarliśmy ze związkiem szpitali, wypłacamy 5% zwyżki wyceny każdego punktu.

Tak że w ramach tarczy oczywiście zagwarantowaliśmy sobie to, że środki będą uzupełniane dotacją z budżetu państwa, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na pewno ze względu na ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze te wpływy ze składki będą mniejsze i naszą rolą będzie przygotowanie systemu na to, aby zapewnić dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania, tak jak to było w przypadku środków na COVID. Przypomnę, że te świadczenia i te polecenia były finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Jan Łopata. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Chciałbym dopytać właśnie w kwestii Narodowego Funduszu Zdrowia, wszak doskonale wiemy, że wpływ COVID-19 i tej epidemii na gospodarkę jest już jednoznaczny, spadek produkcji w kwietniu to dwadzieścia kilka procent, na pewno będzie wzrost bezrobocia, zapowiadane jest również zmniejszenie wynagrodzeń, a z tym wiążą się również plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra. Wysoka Izbo!

Szczególnie w specjalnościach zabiegowych - zakładam, że tu pan poseł się ze mną zgodzi - często kontrakty jednak przewidują, że wysokość wynagrodzenia jest w jakimś stopniu uzależniona od liczby wykonanych zabiegów, co oznacza, że także w trakcie epidemii te koszty się zmniejszyły. Przeprowadziliśmy zresztą takie badanie na grupie szpitali jednoimiennych i zauważyliśmy, że pomimo faktu, że skala działalności standardowej była tam istotnie ograniczona, pomimo tego, że były szpitale jednoimienne, które na całe szczęście nie musiały pracować w pełni swojego potencjału, te koszty istotnie nie wzrosły, wzrosły za to bardzo istotnie przychody, co paradoksalnie prowadziło do sytuacji, w której te 2 miesiące, kiedy funkcjonowały rozwiązania przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli marzec i kwiecień, to były miesiące z punktu widzenia finansów tych szpitali bardzo, bardzo korzystne. Tak że oczywiście absolutna zgoda z panem posłem, że musi być w ten sposób, że system, który przyjmiemy, będzie elastyczny. Jeżeli natomiast chodzi o szczegóły, jestem przekonany, że propozycja, którą przedstawimy, będzie do zaakceptowania, szczególnie, co niezwykle istotne, że mamy sytuację, w której już teraz te środki są przekazywane ze znacznie mniejszym opóźnieniem niż do tej pory.

I jestem przekonany, że stosowana będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie także skierowane jest do ministra zdrowia, a dotyczyć będzie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych dla personelu medycznego, podejmującego pracę w trudnym czasie epidemii COVID-19. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Urszula Rusecka. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Świat od paru miesięcy zmaga się z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Polska na tle większości krajów europejskich, i to również tych dużo, dużo bogatszych od naszego kraju, wypada bardzo dobrze. Nieźle radzimy sobie z tą epidemią.

Natomiast ze szczególnym szacunkiem obserwujemy prace personelu medycznego, który narażając swoje zdrowie, ratuje życie osób, które zachorowały. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, cały personel medyczny, szczególnie te osoby, które są na pierwszej linii frontu. Moje pytania są związane właśnie z pracą służb medycznych. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia wspiera pracowników służby zdrowia, a szczególnie tych, którzy są na pierwszej linii frontu? Czy rząd zamierza przeznaczyć dodatkowe środki finansowe dla personelu medycznego podejmującego pracę w trudnym czasie walki z epidemią? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra Janusza Cieszyńskiego. Wysoka Izbo! Pani Poseł! Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście to, co pani powiedziała, jest w 100% prawdą. Nie udałoby się nam tak skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, gdyby nie poświęcenie służb medycznych, gdyby nie to, że tak naprawdę na pierwszej linii frontu mamy tak zaangażowanych, tak chętnie poświęcających się tej pracy pracowników systemu ochrony zdrowia.

W związku z powyższym zostało także wydane polecenie ministra zdrowia wobec prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, aby sfinansować tym wszystkim osobom specjalne dodatki. Te dodatki wyniosą co najmniej 50% wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim miesiącu, nie więcej zaś niż 10 tys. zł, przy czym jeżeli pracownik utracił możliwość zarobkowania w innym miejscu, ta kwota będzie mogła być też powiększona do limitu 10 tys. zł, o 80% zarobków utraconych w innym miejscu pracy.

To także wyróżnia ich na tle innych sektorów.

Te środki zostały przeznaczone nie tylko na dodatkowe środki na świadczenia, na utrzymanie gotowości, na dodatki do wynagrodzeń, ale także na zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu, na zakup dodatkowego sprzętu i inne wydatki, które pozwoliły udzielać tych świadczeń w bardziej komfortowych warunkach i na wyższym poziomie. Warto wskazać, że jednym z fundamentów wykonywania zawodów medycznych jest właśnie to, aby móc je wykonywać w sposób zgodny z najbardziej aktualną wiedzą lekarską, czyli oznacza to dostęp do najnowocześniejszych terapii, do nowoczesnego sprzętu i tego, co jest w danej chwili potrzebne. Dziękuję bardzo. Jako druga pytanie dodatkowe zada pani poseł Bożena Borys-Szopa. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Interesowałoby mnie bardzo to, ile szpitali przedstawiło listę pracowników objętych tymi regulacjami rozporządzenia, o których pan przed chwileczką mówił. Czy ministerstwo ma możliwość weryfikacji tych danych? W jaki sposób to czyni? W sposób szczególny interesuje mnie moje województwo, województwo śląskie. Jaka to może być przypuszczalnie kwota, a przede wszystkim jaka może być liczba pracowników medycznych, którzy będą mogli z tego skorzystać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy pana ministra. Pani Poseł! Jeżeli chodzi o dokładne dane w rozbiciu na regiony, my jeszcze tymi danymi w pełni nie dysponujemy, ponieważ tutaj opieramy się o wnioski z podmiotów leczniczych. Te wnioski są rozpatrywane tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Wiem, że już pierwsze wnioski zostały rozpatrzone, natomiast one dotyczyły zazwyczaj mniejszych podmiotów, a co za tym idzie, zostały przekazane do tych podmiotów także odpowiednie środki finansowe.

Mówię o całej Polsce.

Natomiast aby on był kompletny, potrzebujemy danych ze wszystkich podmiotów. One zwyczajowo spływają za kolejny miesiąc do połowy miesiąca kolejnego.

Dziękuję bardzo. Panowie posłowie są gotowi do zadania pytania, tylko jeszcze musi być osoba, która na te pytania by odpowiedziała. W takim razie pytanie będzie do pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w sprawie niegospodarności i straty 1 mld zł spółek Skarbu Państwa powstałych przy budowie nietrafionej inwestycji w Elektrowni Ostrołęka. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Czesław Mroczek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po kilku latach działań rządu PiS doszło do katastrofy na rynku energetycznym w Polsce. Niektórzy odbiorcy płacą nawet o 70% więcej. Rząd wystraszony skutkami tej sytuacji postanowił wypłacać rekompensaty dla gospodarstw domowych. W 2019 r. na ten cel przeznaczono 9 mld zł. W bieżącym roku nie ma już tyle pieniędzy i rekompensaty nie obejmą wszystkich gospodarstw domowych. Dlaczego tak się dzieje? Rząd PiS stawia na węgiel, i to w dodatku na rosyjski węgiel. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło, zabiegając o poparcie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, złożyli deklaracje dotyczące budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka, chociaż już wtedy było wiadomo, że ta inwestycja jest nieopłacalna i że nie ma chętnych do finansowania tego zadania. Przymuszono do tego spółki energetyczne: Eneę i Energę. Klęska przyszła szybciej, niż można było przewidywać. Ale to nie jest cała strata związana z tą inwestycją, dlatego że były tam zaangażowane również pieniądze budżetowe.

To, co jest nieszczęściem dla naszego kraju, stało się rajem dla działaczy PiS-u, którzy obsiedli rady nadzorcze i zarządy spółek energetycznych związanych z Ostrołęką, żerując na mieniu publicznym. Proszę państwa, w wyniku tej polityki straconych zostało kilkanaście miliardów złotych (Dzwonek), które mogły być przeznaczone na projekty energetyczne służące zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza i obniżeniu kosztów. Dziękuję bardzo. Poprosimy o udzielenie odpowiedzi pana ministra Macieja Małeckiego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowa elektrownia w Ostrołęce będzie realizowana. Ta inwestycja jest niezbędna do zapewnienia stabilności systemu energetycznego w północno-wschodniej Polsce. Elektrownia w Ostrołęce jest potrzebna ze względu na stały rozwój regionu oraz coroczny wzrost zapotrzebowania na energię w Polsce, także w Polsce północno-wschodniej. Elektrownia w Ostrołęce mogłaby już powstać dawno temu, gdyby nie zaniechania rządu koalicji Platformy z PSL-em. Chodzi przede wszystkim o zaniechania w procesie dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. To była jedna z kluczowych przesłanek, która wpłynęła na podjęcie wcześniejszej decyzji o budowie bloku węglowego.

A czy faktycznym powodem zablokowania budowy w Ostrołęce nie był wasz deal z Rosją na budowę elektrowni jądrowej koło Kaliningradu?

A skąd się wzięły problemy, o których dzisiaj mówicie, kiedy tak troszczycie się o ceny prądu w Polsce? Czy czasem nie z decyzji rządu Donalda Tuska w 2008 r. Czy nie z decyzji z 2014 r. Ewy Kopacz i Rafała Trzaskowskiego, którzy zgodzili się na niekorzystne dla Polski zmiany w polityce klimatycznej Unii? Czy to nie Ewa Kopacz i Rafał Trzaskowski oddali Komisji Europejskiej decydujący wpływ na polską energetykę?

I to jest właśnie pokłosie tamtych decyzji Ewy Kopacz, Rafała Trzaskowskiego i wcześniej Donalda Tuska.

To świadczy o poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za kluczowe inwestycje w Polsce i takie poczucie obowiązku i odpowiedzialności ma rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że te inwestycje muszą też służyć transformacji energetycznej. Orlen, który kupił 80% akcji Grupy Energa, poinformował dokładnie, że planowana jest konwersja tej elektrowni na gaz. Należy podkreślić, że zmiana technologii jest możliwa również dzięki konsekwentnej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. To rozbudowa terminala gazowego w Świnoujściu im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i budowa gazociągu Baltic Pipe pozwolą bezpiecznie inwestować w nowe instalacje gazowe. Budowa bloku w Ostrołęce ma także duże znaczenie dla niezawodności i stabilności połączenia międzysystemowego między Polską a Litwą. My pomagamy Litwie, pomagamy krajom bałtyckim w uniezależnieniu się od rosyjskiego systemu elektroenergetycznego. To wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości politykę solidarności energetycznej w Europie i to powinno być przykładem dla wielu państw unijnych. A wobec trendów, jakie panują w Komisji Europejskiej, długookresowo technologia gazowa jest optymalna kosztowo, ekonomicznie i Ostrołęka wpisuje się w szerszy trend transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego zmierzającego do wykorzystania nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Krzysztof Gadowski.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Udowodnił pan, panie ministrze, że pan śmieje się z tego, co pan mówi, czyli potwierdza pan tezę, którą mój kolega przed chwilą postawił, że rzeczywiście pieniądze, ten 1 mld czy 1,5 mld zł, zostały ewidentnie zmarnowane przy realizacji tej inwestycji. W 2018 r. rozpoczęliście inwestycję. Miała kosztować po przetargu 5 mld.

Czy dołożył staranności przy realizacji tej inwestycji, przy podjęciu tej decyzji w 2018 r., że będziecie budować tę elektrownię? Kto personalnie odpowiada za ten chaos, za te zmarnowane miliardy złotych, które dzisiaj wychodzą na jaw? Dziękuję bardzo. Prosimy pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dużo oskarżeń padło ze strony posłów opozycji, ale było jak zwykle: populizm i brak konkretów.

Zbudowana zostanie w oparciu o technologię gazową. Dlaczego? Dlatego że radykalnie zmieniło się otoczenie makroekonomiczne. i Komisja Europejska, również dzięki waszej bierności, waszej zgodzie, konkretnie Ewy Kopacz i Rafała Trzaskowskiego w 2014 r., mogła zradykalizować podejście do polityki klimatycznej. Ta polityka klimatyczna nie zawsze przystaje do realiów życia gospodarczego, na co państwo też kiwaliście głowami, kiedy podawałem przykłady krajów azjatyckich, gdzie nie ma takich radykalnych rozwiązań. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie się ścigał w polityce klimatycznej kosztem Polaków. Podejmujemy wyzwanie, podjęliśmy wyzwanie, jakim jest transformacja energetyczna, ale robimy to w sposób bezpieczny dla polskiej gospodarki, w sposób bezpieczny dla konkurencyjności polskich firm i w sposób bezpieczny dla budżetów polskich rodzin.

Podaję przykładowo blok, który może być budowany. Projekt jest korzystny także dla regionu Ostrołęki. Pozwoli na przyspieszenie rozwoju, da impuls do ożywienia gospodarczego w północno-wschodniej Polsce. Szczególnie dzisiaj, kiedy wychodzimy z pandemii i odmrażamy gospodarkę, to jest bardzo ważne. W czasie odmrażania gospodarki i powrotu na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego, którego Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość zazdrościło wiele krajów Europy, duża będzie rola spółek Skarbu Państwa. Nie oczekuję od posłów obecnej opozycji, że państwo podzielicie nasze stanowisko, bo mieliście na to zupełnie inne spojrzenie. Wy chcieliście spółki prywatyzować, wyprzedawać, my chcemy, żeby spółki rozwijały się i były lokomotywami polskiej gospodarki. Pan minister udaje, że nie wie, kto pytanie zadawał, ale to jest dobry moment, żeby w ramach sprostowania odnieść się do tego, o czym mówił pan minister.

W 2015 r. rząd Platformy i PSL-u powiedział, że tam powinna powstać elektrownia gazowa. Dzisiaj, po kilku latach, wracacie do pomysłu bloku gazowego i mówicie, że nic się nie stało. Stało się, kochani. Pytam o niegospodarność.

Widzę, że pan marszałek kolegom z opozycji musi rzucić koło ratunkowe w postaci dodatkowej możliwości wypowiedzi.

To jest dobra okazja, żeby to jeszcze raz wybrzmiało na tej sali. To jest sytuacja, która wpływa na zmianę otoczenia makroekonomicznego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zachowuje się w sposób odpowiedzialny, bo elektrownia w Ostrołęce jest potrzebna.

To rząd Platformy i PSL-u pozwolił na to, żeby polityka klimatyczna miała bardzo mocny wpływ na polską gospodarkę. Rok 2014 - Ewa Kopacz, Rafał Trzaskowski, który zapowiadał wtedy, że ceny prądu nie pójdą w górę.

Dziękuję bardzo panu ministrowi. Kolejne pytanie będzie zadane w sprawie wspierania przez rząd kół gospodyń wiejskich. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pani minister Anna Gembicka. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W dniu 19 maja br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa przewiduje kontynuację udzielania pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich zainicjowanej już w 2018 r. przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Czy mogłabym panią minister poprosić o przybliżenie Wysokiej Izbie warunków i zasad udzielania wsparcia finansowego kołom gospodyń wiejskich i wyjaśnienie, jaki będzie miało to wpływ na rozwój społeczności lokalnej? Wiemy, że te wspaniałe kobiety, które tworzą te małe ojczyzny, dbają o kulturę i szerzenie tradycji. Naprawdę zasługują na to, aby je wspierać i im pomagać, aby przede wszystkim to, co piękne w naszej tradycji, promować nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Pani minister, bardzo proszę o udzielenie informacji. Dziękuję bardzo. Proszę panią minister Annę Gembicką o udzielenie informacji. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło gospodyń wiejskich to organizacja rozwijająca się bardzo prężnie, jednocześnie z piękną długoletnią tradycją. Od 2 lat mamy do czynienia z prawdziwym renesansem tej formy działalności, o czym świadczy bardzo dynamiczna, barwna działalność kobiet gospodarnych i wyjątkowych.

W aż 96% powiatów w Polsce działa co najmniej jedno koło gospodyń wiejskich. W 2018 r. zarejestrowało się 5048 kół gospodyń wiejskich, w 2019 r. zarejestrowanych było już 8828 kół, a według stanu na 11 maja tego roku mamy ich już 9113. Liczba członków kół to aż 239 tys. osób.

Co ważne, te wszystkie środki będą przeznaczone właśnie na wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich. Wiemy, że te środki będą bardzo dobrze wydane, bo ich działalność jest tak naprawdę działalnością rozwojową na rzecz polskiej wsi. Pomoc finansowa będzie przyznawana w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek zarejestrowanego koła gospodyń wiejskich. Wnioski będzie można składać do kierowników biur powiatowych agencji. Będzie to można zrobić na formularzu udostępnionym przez agencję. Podobnie jak w poprzednich latach ta pomoc finansowa będzie mogła zostać przeznaczona na działalność statutową. To jest bardzo szeroki katalog działań. Każdy zarejestrowane koło, które złoży wniosek, będzie mogło otrzymać 3, 4 lub 5 tys. zł, w zależności od liczebności. Ustawa będzie miała korzystny wpływ na rozwój lokalnych inicjatyw społecznych, na rozwój wsi zarówno w tej warstwie gospodarczej, bo zawsze powtarzam, że koła gospodyń to są takie małe inkubatory przedsiębiorczości, ale z drugiej strony na tę warstwę kulturalną, na zachowanie naszego dziedzictwa i tradycji. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za działanie tej grupy społecznej, która jest bardzo aktywna, która tworzy tradycję w Polsce. Tak jak zostało powiedziane, Polska jest silna rodziną i tradycją. bardzo podziękować, bo to jest wielka sprawa.

Myślę, że to by było bardzo zasadne. Po to aby wszystko było w porządku, jasne i klarowne, bo rozliczenie jest bardzo proste. Pięknie dziękuję. Dziękujemy bardzo, pani poseł, za zadanie dodatkowego pytania. Prosimy panią minister o udzielenie odpowiedzi.

Tak jak powiedziałam wcześniej, kwestia wypłacania będzie w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chcemy przystąpić do tego wypłacania jak najszybciej, bo wiemy, że koła oczekują na te środki, tym bardziej że w okresie letnim zazwyczaj odbywa się dużo projektów, dużo inicjatyw, na które często te środki są wydawane. Co ważne, przy okazji składania sprawozdań czy wnioskowania o środki koła mogą liczyć na pomoc specjalnie wyznaczonych do tego pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc nie zostawiamy ich samych. Rozmawiamy, jesteśmy w kontakcie z kołami gospodyń. Wiemy, że cały czas jest potrzeba organizacji różnych szkoleń, różnych działań podnoszących kompetencje. W zeszłym roku udało się nam zorganizować ponad 40 takich spotkań, brali udział w tych spotkaniach też przedstawiciele urzędów skarbowych, którzy odpowiadali na pytania, które się pojawiały.

Mam nadzieję, że będzie możliwe ich przeprowadzenie w formie stacjonarnej. Jeżeli nie, to będziemy chcieli zorganizować webinary, tak żeby w sposób zdalny móc się połączyć, móc wziąć udział w takim szkoleniu. Wiemy, że jest cały czas potrzeba podnoszenia kompetencji właśnie w zakresie działalności organizacji pozarządowych, w zakresie działalności kół gospodyń wiejskich. Takie działania cały czas prowadzimy.

Przygotowujemy też nową odsłonę strony internetowej. Chcemy, żeby wszystkie informacje, które są potrzebne do funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, były zawarte właśnie w tym miejscu, żeby jak najlepiej odpowiadać na te pytania. Chcemy na bieżąco odpowiadać na te potrzeby, które są nam zgłaszane. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie skierowane będzie do ministra funduszy i polityki regionalnej. Zada je pan poseł Waldemar Andzel, a odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pan minister Grzegorz Puda. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki. Fundusz ten ma wspierać transformację regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla.

Mam pytania do pana ministra: Ile ze wspomnianego 0,5 mln euro na przygotowanie planu sprawiedliwej transformacji otrzyma województwo śląskie? Jakie podmioty będą odpowiedzialne za przygotowanie planu sprawiedliwej transformacji dla wskazanych województw? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana ministra Grzegorza Pudę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Informację o otrzymaniu wsparcia z programu wsparcia reform strukturalnych dostaliśmy 11 maja. Wartość wsparcia to 500 tys. euro, czyli, przeliczając na złotówki, ok. 2 mln zł. Celem tego wsparcia jest wzmocnienie ogólnej zdolności państw członkowskich w zakresie przygotowania oraz wdrożenia instytucjonalnych, strukturalnych i administracyjnych reform sprzyjających wzrostowi. Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że to wsparcie ma charakter zewnętrznego doradztwa eksperckiego, a co się z tym wiąże, wsparcie będą realizowali eksperci wyłonieni w przetargu przez Komisję Europejską. Trzeba także w tym punkcie podkreślić, że wciąż nie zostały zakończone rozmowy z Komisją Europejską odnośnie do zakresu wsparcia.

Tak jak wcześniej pan poseł zauważył, są to podregiony: na Śląsku - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski i sosnowiecki, w Wielkopolsce - podregion koniński, a na Dolnym Śląsku - podregion wałbrzyski. Jednakże stoimy na stanowisku, że wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno zostać skierowane także do województw: lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego, które również odczuwają skutki procesu transformacji. Wiadomo, o to walczymy. W dniu 20 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wstępne rozmowy dotyczyły możliwości ukierunkowania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce. I odnośnie do pytania drugiego: jak wspomniano, wsparcie doradcze będzie realizowane przez ekspertów wybranych w związku z zamówieniem publicznym realizowanym przez Komisję Europejską.

Mamy nadzieję, że prace grupy roboczej przy naszym ministerstwie będą pomocne w wypracowaniu takiej ścieżki wsparcia. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada także pan poseł Waldemar Andzel. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, za odpowiedź, za działania, które podejmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w tej dziedzinie.

Dziękuję bardzo. Prosimy pana ministra. Wysoka Izbo! Otóż negocjacje w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tak naprawdę są dopiero na mocno początkowym etapie. Po przedstawieniu propozycji przez Komisję Europejską w dniu 14 stycznia Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wypracowują swoje stanowiska. Co za tym idzie, prace w Radzie Unii Europejskiej, w które bezpośrednio angażuje się nasze ministerstwo, są mniej więcej na końcowym etapie, ale oczekujemy na przedstawienie przez prezydencję chorwacką trzeciej, i liczymy na to, że już ostatniej, propozycji kompromisu. Kolejnym etapem tych prac będą negocjacje trójstronne pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie skierowane jest do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a dotyczy pomocy finansowej oraz materiałowej, jaką rząd przeznaczył dla DPS-ów będących jednostkami, których organami prowadzącymi są samorządy. Pytanie skierowali państwo posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Joanna Borowiak i Mariusz Trepka. Jako pierwsza zada pytanie pani poseł Joanna Borowiak. Wysoki Sejmie! Pani Minister! Osoby starsze stanowią grupę szczególnie narażoną na zachorowanie, a także na skutki zakażenia koronawirusem.

One są prowadzone przez samorządy. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pensjonariuszy rząd jednak nie pozostawił DPS-ów bez pomocy.

Aktualnie sytuacja epidemiczna w Polsce poprawia się, stabilizuje, jednak potrzebne jest ciągłe jej monitorowanie.

Kierując się troską o seniorów, o ich bezpieczeństwo, uprzejmie proszę panią minister o odpowiedź na pytanie: Jaki był zakres pomocy finansowej, a także pomocy materiałowej, udzielonej dotąd przez rząd dla pensjonariuszy oraz pracowników domów pomocy społecznej w związku z epidemią koronawirusa? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli pani minister Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Szanowni Państwo! Tak, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w swoim obszarze działania domy pomocy społecznej, nad którymi nadzór sprawuje wojewoda i które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli najczęściej powiaty albo, na zlecenie powiatów, różne organizacje pozarządowe. Szanowni Państwo! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma w obszarze działania domy pomocy społecznej, nie mylić z zakładami opieki leczniczej. Pani poseł powiedziała, że mamy 824 domy pomocy społecznej - wszystko się zgadza - i w tych domach pomocy społecznej jest 81 tys. mieszkańców.

Szanowni Państwo! Pani poseł pytała o pomoc, jaką rząd premiera Mateusza Morawieckiego i ministerstwo, które mam zaszczyt reprezentować, skierowały do domów pomocy społecznej. Otóż skierowaliśmy 20 mln zł w gotówce z rezerwy celowej budżetu państwa jako działanie ponadplanowane, i to jest decyzja z 3 kwietnia 2020 r., na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności.

Tutaj mamy zaplanowane 380 mln zł do przekazania poprzez ROPS-y do domów pomocy społecznej i to w tej chwili się dzieje. Bardzo nam zależało od początku, wiedzieliśmy, że konieczne jest wsparcie dodatkowe, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej.

Sytuacja w tym czasie jest monitorowana.

Nie dawniej niż przedwczoraj pan minister tu niedawno obecny, minister Cieszyński, zaakceptował trzeci wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o środki, które poprzez Agencję Rezerw Materiałowych zostaną skierowane do domów pomocy społecznej. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zada pani poseł Lidia Burzyńska. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję pani minister za przedstawienie, w jaki sposób rząd premiera Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy, zarówno finansowo, jak i materiałowo, mimo że to jest ich zadanie, ale senior jest rzeczą, jest wartością dla rządu, dla społeczeństwa, dla ministerstwa bardzo istotną. Pani minister, pani to powiedziała w swoim wystąpieniu, niemniej jednak proszę o wyartykułowanie tego jeszcze raz, ponieważ DPS-y są to miejsca, gdzie zarażenie jest najbardziej potencjalne, chociażby z racji wieku pensjonariuszy, bo są to osoby starsze i - jeszcze jedno - ponieważ chorują, czyli żyją z chorobami współistniejącymi. Pani minister, czy sytuacja zdrowotna w domach opieki społecznej jest w dalszym ciągu monitorowana i czy przewidziane jest (Dzwonek) dalsze wsparcie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią minister.

W swoich raportach dyrektorzy wydziałów polityki społecznej przekazują aktualne i szczegółowe informacje.

Służby wojewodów są w stałym kontakcie z domami pomocy społecznej, z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadziliśmy tam bardzo dużo różnych rekomendacji, które zostały wdrożone przez domy pomocy społecznej, i naprawdę. Tam są również dzieci.

Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia w tym zakresie.

Chciałoby się, żeby nie było w ogóle zakażeń, to jest oczywiste, natomiast one są i tam, gdzie one występują, staramy się w miarę możliwości pomagać. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie będzie także skierowane do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, a dotyczyć będzie środków pieniężnych, jakie już zostały wypłacone przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Joanna Lichocka. Panie Marszałku! Chciałabym otrzymać dość szczegółowe informacje na temat skali pomocy, która jest kierowana do przedsiębiorców małych, dużych, średnich, tych, którzy w sytuacji ogromnego jednak kryzysu ratują miejsca pracy i otrzymują pomoc od rządu.

Natomiast ja mam wrażenie, że jest mało informacji na temat konkretów, tzn. chciałabym, żeby państwo publikowali albo chociaż tutaj przedstawili informacje o największych przelewach, jakie poszły właśnie na ratowanie miejsc pracy, o konkretnych firmach, bo ci ludzie są.

I bardzo bym była wdzięczna, pani minister, gdyby przynajmniej kilka przykładów, może największych firm albo największych przelewów, które zostały przekazane właśnie na ratowanie miejsc pracy, zostało tutaj przedstawionych. I przy tej okazji chciałabym też dowiedzieć się na temat skuteczności współpracy z samorządami. Wiemy oczywiście, że są samorządy, są powiatowe urzędy pracy, które niestety nie pracują tak, jak byśmy sobie tego życzyli, jak przedsiębiorcy by sobie tego życzyli. Myślę oczywiście o Warszawie, gdzie skuteczność rozpatrzenia wniosków jest na poziomie kilkunastu procent i to się nie zmienia. Tam rozpatrzenie wniosków jest na poziomie 90%. To nie jest daleko od Warszawy, natomiast tam pomoc już dotarła, bo nie ma obstrukcji albo nie ma nieudolności Platformy Obywatelskiej i pana Trzaskowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na zadane pytanie udzieli pani minister Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Za nami już prawie 2 miesiące działania tarczy antykryzysowej, tarczy, która w pierwszej kolejności chroni miejsca pracy, wspiera przedsiębiorców, ale także samozatrudnionych, a dla wielu firm jest może jedyną szansą na przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że poszczególne instrumenty tarczy antykryzysowej stanowią realną pomoc w tym szczególnie trudnym dla gospodarki czasie. Epidemia koronawirusa i jej negatywne skutki odczuwane są niemal w każdej dziedzinie życia. Tarcza antykryzysowa, szanowni państwo, działa, a przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z instrumentów w niej zawartych. W tarczy jest szereg instrumentów. Tarczę realizują zarówno wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, tarczę doskonale realizuje Polski Fundusz Rozwoju. Szanowni państwo, to ogromne pieniądze przeznaczone na ochronę istniejących miejsc pracy. Myślę, że widać to również w statystykach rynku pracy, gdzie, owszem, przybywa osób zarejestrowanych jako bezrobotne, natomiast nie przybywa ich tak lawinowo i skokowo, jak mogłoby przybywać w momencie, kiedy nie byłoby tych instrumentów.

Jednym z elementów tarczy jest umarzalna, niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. 3 miesiące przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od momentu otrzymania pożyczki i taka pożyczka ulega umorzeniu.

Większość urzędów, szanowni państwo, tak jak pani poseł powiedziała, doskonale radzi sobie z realizacją i obsługą instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej, bo rząd, szanowni państwo, pomyślał o wszystkich działaniach w ramach tarczy antykryzysowej, nie tylko o tym, aby przekazać środki na realizację tego tak ważnego dla nas wszystkich zadania, ale również o tym, żeby zabezpieczyć koszty związane z obsługą tego zadania. To dla nas wszystkich, szanowni państwo, było kluczowe: żeby nie zostawić podmiotów, które realizują to zadanie, bez dodatkowego wsparcia. Kto inny miałby zrealizować to zadanie jak nie urzędy pracy, które na co dzień zajmują się wsparciem przedsiębiorców i pomocą im, a z drugiej strony zajmują się pomocą osobom, które w tej trudnej sytuacji utraciły pracę, czyli pełnią rolę tego pośrednika.

Niestety, tak jak pani poseł powiedziała, Warszawa nie do końca potrafi sobie poradzić z realizacją tego zadania. Szanowni państwo, o tarczy nie mówimy od dnia dzisiejszego, o tarczy mówimy od marca. Już w marcu wiadomo było, że będą przygotowywane programy, których realizatorami będą samorządy, te samorządy, które są blisko mieszkańców. Szanowni państwo, przekazaliśmy środki finansowe na realizację tego zadania, przekazaliśmy środki na obsługę tego zadania, stworzyliśmy szybkie instrumenty informatyczne dotyczące realizacji tego zadania. Jesteśmy w stałym kontakcie z urzędami pracy, mamy wideokonferencje, nie pozostawiliśmy tych instytucji samych. W Warszawie stopień rozpatrzenia wniosków, szanowni państwo, to zaledwie 16%. Pani Poseł! Tych wniosków nie tylko w Warszawie jest dużo. Ja powiem, jak świetnie radzi sobie Łódź.

Dlatego dziwi mnie, że tu, w stolicy, jest takie podejście do przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tego wsparcia.

Dziękuję bardzo, pani minister, za udzielenie odpowiedzi. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Barbara Bartuś. Dziękuję. Wysoka Izbo! Pani Minister! Rozpocznę od podziękowań za to wszystko, co się dzieje.

Przy tej okazji chciałabym też podziękować wszystkim urzędnikom, zarówno samorządowym, jak i pracownikom urzędów pracy, ale przede wszystkim urzędnikom, pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownikom tych wszystkich jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju, który tak często jest krytykowany, za ten ogrom pracy, który wykonują, za tę pracę popołudniami, wieczorami, za tę pracę sobotnio-niedzielną, za to, że przedsiębiorcy otrzymują tę pomoc, że o tę pomoc mogą się zwracać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Za to wszystkim bardzo dziękuję. Myślę, że to jest podziękowanie od nas wszystkich. Ale też, pani minister, byłabym wdzięczna, gdyby pani mogła - są jeszcze (Dzwonek) 3 minuty - powiedzieć więcej właśnie o tych świadczeniach, w sprawie których przedsiębiorcy mogą się zwracać, o świadczeniach postojowych, o dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników, o tej pomocy, która jest realna i z której można skorzystać. Dziękuję bardzo. Prosimy panią minister o udzielenie odpowiedzi. O tych instrumentach można mówić naprawdę wiele, wiele dobrych rzeczy, bo tak jak powiedziałam, one po prostu działają, a zainteresowanie przedsiębiorców tymi instrumentami jest bardzo duże. Tutaj pani poseł powiedziała: A po co cztery tarcze? Szanowni państwo, my rozmawiamy z przedsiębiorcami, na bieżąco monitorujemy sytuację i kolejna tarcza to jest odpowiedź na oczekiwania kolejnej branży i kolejnej grupy przedsiębiorców. w zakresie ochrony miejsc pracy. I to jest dla nas najważniejsze. Realizujemy zadania również, tak jak powiedziałam, przez wojewódzkie urzędy pracy. To są zadania w zakresie ochrony miejsc pracy.

Taki wniosek składa i otrzymuje wsparcie na każdego pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Można również składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie postojowe lub o umorzenie składek ZUS-owskich. Szanowni Państwo! Informacje na temat tarczy antykryzysowej są szeroko, myślę, upowszechniane w wielu miejscach. Mogę jeszcze powiedzieć, że w urzędach pracy jest realizowane świetne rozwiązanie wspierające organizacje pozarządowe, wspierające samozatrudnionych, mikro-, małe, średnie firmy. To jest pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak powiedziałam, szanowni państwo, obserwujemy, monitorujemy sytuację na rynku pracy, a myślę, że reakcją jest to, co dzieje się na rynku pracy, czyli nie zaobserwowaliśmy lawinowego, skokowego przyrostu zatrudnienia.

Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie skierowane jest do ministra infrastruktury, a dotyczy rządowych rozwiązań dla branży transportowej w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Paulina Matysiak. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać o rządowe rozwiązania dla branży transportowej w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami.

Zgodnie z zapisami tarczy 3.0 do przewoźników kolejowych będzie mogło trafić wsparcie na pokrycie braku wpływów ze sprzedaży biletów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i rekompensata ulg ustawowych na poziomie takim samym jak w 2019 r., ale nie uchwalono przepisów chroniących upadający rynek przewozów autobusowych. Takie przepisy wprowadził Senat przez dodanie formuły „transport drogowy gminny i powiatowy” wszędzie tam, gdzie był przywoływany transport kolejowy. Dzięki temu przewoźnicy autobusowi mogliby otrzymać takie wsparcie i rekompensaty za przejazdy ulgowe jak przewoźnicy kolejowi. Te poprawki odrzucono bez dyskusji.

Pracownicy nie wiedzą, kiedy i w jakiej wysokości otrzymają zaległe wypłaty. W pozytywnym świetle w poprzednim pytaniu został przywołany mój okręg wyborczy, sieradzki. Jeśli chodzi o transport, to niestety nie jest tak różowo, chodzi chociażby o wspominany przeze mnie PKS Zduńska Wola, który zawiesił szereg regionalnych połączeń, czy miejskie zakłady komunikacji w poszczególnych miastach: Kutnie, Zgierzu, Pabianicach, Sieradzu, które nie łapią się na wsparcie z żadnej tarczy. Nasuwa się kilka pytań. Co państwo zamierzają zrobić, żeby pomóc przewoźnikom? Co powiecie maturzystom, którzy nie będą mieli czym dojechać na egzaminy, które będą już niebawem? Co mają zrobić osoby, które chcą dojechać do pracy, ale nie mają czym? Proszę o konkrety, o fakty, liczby, terminy wprowadzenia proponowanych przez rząd rozwiązań. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Bardzo proszę, pan minister. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Faktycznie epidemia koronawirusa dotknęła Polskę nie tylko w sensie zdrowotnym, ale również w sensie gospodarczym. Branża transportu autobusowego i kolejowego też bardzo mocno to odczuwa. Zawieszone lekcje w szkołach, zawieszone zajęcia na studiach, praca zdalna, wiele osób, które pozostały ze swoimi dziećmi w ramach opieki nad nimi - to wszystko spowodowało, że Polacy w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie przemieszczali się tak gremialnie, nie podróżowali tak codziennie i to faktycznie bardzo negatywnie wpłynęło na transport zbiorowy, i ten autobusowy, i ten kolejowy. Poszczególne elementy tarczy antykryzysowej, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich 2 miesięcy, wychodzą naprzeciwko wielu postulatom, które padały zarówno ze środowiska kolejowego, jak i środowiska przewozów autobusowych. Oczywiście te dwie dziedziny transportu różnią się od siebie nie tylko formą przemieszczania się, ale także formą organizacyjną. Podmiotów, które zajmują się transportem kolejowym, w całej Polsce jest zdecydowanie mniej. Są to podmioty albo państwowe, albo samorządowe. Natomiast transport autobusowy miał to do siebie, że został pozostawiony na wolnym rynku. Transport autobusowy był prowadzony głównie przez podmioty komercyjne, głównie przez firmy, które na tym zarabiały. Kiedy byli klienci, kiedy byli pasażerowie, wtedy był zarobek, ale kiedy ze względu na sytuację zdrowotną czy epidemiczną tych pasażerów było zdecydowanie mniej - i tu potwierdzam te wartości, które przywołała pani poseł, czyli od 80 do 90% mniej - wtedy faktycznie zaczęły się problemy tych firm przewozowych. One oczywiście mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej, z tych instrumentów wsparcia, które przed chwileczką podała pani minister Alina Nowak. To naprawdę procedura nieskomplikowana, nietrudna, a pozwala na to, aby uzyskać wsparcie finansowe, na to, aby nie zwalniać pracowników, i na to, aby ten trudny okres przeżyć. Pani poseł, pozwolę sobie na te szczegółowe pytania odpowiedzieć na piśmie. Mamy tu przygotowany cały pakiet informacji. To oznacza, że faktycznie transport zbiorowy jest państwu bardzo bliski. Natomiast opowiem o jednym narzędziu, które w tej chwili jest realizowane.

W tej chwili wojewodowie we wszystkich województwach - i tutaj, szanowni państwo, bardzo proszę o uwagę, o zainteresowanie się tym tematem i przekazywanie tej informacji do samorządów - prowadzą nabór na utworzenie nowych linii użyteczności publicznej. W mojej ocenie, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury, wielu przewoźników komercyjnych, którzy mają w tej chwili problemy, powinno na podstawie porozumień z samorządami zostać zaangażowanych do tego, aby być operatorami na tych liniach użyteczności publicznej, a tym samym móc od momentu świadczenia usług otrzymywać maksymalnie do 3 zł za wozokilometr na wszystkich nierentownych liniach. 3 zł, szanowni państwo, to naprawdę bardzo dużo. Naprawdę to wsparcie rządowe, wsparcie, które zostało zawarte w tej trzeciej odsłonie tarczy antykryzysowej, jest tutaj bardzo istotne. Zachęcamy wszystkich przewoźników i samorządowców do tego, aby aplikowali, aby składali wnioski. Środków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest naprawdę bardzo dużo.

Są one dostępne dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które w trakcie roku będą chciały z nich skorzystać. Zachęcamy do tego, bo to naprawdę pozwoli nie tylko prowadzić ofertę transportową w danych gminach, powiatach czy regionach naszego kraju, ale również pozwoli na to, aby podmioty przewozowe, podmioty prywatne mogły w tym czasie w miarę normalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o marzec, stan epidemii został ogłoszony, mówię z głowy, mniej więcej w połowie tego miesiąca, czyli na początku marca transport funkcjonował w miarę normalnie. Ci, którzy mieli kupić bilety miesięczne, i to zarówno w przewozach autobusowych, jak i w przewozach kolejowych, zrobili to. Tak że wpływy do spółek przewozowych z tego tytułu w marcu były niezachwiane. Dlatego te problemy w tym miesiącu jeszcze nie były tak widoczne jak w kwietniu czy w maju, w których to miesiącach, tak jak powiedziałem podczas swojego pierwszego wystąpienia, faktycznie przewozy kolejowe i autobusowe były albo zawieszane, albo mocno ograniczane.

Najprostszy przykład: zamiast czterech wagonów jechał jeden, bo wiadomo że na tylu pasażerów nie było takiej potrzeby.

Natomiast mamy informację, że regionalni przewoźnicy również starali się to zrobić, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Jeszcze raz powtarzam, że wszystkie działania, które zostały skierowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, pana ministra Andrzeja Adamczyka, zostaną państwu, paniom i panom posłom, przedstawione w formie pisemnej. Mam nadzieję, że one rozwieją wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o intencje naszych działań. Dziękuję bardzo. Pytanie to kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Barbarę Bartuś. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Przez ostatnie 4,5 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestował bardzo dużo w budowę infrastruktury. Czasami narzekamy na utrudnienia, które wynikają z budowy dróg, na ruch wahadłowy, ale przecież nie od razu Kraków zbudowano. Sieci dróg szybkiego ruchu czy zmodernizowane linie kolejowe to podstawa sprawnego i spójnego transportu ludzi i rzeczy. Bez tego typu infrastruktury trudno byłoby mówić o państwie nowoczesnym. Nasz rząd wykorzystuje inwestowanie w infrastrukturę jako walkę z wykluczeniem komunikacyjnym różnych regionów oraz jako ważny element rozwoju, i to nie tylko rozwoju komunikacji w naszym kraju, ale też rozwoju gospodarki. Epidemia koronawirusa nie zatrzymała w naszym kraju prac infrastrukturalnych, drogowych czy kolejowych, przynajmniej tych, za które odpowiada rząd. Niestety, w samorządach bywa to różnie. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów zapewnia utrzymanie stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. I tak realizowany jest „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023”, którego celem jest budowa dróg szybkiego ruchu i stworzenie spójnej sieci transportowej Polski. Limit programu dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości został zwiększony i obecnie wynosi 142,5 mld zł. Program budowy 100 obwodnic, czyli budowa obejść miast średnich i mniejszych, jest kluczowym elementem poprawy przepustowości oraz jakości życia mieszkańców. Stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program ma za zadanie stworzenie obwodnic w 100 miejscowościach.

Mam nadzieję, że w wystąpieniu pan minister powie coś więcej na temat listy rezerwowych, na temat tych 53 miast, które są na liście rezerwowych.

Program zakłada przebudowę 9 tys. linii kolejowych. Poprzez realizację tego programu nastąpić ma poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a także między innymi ważnymi ośrodkami gospodarczymi. Dodatkowo zostaną zapewnione połączenia kolejowe z portami morskimi w celu integracji różnych gałęzi transportu.

Program „Kolej+”, przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2019 r. - jego głównym celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej, z miastami wojewódzkimi, oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów przy wsparciu ze środków publicznych. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu wynosi ponad 6,5 mld zł.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom blisko 80% połączeń uruchamianych przez przewoźnika ma być zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru, a co najmniej 77% pociągów ma mieć bezprzewodowy Internet.

Zbudowane zostaną nowe przystanki kolejowe, odbudowane te, które od lat nie istnieją. Będzie to jeden z elementów odmrażania polskiej gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji publicznych. Szanowni Panowie Ministrowie! Tak jak powiedziałam na początku, inwestowanie w infrastrukturę to ważny element rozwoju komunikacji, ale też gospodarki. są tym elementem, który może w największym stopniu pobudzić gospodarkę w dobie kryzysu i spowolnienia oraz pomagać walczyć z bezrobociem.

Mam pytanie też do pana ministra: Jak teraz rząd zabezpiecza w kontraktach obecnych podwykonawców? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Rafała Webera. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Ja będę mówił o tych pierwszych, natomiast później, w dalszej części wystąpienia, pan minister Andrzej Bittel - o inwestycjach kolejowych. Szanowni Państwo! Inwestycje infrastrukturalne mają na celu stworzenie spójnych, sprawnych połączeń drogowych i kolejowych. Mają one spowodować, że przewóz ludzi lub rzeczy będzie bezpieczny, komfortowy, wygodny i punktualny. Drogi szybkiego ruchu skracają dystans, powodują, że podróż między punktami A i B jest szybsza i krótsza. Dziękuję całemu klubowi Prawo i Sprawiedliwość za tę informację.

W takim bardzo telegraficznym skrócie opowiem o wartościach inwestycji w ramach programów rządowych, programów, które zostały stworzone i są realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i pana premiera Mateusza Morawieckiego. W tej chwili są to cztery programy. W ramach tego programu w tej chwili, czyli konkretnie dzisiaj, w realizacji znajdują się 94 zadania o wartości blisko 53 mld zł. Tak że to są te środki, które teraz są już zaangażowane, które są przekazywane polskim wykonawcom i podwykonawcom, które pracują na rzecz polskiej gospodarki.

One nie tylko spowodują, że będziemy mieli bezpieczne, wygodne, komfortowe połączenia drogowe, ale również sprawią, że te środki zostaną wpompowane w polską gospodarkę. W tym roku ogłosimy co najmniej 15 przetargów na realizację tych zadań, tak że to kolejne środki finansowe, które zaangażujemy. Takie obwodnice jak Żodyń, Gostyń, Gryfino, Strzelce Krajeńskie, Brzezie, Wąchock - te przetargi zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Na tę chwilę mamy podpisanych 71 programów inwestycyjnych, oczywiście z biegiem czasu będziemy podpisywać kolejne. Fundusz Dróg Samorządowych - w tym roku 3200 mln zł jako wsparcie rządowe na inwestycje w drogi lokalne. To pozwoli ogłosić blisko 2300 przetargów w ramach listy podstawowej, ale już mamy informacje o oszczędnościach, już mamy informacje o tym, że do tej listy podstawowej będą dołączone zadania z listy rezerwowej, tak że kolejne dziesiątki zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych będą realizowane. Pan minister finansów w ciągu najbliższych dni będzie sukcesywnie informował samorządowców o tym, że subwencja będzie zwiększana i będą oni mogli realizować zadania inwestycyjne. I bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Andrzeja Bittela. Wysoka Izbo! Realizujemy wiele przedsięwzięć kolejowych, o których państwa często i licznie informujemy. Najważniejszy, „Krajowy program kolejowy”, który jest programem niezwykle zaawansowanym, którego wartość wzrosła o 10 mld od momentu jego uchwalenia, który służy rozwojowi infrastruktury liniowej, mającej na celu jak najlepsze skomunikowanie różnych części Polski ze sobą, jest realizowany na poziomie ponad 56%, zakończony w

Program inwestycji dworcowych”, strategia taborowa - pani poseł o tym wspominała - to są programy, które mają na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury kolejowej, ale też zapewnienie dobrego, przyjaznego, przyjemnego przejazdu. Liczymy, że polscy pasażerowie i goście licznie wrócą na polską kolej. Dziękuję bardzo. Tych zgłoszeń jest bardzo dużo.

Pierwsza pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Bardzo cieszą te dane podane i przez panią poseł Barbarę Bartuś, i przez panów ministrów Webera i Bittela. To są fakty i choćbyśmy chcieli zaklinać rzeczywistość, tak one wyglądają. Cieszy fakt, o którym wczoraj usłyszeliśmy, że to Polska właśnie, na skutek zabiegów pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, [[Wesołość na sali]] wspólnie z krajami Unii Europejskiej (Oklaski), Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza.

To ogromne pieniądze z tarcz finansowych przeznaczone na rozbudowę takich działań (Dzwonek), jak drogi dla polskich wykonawców.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę o trzymanie się limitu czasu, żeby wszyscy państwo mogli zadać pytania. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Propaganda. To miał być pokaz sukcesu, ale niestety prawda jest inna. Luxtorpeda”, program zapowiadany przez premiera Morawieckiego, leży. Gdy chodzi o projekty kolejowe - opóźnienia, opóźnienia, zejścia wykonawców z placów budów. Leży linia kolejowa nr 7 Warszawa - Lublin, leży linia kolejowa Warszawa - Radom. Gdy chodzi o projekty drogowe - podobnie, opóźnienia. S12, o którą pytała pani posłanka Milczanowska, stoi w miejscu, nic się nie dzieje.

Nawet nieruszona, a przecież ta droga jest wpisana do programu europejskiego sieci TEN-T.

Propaganda, propaganda, propaganda. 2 lata temu nie wykorzystaliście z Krajowego Funduszu Drogowego 2 mld zł. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Przemysław Koperski, Lewica. Nie ma pana posła? Przepraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Pan minister był uprzejmy napisać, że ta linia kolejowa ma niski priorytet. Chciałem podkreślić, że wszystkie samorządy z regionu, miasto Bielsko-Biała, Aglomeracja Beskidzka, powiat cieszyński, Cieszyn, gminy, które leżą na tej trasie, podjęły uchwały, że ta inwestycja jest kluczowa dla subregionu południowego województwa śląskiego. Pan minister twierdzi inaczej. Mówicie państwo również, że wkład 15-procentowy to na dzień dzisiejszy dla samorządów żaden problem. Panie ministrze, 15% z 220 mln zł to jest gigantyczna kwota, której na dzień dzisiejszy samorządy nie mają.

Dziękuję uprzejmie.

Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Chciałem podziękować za tę informację, bo ona jest też przyczynkiem do możliwości zadania pytań.

Specjalnie dla tej inicjatywy powołaliśmy stowarzyszenie wzdłuż drogi Bytom - Kołobrzeg. Są oczywiście odcinkowe obwodnice, ale to naprawdę jest wąskie gardło. To się wiąże też z obwodnicami. Obwodnica Ujścia, obwodnica Obornik czy na południu kończona obecnie obwodnica Kępna. Tu potrzebna jest decyzja. Druga sprawa to obwodnice. Dziękuję za tę informację, że Gostyń w ciągu drogi S12 jest rozpoczęty, ale sąsiednie Jaraczewo nie jest w to włączone. Obwodnica Kalisza też jest w tym wykazie, co prawda nie w tym roku, ale w latach następnych. Dlaczego jest próba zmiany przebiegu tej trasy? Na terenie gminy Skalmierzyce jest wyznaczony ten przebieg.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

Tylko w roku 2019 pojawiła się rekordowa kwota w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - ponad 250 mln zł.

Te drogi oczywiście służą przede wszystkim mieszkańcom, ale również służą rozwojowi gospodarczemu Polski, regionu dolnośląskiego. W tym kontekście chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność, radość za dwa południowe odcinki dróg ekspresowych S3 i S8, bo te odcinki będą przebiegały przez Pogórze Sudeckie. To jest teren, który należy do najbiedniejszych obszarów województwa dolnośląskiego. Dziękuję za te działania. Pojawiły się również decyzje związane z budową nowych obwodnic, m.in. Milicza, również Oławy. W tym kontekście chciałbym spytać pana ministra, czy jest w obecnej sytuacji. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Obietnice to jest to, co najlepiej PiS-owi wychodzi. A ja chciałabym porozmawiać o realizacji tych obietnic i o wiarygodności. W 2017 r. pani minister Rafalska wraz z wojewodą Dajczakiem składali obietnicę, że znajdzie się 1 mln zł na STEŚ dla obwodnicy Słubic. Również we wrześniu, kiedy była kampania wyborcza, takie obietnice składali. Obwodnicę Kargowej w województwie lubuskim obiecał mieszkańcom sam prezydent Andrzej Duda i przedstawiciel GDDKiA. Nie ma. To proszę przypomnieć, panie ministrze, panu prezydentowi, że mieszkańcy województwa lubuskiego lubią, jak się tych obietnic dotrzymuje.

Więcej, osobiście byłam u pana ministra Adamczyka i rozmawiałam o tych sprawach. Pan minister obiecał, że znajdzie rozwiązania. Nie znalazł również (Dzwonek) czasu, żeby mi odpowiedzieć na pytania. Jaka jest wiarygodność pana ministra Adamczyka? Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowni Panowie Ministrowie! Chciałbym w imieniu moich wyborców, wyborców pana posła Hoffmanna i wielu tych, którzy są z okręgu konińskiego, do tych sukcesów, o których mówi rząd, dopisać też północną obwodnicę Koła, którą osobiście obiecał pan premier Morawiecki w czasie kampanii. Chciałbym też, żeby udało się wreszcie zrealizować kompleks handlowo-usługowy z dworcem PKP w Koninie, o którym tutaj 9 stycznia mówił pan minister Adamczyk, że już rozpocznie się ta inwestycja. Chciałbym zapytać, czy ta inwestycja już się rozpoczęła i kiedy jest szansa na jej realizację, podobnie jeśli chodzi o tę obwodnicę Koła, bo tam była mowa, że będzie szansa na listę poszerzoną i że ona się tam znajdzie. Czy się znajdzie, czy się nie znajdzie? Trzecia ważna inwestycja to jest modernizacja drogi krajowej nr 15 Gniezno - Żydowo - Czeluścin w kierunku Wrześni.

Czy jest szansa na to, że te inwestycje znajdą się w programie i będą realizowane ze środków publicznych? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Oddano ją do użytku 17 sierpnia 1877 r., więc blisko 150 lat temu. Przez ten czas właśnie blisko 150 lat wielokrotnie była modernizowana, przebudowywana, ale dopiero dzięki pieniądzom Unii Europejskiej, tak można powiedzieć, jest całościowa próba przebudowania tej linii.

Czy zostanie przy tej modernizowanej linii taki obraz zniszczeń?

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że nie od razu zbudowano Kraków. Tak. Nie daliście rady. Nie zmarnujcie tego, co rozpoczęliśmy siłą polskich firm, siłą miliardów złotych z polskiego budżetu i budżetu Unii Europejskiej. Jak możecie mówić dzisiaj na konferencji w obecności pana prezydenta i premiera, chwaląc się budżetem Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć, że ten budżet, wynoszący 60 mld euro, 37 mld w dotacjach, pozostałe w pożyczkach, wymaga, po pierwsze, tego, czego nie rozumiecie: spełnienia wymogów ładu ekologicznego i państwa prawa. Przestrzegam więc was: przestrzegajcie prawa, żeby nie zmarnować tych pieniędzy, które mają trafić do polskiego budżetu. To miesiące pracy.

2 lata opóźnienia. Kiedy będzie zakończenie? O to chciałem państwa zapytać, prosząc o odpowiedź, bo w tej sprawie, w sprawie tych inwestycji po prostu nie daliście rady.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na konferencji prasowej z przejeżdżającymi pociągami - proszę państwa, to jest bardzo ważny szczegół - hucznie zapowiedziany został program 200 prezydenckich przystanków. Na stronie internetowej można zapoznać się z informacją na ten temat, która kończy się stwierdzeniem: Program jest otwarty na zmiany i nowe propozycje. I właśnie: Czy to jest już zatwierdzony program? A może jakaś wstępna faza projektu? Chciałabym się dowiedzieć, kto i do kiedy może składać propozycje zmian czy nowych przystanków. Czy będą konsultacje z samorządami i organizacjami i kiedy poinformuje o nich ministerstwo? Jakiego rodzaju finansowanie jest przewidziane? Koszt budowy czy modernizacji w 100% będzie pokrywany przez państwo czy przewidywany jest obowiązkowy wkład samorządów? A jeżeli tak, to na jakim poziomie? Jak wyglądają ramy czasowe poszczególnych etapów w tym programie? I wreszcie, czy ministerstwo będzie realizowało program 200 przystanków prezydenckich, nawet jeżeli prezydent Andrzej Duda nie zostanie wybrany na prezydenta na drugą kadencję?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie o drogę S12, a mianowicie o odcinek od Piotrkowa Trybunalskiego do Kozenina, który stanowi obwodnicę miejscowości Sulejów. Dlaczego w tej sprawie nic się nie dzieje? Mimo że rok temu została wydana decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności, do dzisiaj nic się nie dzieje. Dlaczego mimo obietnic posłów Prawa i Sprawiedliwości nawet nie zaplanowano węzła włączającego do autostrady A1, która właśnie jest budowana? To są zasadnicze pytania przede wszystkim mieszkańców Sulejowa, którzy uważają, że to jest najważniejsza inwestycja w historii Sulejowa, którzy uważają, że bez tej inwestycji nie da się tam normalnie żyć.

Dlaczego mimo interpelacji, mimo stanowisk samorządów, mimo podpisów mieszkańców państwo wciąż nie zgadzają się na wybudowanie tego przystanku kolejowego? Przypominam, że w powiecie rawskim nie ma żadnego przystanku, najbliższe są kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Opocznie i w Skierniewicach.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Ewa Szymańska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Są to obwodnice Głogowa, Kaczorowa i Legnicy, w której mieszkam. Obwodnica Legnicy ma być budowana w ciągu drogi krajowej nr 94 i będzie przebiegać zarówno w granicach administracyjnych Legnicy, jak i poza nią. Budowa obwodnic w dużej mierze uzależniona jest od dobrej współpracy z miejscowymi samorządami. Wiem, że w części miejskiej media informowały już o rozpoczęciu prac. Jest to najbardziej zakorkowany odcinek tej autostrady. Nie ma pasa awaryjnego. Są prowadzone prace dotyczące wyboru najlepszej koncepcji zmiany tej sytuacji, czy to poprzez dobudowanie kolejnych pasów ruchu wraz z pasem awaryjnym, czy to budowanie drogi równoległej z innym przebiegiem. Proszę o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie już są te prace.

Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o nazwy i obietnice, to wymyślacie rzeczy pięknie, natomiast w praktyce jest bieda. W 2012 r. rząd Platformy i PSL-u oddał pierwszy odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy, obwodnicę Mińska Mazowieckiego, po 4 latach od objęcia rządów. Po 5 latach waszych rządów nie skończyliście nawet tego drugiego odcinka, który my rozpoczęliśmy w 2015 r. I tak wygląda ta historia waszych rządów. W państwie, gdzie następuje zmiana rządów, powinna być kontynuacja najważniejszych spraw dla państwa, takich jak budowa infrastruktury drogowej. To nic nadzwyczajnego. Jak są pieniądze, to powinny być drogi. To jest efekt waszych rządów. Kolejnym wielkim problemem jest brak bezkolizyjnych skrzyżowań kolei z drogami. Wymyślacie jakiś program „Kolej+” Dlaczego nie ma bezkolizyjnego skrzyżowania w dużym mieście powiatowym Mińsku Mazowieckim? Dlaczego nie ma takiego skrzyżowania w mieście Mrozy?

Róbcie normalną rzecz. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Droga S10 Bydgoszcz - Toruń to droga kluczowa dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, to droga oczekiwana przez mieszkańców, gdyż droga ta była dla wielu mieszkańców naszego województwa, dla wielu naszych krewnych i przyjaciół drogą ostatnią. Droga ma być realizowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi S10 13 lutego pytałem, kiedy można się spodziewać wniosku do Eurostatu w sprawie zaopiniowania realizacji tej drogi w formule PPP. Takie zaopiniowanie jest niezbędne, aby Rada Ministrów mogła podjąć w tej sprawie stosowną uchwałę. Przedstawicielka ministerstwa poinformowała, że taki wniosek został złożony. Z rozmów z przedstawicielami Eurostatu wynika, że wydanie takiej decyzji jest bliżej niż dalej. Tymczasem niedawno pan, panie ministrze, poinformował, że taki wniosek nie został złożony. Niedawno członek Rady Ministrów pan Łukasz Schreiber poinformował, że prace w ramach tej drogi są na końcowym etapie i Rada Ministrów za kilka dni ma przyjąć dokument w tej sprawie. To dokument będzie bez opinii Eurostatu? Wiem, panie ministrze, że panu trudno będzie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć wobec tej deklaracji pana ministra Schreibera.

Prosiliście, by wszyscy mogli zadać pytania, więc proszę trzymać się czasu i szybko podchodzić do mównicy, bo tracimy czas. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, PSL-Kukiz15. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Temat obwodnicy Pyrzyc. Niestety państwo piszecie w swoim programie wieloletnim, że chcecie otworzyć linię kolejową Stargard - Myślibórz, natomiast generalna dyrekcja, szanowni państwo, już realizuje obwodnicę Myśliborza, uniemożliwiając w tej sposób, szanowni państwo, odtworzenie tej linii. Marszałek województwa chce wyłożyć pieniądze na budowę obwodnicy Pyrzyc, mieszkańcy, gmina Pyrzyce też. Państwo nie chcecie zgodzić się na to, żeby na starej linii kolejowej tę obwodnicę zbudować. Odpuśćcie sobie, szanowni państwo, bo jeżeli odpuściliście w Myśliborzu, to już nie ma sensu odtworzenia tego. Dajcie zgodę. Nie chcemy od was pieniędzy, tylko pozwólcie zrealizować samorządom lokalnym obwodnicę Pyrzyc. Potrzebujemy tylko zgody, szanowni państwo.

Samorządy wiedzą, jak to zrobić. Prosimy, żebyście nie trwali w tym uporze, bo to nie ma sensu. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zanim przejdę do najważniejszej inwestycji zarówno dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, jak i dla Śląska, czyli odbudowy kolei Jastrzębie-Zdrój - Katowice, przypomnę kilka faktów.

I dziękujemy za to, że tak bardzo sprawnie działają. Dali radę. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że ta inwestycja, która jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości, czyli Jastrzębia-Zdroju, blisko 100-tysięcznego miasta, ma szansę realizacji dzięki działaniom obecnego marszałka województwa śląskiego pana Chełstowskiego, który daje możliwość przesunięcia tej inwestycji dość wysoko w rankingu, jak również projektowi, który przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. To jest, szanowni państwo, 525 mln dla tej inwestycji. Dzisiaj jest pytanie: Czy samorząd Jastrzębia-Zdroju, okolicznych miejscowości da radę? Wysoka Izbo! Przez ostatnie 5 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości starał się dorównać sukcesom w budowie dróg, szybkich tras Platformie Obywatelskiej i PSL.

Nie daliście rady. Jeszcze gorzej jest w moim okręgu wyborczym. Co zrobiliście przez te 6 lat? Zdołaliście podzielić ten projekt na sześć etapów i dopiero teraz, w maju tego roku, została podpisana umowa na pierwszy etap. Panie ministrze, to są fakty. która ogłasza sukces budowy drogi w 2016 r., otoczona wianuszkiem posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie zrobiliście jej, w ogóle jej nie ma w finansowaniu. To droga łącząca Bielsko-Białą z Krakowem, jedna z kluczowych dróg i bardzo potrzebna. Nie zrobiliście tego. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł Wiesław Szczepański. A pan poseł Stefan Krajewski przygotowuje się do wystąpienia. Panowie Ministrowie! Powiedział pan minister, że w tej chwili rząd, ministerstwo rozpoczęło nabór do programu „Kolej+”

Powiedział pan wcześniej, panie ministrze, że przecież sprzedano bilety miesięczne.

Chciałbym wiedzieć, czy on został zrealizowany czy nie. W świetle tego, co dzieje się dzisiaj, jeśli chodzi o tabor kolejowy, czy państwo nie powinniście wziąć pod uwagę ewentualnie roli wiodącej jako zamawiający i umówić się z marszałkami, że zakup elektrycznych zestawów będzie organizowany centralnie, dlatego że dzisiaj kupno pojedynczego zestawu to są olbrzymie koszty? Bardzo proszę, pan poseł Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Litwa, Łotwa i Estonia dużo lepiej sobie radzą z budową Rail Baltica w porównaniu z Polską. Raport NIK, który pojawił się w 2019 r., nie zostawia suchej nitki na działaniach zarówno ministerstwa, jak i PKP PLK. Opóźnienia, pieniądze, które są wydawane w sposób niewłaściwy, niegospodarny. Wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego, mieszkańcy Białegostoku czekają na to, że nastąpi przyspieszenie Wszystko się ciągnie, ślimaczy, nie ma działań na tych drogach. Czy mamy wydawać pieniądze na kolejne projekty, na kolejne planowane przebiegi tej obwodnicy zamiast na wykonanie odcinka przebudowy?

Oczywiście chwalicie się, jak to wszystko pięknie wygląda. 22 miesiące opóźnienia na trasie Lewki - Hajnówka, mała trasa, nawet nie ma trakcji elektrycznej. Dziękuję. Przygotowuje się pani poseł Małgorzata Pępek. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rząd Prawa i Sprawiedliwości daje radę. Dajemy radę. A oto konkrety. Fundusz Dróg Samorządowych - historyczny, jakiego dotąd nie było. 36 mld zł na modernizację i budowę dróg powiatowych i gminnych.

Panie ministrze, mieszkańcy mojego regionu i samorządowcy dziękują bardzo za to, że będą mogli jeździć nowoczesnymi i bezpiecznymi drogami. Ale dajemy radę także, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, bo „Krajowy program kolejowy do 2023 r.” to również program historyczny, to ponad 75 mld zł, ale to także program inwestycji dworcowych, o który chcę zapytać. Jest blisko 200 dworców do modernizacji, w tym także długo oczekiwana modernizacja dworców we Włocławku i w Grudziądzu. Panie Ministrze! Czy wobec sytuacji walki ze skutkami gospodarczymi koronawirusa te inwestycje dworcowe we Włocławku i w Grudziądzu nie są zagrożone? Bardzo proszę o uspokojenie w tym zakresie mieszkańców. Tak jak było powiedziane na początku, bardzo ważna jest realizacja inwestycji, ponieważ to właśnie one (Dzwonek) stymulują gospodarkę. Przygotowuje się pani poseł Wanda Nowicka. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W sprawie inwestycji infrastrukturalnych na Żywiecczyźnie, Podbeskidziu i ziemi cieszyńskiej mieliśmy prawdziwy festiwal obietnic ze strony przedstawicieli PiS-u. Najlepiej wam wychodzi propaganda, lecz nie realizujecie tego, co obiecaliście. Priorytetowa inwestycja, którą należy wykonać, to odcinek drogi ekspresowej S52: Bielsko-Biała - węzeł Suchy Potok - Wadowice - Głogoczów - Kraków, czyli tzw. Beskidzka Droga Integracyjna. Świetnie obiecywaliście.

Następna inwestycja: dokończenie rewitalizacji linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń na odcinkach Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Lipnik z dobudową drugiego toru oraz Wilkowice Bystra - Łodygowice - Żywiec, z dobudową również drugiego toru, i Cięcina - Zwardoń. Kolejna ważna inwestycja: rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Jeleśnia - Sucha Beskidzka. Nie można również zapomnieć o dofinansowaniu na rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku [[Dzwonek]] Bielsko-Biała - Skoczów.

Przygotowuje się pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Ja bez kartki, jakby co. Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie dotyczy planowanej drogi ekspresowej S11 w śladzie drogi krajowej nr 11, która ma być kluczowa dla połączenia północy Polski, Kołobrzeg, z południem, Piekary Śląskie, i łączyć się z autostradą A1 w województwie śląskim. Inwestycja ta napotyka coraz to nowe problemy, a jej realizacja jest ciągle przesuwana. W Tarnowskich Górach ma powstać obwodnica miasta oraz odcinek, który zakłada przecięcie miasta między dwiema dzielnicami, odcinając praktycznie jedną z nich. Koszt inwestycji dla województwa śląskiego to ok. 3 mld zł. Dla 60-kilometrowego odcinka, w większości planowanego po nowym śladzie, miał być wybrany ostateczny wariant przebiegu drogi. Sam projekt kosztować ma blisko 3 mln zł. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie drogi dla regionu, jak i całego kraju, proszę o odpowiedź na piśmie. Jakie są przyczyny tak dużych opóźnień w realizacji tej inwestycji? Czy znany jest ostateczny przebieg i czas realizacji inwestycji? Czy wzięto pod uwagę protesty mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy alarmują, że droga praktycznie (Dzwonek) podzieli miasto i zniszczy tereny zielone, w tym lasy. Dziękuję. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Zrównoważony rozwój naszego kraju, naszej ojczyzny to są fakty, to są działania. To nie są puste słowa, to nie są obietnice z czasów tekturowego państwa i kamieni kupa.

Tutaj jest więc dbałość właśnie o tę Polskę powiatową, Polskę gminną. Ogłoszony w maju br. przez pana prezydenta i ministra infrastruktury program przystankowy zakłada wybudowanie 200 przystanków. To po pierwsze. I trzecie pytanie: Czy jest to lista zamknięta?

Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo Ministrowie! Panie i Panowie Posłowie! Państwo z PiS-u, jesteście ekspertami. Rzeczywiście jesteście ekspertami, ale nie w dziedzinie rozwoju i infrastruktury, lecz propagandy sukcesu, PR-u, za 2 mld zł podarowane publicznej telewizji. Ale jednak niszczycie: kolejowy Y, tak ważny dla całej Polski. Budujecie autostradę w taki sposób, że jest to piekło dla wszystkich podróżujących między Łodzią a Katowicami. Wasz wojewoda ogłosił budowę obwodnicy Nowosolnej przez środek wpisanego do rejestru zabytków skrzyżowania. Nie daliście państwo rady i nie dacie. Proszę o informacje na ten temat na piśmie, szanowni państwo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Czuję się do tego szczególnie upoważniony, ponieważ przez 4 lata jako przedstawiciel rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojewoda wielkopolski partycypowałem w realizacji tego programu. Przede wszystkim chcę podziękować panom ministrom za ten program, bo to jest program przełomowy, szanowni państwo. Zdecydowanie daliśmy radę, dlatego że to jest program, który pozwala przebudowywać, budować. To jest program, który wspiera samorządy, i to na terenie całego kraju - 36 mld zł. Dla mojej Wielkopolski to jest 700 tys. dotychczas na realizację tego programu. To są pieniądze, szanowni państwo, które docierają do tych najmniejszych gmin - wcześniej te samorządy z powodu swoich ograniczeń budżetowych nie mogły budować dróg powiatowych i gminnych. Teraz mogą. I to jest kwestia fundamentalna. I, szanowni państwo, może pewna niespodzianka dla was. Otóż także w imieniu waszych samorządowców z Wielkopolski chcę podziękować panom ministrom, chcę podziękować panu premierowi, bo takie sygnały odbierałem i jako wojewoda, i także teraz jako poseł. Pan minister rozwiał wszelkie moje wątpliwości, mówiąc, jakie będą środki na realizację tego programu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Wiem, że kilka przetargów zostało już ogłoszonych, głównie w ramach południowej obwodnicy Białegostoku, ale żaden chyba jeszcze nie został rozstrzygnięty, a jeden został unieważniony. Co z obwodnicą Siemiatycz, co z obwodnicą Bielska Podlaskiego? Jest to droga śmierci, w każdym tygodniu są tam wypadki. W jakim standardzie będzie budowana i w ogóle czy będzie ona przebudowana? Panie Ministrze! Jeszcze kilka pytań odnośnie do kolei. Kolejowa obwodnica Białegostoku, bardzo ważna inwestycja. Zaproponowaliście wiele wariantów, ale niestety na większość z nich nie zgadzają się mieszkańcy. Kiedy w końcu zostanie wyłoniony konkretny wariant i kiedy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami? Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Na koniec jeszcze odcinek Białystok - Czyżew. Został rozstrzygnięty przetarg, są duże opóźnienia. Kiedy mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli się cieszyć szybką koleją między Białymstokiem a Warszawą? Jaka to będzie kolej, jakich prędkości, bo też jest wiele wątpliwości co do tego, i kiedy ta inwestycja zostanie zakończona? Bardzo proszę, pan poseł Paweł Rychlik. Potem przygotowuje się pan poseł Suchoń. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W 2014 r. powstała droga ekspresowa S8 łącząca Warszawę z Wrocławiem, przebiegająca przez Sieradz. Spowodowało to wygenerowanie dodatkowych obciążeń na drogach krajowych nr 45 i 43 i w sumie codzienne zakorkowanie i paraliż Wielunia. Jako poseł, a zarazem mieszkaniec Wielunia podjąłem działania mające na celu przybliżenie tego problemu w generalnej dyrekcji, jak i w Ministerstwie Infrastruktury. I tutaj serdecznie dziękuję za wielokrotne spotkania z panem ministrem Adamczykiem, z panem ministrem Weberem, z panem ministrem Żuchowskim z generalnej dyrekcji, co skutkowało opracowaniem planu przebiegu tej obwodnicy, która łączy drogi krajowe przebiegające przez Wieluń.

W związku z powyższym pragnę zapytać, na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji, tak samo inwestycji dotyczącej Błaszek i Łowicza. Wskutek pandemii, czego pokłosiem jest kryzys gospodarczy, który mimo wszystko tak głęboko Polski nie będzie dotykał. Pytanie: Czy program 100 obwodnic nie jest zagrożony, a te drogi będą budowane (Dzwonek) zgodnie z wcześniejszym harmonogramem? Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Przepraszam za wcześniejsze problemy komunikacyjne.

Otóż sam Fundusz Dróg Samorządowych pozwolił na sfinansowanie ponad 200 km dróg. To 170 zadań: 42 drogi powiatowe, 128 dróg gminnych.

Kolejny program, program 100 obwodnic, pozwolił na przygotowanie inwestycji dla budowy siedmiu obwodnic: obwodnicy Limanowej, Nowego Targu, Piwnicznej, Makowa Podhalańskiego, wschodniej obwodnicy Tarnowa, Trzebini czy Wadowic. Tutaj trzeba zwrócić w szczególności uwagę na obwodnicę Piwnicznej, która jest projektowana, a która pozwoli na przyszłe połączenie również projektowanej sądeczanki z obwodnicą Piwnicznej i stworzenie szybkiego szlaku komunikacyjnego do granicy państwa. Chciałbym na zakończenie też podziękować za prace, które trwają nad sądeczanką oraz koleją Podłęże - Piekiełko.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, przygotowuje się do zadania pytania. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z przykrością muszę powiedzieć, że w ostatnich miesiącach Ministerstwo Infrastruktury zamieniło się raczej w ministerstwo inwigilacji i propagandy. Inwigilację w przewozach kolejowych wszyscy widzieliśmy, to jest skandaliczne, natomiast ta propaganda poraża. Choćby inwestycje w drogi szybkiego ruchu - w tym roku zaledwie 12 mld zł, to jest zaledwie 60% tego, co było w roku poprzednim. Czas od otwarcia ofert do podpisania umowy wydłużył się ze 118 dni w 2014 r. do 241 w 2018 r. - absolutna nieudolność - nie mówiąc już o czasie od ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy z wykonawcą: w poprzedniej perspektywie - 355 dni, 2018 r. - 723 dni. To jest absolutny nokaut organizacyjny i nie dziwię się, że nie ma pana ministra Adamczyka, który lubi błyszczeć w blasku fleszy podczas konferencji prasowych, ale kiedy trzeba odpowiadać na trudne pytania, to pana ministra nie ma. Jeżeli popatrzymy na program 100 obwodnic, to tak dziwnie się składa, że przez najbliższe 3 lata niemalże się nie dzieje nic, a eksplozja następuje przed kolejnymi wyborami. Ze zdziwieniem usłyszałem, że linię 190 z Bielska-Białej do Cieszyna ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości, rząd PiS uważa za mającą niski priorytet.

to są rzeczy, które nas dzisiaj interesują. Pan poseł Krzysztof Gadowski przygotowuje się. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Na początku krótki apel, zwłaszcza do tej części opozycji, która w sposób wyjątkowo nieudolny pokazuje tutaj również jakieś karteczki z napisami, żebyście państwo najpierw uzgodnili między sobą i ze swoim kandydatem na prezydenta panem Rafałem Trzaskowskim kwestie likwidacji inwestycji, które są w strategii państwa polskiego na wiele najbliższych lat.

Druga kwestia. Nie powiedział tego pan minister, a warto to podkreślić: jest deklaracja jasna rządu dla rynku, również wykonawców, o tym, iż na inwestycjach infrastrukturalnych rząd nie będzie oszczędzał. I to powinno wybrzmieć właśnie w tym czasie kryzysu, trudnym dla gospodarki, dla życia społecznego. Po trzecie, chciałbym również do jakiegoś konkretnego przykładu się odwołać i chciałbym prosić pana ministra o udzielenie odpowiedzi na temat stanu przygotowań do budowy przyszłej odcinka drogi S11 w województwie śląskim, 54 km. Wspominali tutaj niektórzy posłowie o różnych innych (Dzwonek), bym powiedział, miejscach w kraju.

Pan poseł Krzysztof Gadowski. Pan poseł Marek Polak przygotowuje się. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! To wam świetnie wychodzi i to trzeba powiedzieć. To jest ten program rozpisany, który realizujecie. Ja myślałem, że dzisiejsza dyskusja będzie o tym, co udało się rządowi Prawa i Sprawiedliwości zrealizować w ramach tych programów. Oczywiście otwieracie kolejne nowe, dzieje się to zawsze przed wyborami. Były obietnice, że coś będzie robione, były obietnice, że będzie realizowana inwestycja, że miasto Jastrzębie zostanie połączone z Katowicami, ba, że pójdzie to dużo dalej. Przyjechał pan minister Horała, który mówił, że Jastrzębie zostanie włączone w nitkę szybkiej kolei, aż do dworca centralnego i dalej. Panie ministrze, w ramach tych programów chyba się troszkę zakiwaliście. Chciałem zapytać: Z jakiego w końcu programu czy w ramach którego programu inwestycja dla Jastrzębia będzie zrealizowana - czy w ramach tego programu dużych prędkości z połączeniami transgranicznymi, czy w ramach programu „Kolej+” Naprawdę trudno dzisiaj się doczytać, skąd i za jakie pieniądze będzie ta inwestycja realizowana. Pan poseł Marek Sowa przygotowuje się. Zdalnie? Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

To bardzo dobry program, który daje możliwość nie tylko rewitalizacji istniejącej i zlikwidowanej infrastruktury, ale otwiera też drogę do budowy nowych połączeń kolejowych, zwłaszcza w małych, wykluczonych komunikacyjnie miejscowościach. Myślę, że rozwój lokalnej infrastruktury kolejowej znacznie ułatwi mieszkańcom tych miejscowości dostęp do wielkomiejskich ośrodków akademickich, dużych stref przemysłowych, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju, a także do rozwijania umiejętności, talentów i zainteresowań. Krótko mówiąc, poszerzy ich horyzonty zarówno myślowe, intelektualne, jak i gospodarcze. Chciałem więc zapytać pana ministra, jak duże jest zainteresowanie samorządowców tym programem. Proszę bardzo, pan poseł Marek Sowa. Wysoka Izbo! Byłem przekonany, że pani Bartuś, przedstawiając pytania odnośnie do tej informacji, zada dramatyczne pytanie: Dlaczego nie budujecie sądeczanki? Jedyne, co przy sądeczance zrobiliście, to przesunęliście budowę tej inwestycji do roku 2028. Pytam: Dlaczego to robicie mieszkańcom Sądecczyzny? Uwięziliście tę drogę na liście rezerwowej i nie macie zamiaru jej budować. A przecież wszystko się miało w 2015 r. zmieniać.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość. Przygotowuje się pan poseł Frysztak. Wysoka Izbo! Tak, rzeczywiście, drodzy państwo, daliście radę - zlikwidować tysiące kilometrów linii kolejowych, to wam się udało. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować za program „Kolej+”, który został ogłoszony kilka miesięcy temu, a kilka dni temu ogłoszono nabór na ten program. Cieszę się, że takie miejscowości jak Turek w Wielkopolsce, prawie 30-tysięczne miasto, będą miały możliwość uczestniczyć w tym programie. W związku z tym chciałem zapytać, ilu Polaków zostało wykluczonych z komunikacji kolejowej poprzez działania rządu PO-PSL.

Jak wiemy, gminom i powiatom będzie ciężko, a wiele urzędów marszałkowskich myśli tylko o dużych metropoliach, dlatego chciałbym, abyście państwo ministrowie nakłaniali urzędy marszałkowskie do tego, by w tym programie uczestniczyły.

Panowie Ministrowie! Na początek panów zaocznie przeproszę, dlatego że będę się nad wami pastwić. Dlaczego? Konkretne przykłady: najlepiej wychodzi wam opowiadanie, wdrażanie kolejnych projektów i wszystkie muszą mieć „+” Dziś wasz minister mówi, że będziecie robić warzywniak+. Gratuluję, ale najpierw skończcie to, co zaczęliście, bo nie skończyliście niczego.

Przetarg nadal nie został ogłoszony, a obiecujecie nowe przystanki na tej linii. Jeśli chodzi o linię kolejową nr 8 relacji Radom - Warszawa, tak ważnej dla lotniska w Radomiu, to przypomnę: Już prezes Merchel mówi, że będzie opóźnienie. Jesteście po czasie. Wy ze wszystkim sobie nie dajecie rady. Na budowie tej linii kolejowej hula wiatr, hula wiatr, dosłownie, brak ekip. Jeśli chodzi o to, co wam najlepiej wychodzi, to obietnice, np. obietnica budowy S12. Tam staracie się robić dużo zamieszania. Co w tym czasie zrobił? W tym czasie nic nie zrobił. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Dlaczego się nie znalazł? Dlatego że rządzący wtedy burmistrz z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że perspektywa roku 2023 jest za daleka i on to zrobi ze środków samorządu, nie będzie się starał o to, żeby dworzec był na tej liście. Oczywiście kadencja samorządu się skończyła, burmistrza już nie ma. Dzisiaj mamy rok 2020, a dworzec jest niezrobiony. Pierwsze pytanie. Czy jest szansa, żeby po roku 2023 podobny program był realizowany i żeby wtedy dworzec szczecinecki znalazł się na liście? Druga rzecz. Pewną cechą rządów Platformy Obywatelskiej było to, że zwijaliście Polskę powiatowo-gminną. Likwidowaliście połączenia autobusowe, połączenia kolejowe. Czy macie panowie taką informację? Jakie działania podejmujecie, żeby zmniejszyć wykluczenie komunikacyjne obywateli Polski? W odniesieniu do tych zarzutów, które tutaj padają, jedna rzecz. Państwa obietnice, rok 2015. Koncert życzeń.

z PiS-u! Na tej liście był dworzec w Koszalinie, osobiście pan minister Szefernaker i pan poseł Hoc obiecywali remont swoim wyborcom. Jak straszył, tak straszy dalej. Na tej liście był dworzec w moim mieście powiatowym, w Gryficach, w którym, panie ministrze, żeby osoba niepełnosprawna mogła wjechać do pociągu, musi zadzwonić do maszynisty, a ten wtedy zatrzymuje pociąg 200 m przed dworcem, bo tam jest stara towarowa rampa, i tam ta osoba na wózku może wjechać do tego pociągu. To jest ten właśnie program+.

Nie ma nic. Po prostu nie dajecie rady, niestety. To jest jedyny port lotniczy, który obsługuje północno-zachodnią Polskę, jedyny port lotniczy, który obsługuje 3 mln mieszkańców, dalej jest już tylko Berlin. To jest port lotniczy, w którym pan ma 42% udziałów, czyli jest pan większościowym udziałowcem.

Pan poseł Andrzej Szewiński przygotowuje się do pytania. Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo!

A przykładem tego, że daliśmy radę, jest oddanie obwodnicy Częstochowy przed terminem. Tak, panie ministrze, czy nie? Szanowni Państwo! Chciałbym podziękować panu premierowi i rządowi Prawa i Sprawiedliwości za Fundusz Dróg Samorządowych, który za waszych czasów... Schetynówki.

Pan poseł Andrzej Gawron przygotowuje się do zadania pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odniosę się też do obwodnicy, o której wspomniał mój przedmówca. Jeszcze kilka miesięcy temu, będąc wiceprezydentem miasta Częstochowa, słyszałem. o tym, że obwodnica będzie miała stawkę zerową, jeżeli chodzi o opłaty. Dlatego moje pytanie jest następujące: Czy stawka zerowa będzie podtrzymana?

Niestety pod Częstochową właśnie w tym miejscu musicie państwo czekać. Mam nadzieję, że te obietnice będą dotrzymywane i że uda się państwu. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Gawron. Pani poseł Małgorzata Janyska. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie!

Prosiłbym, żeby o tym pamiętać. Ta miejscowość jest przedzielona drogą krajową DK46.

Jeżeli chodzi o dzisiejszą dyskusję, to chciałbym się zwrócić do posłów opozycji, szczególnie do posłów Platformy Obywatelskiej.

Zostały zmienione warunki, na których te drogi mogły powstawać. Ludzie nawet kilkanaście lat czekali na to, żeby w tej chwili te drogi zostały wybudowane. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Zaproponowane rozwiązania to cztery warianty. Pierwsze dwa dotyczą obwodnicy od strony północnej Janowa Lubelskiego, trzeci i czwarty - od strony południowej, ale forsowany do realizacji jest wariant pierwszy i drugi, wariant, który dzieli miejscowości Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Poduchowna kosztem wyburzenia domów, wyburzenia gospodarstw, bo tak zaplanowaliście. 700 gospodarstw podpisało się pod protestem do generalnej dyrekcji dróg i autostrad, a także do urzędu miasta Janów, od którego ludzie zostaną odcięci właśnie tą drogą, którą im obiecaliście, bo obiecujecie i planujecie bez sensu. Ludzie nie po to czekali latami na obwodnicę Janowa, żeby dzisiaj pozbawiać ich domostw. Kolejna rzecz. Kolejna kwestia. Dlaczego, panie ministrze? bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wtedy Rzeszów uzyska najszybsze połączenie komunikacyjne z Warszawą przez Lublin.

Chciałbym uzyskać od panów ministrów zapewnienie, że ta inwestycja jest i pozostanie priorytetem rządu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Ireneusz Raś, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Waldemar Andzel przygotowuje się do pytania. Wysoki Sejmie!

No to o czym my mówimy?

To wszystko będzie. To są kluczowe odcinki i wszystko leży. Pani poseł Bartuś, która teraz wychodzi, mówiła, że samorząd nie daje rady.

No tną te inwestycje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości inwestycje infrastrukturalne są priorytetowe.

Zadanie podzielone jest na etapy.

Chciałbym uzyskać informację na temat inwestycji lotnisko - Podwarpie, czyli budowy drugiej jezdni oraz przebudowy drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Na jakim etapie są obydwie inwestycje? Kiedy planowane jest zakończenie ww. zadań? Jeszcze raz dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości za inwestycje infrastrukturalne, które są realizowane w kraju. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mimo wielu dzielących nas różnic zawsze wspieram działania rządu w zakresie rozwoju transportu publicznego. Ok. 14 mln osób w Polsce nie ma dostępu do komunikacji zbiorowej. To dramat szczególnie mniejszych miejscowości, których mieszkańcy nie mają jak dojechać do szkoły, do pracy, do lekarza. Program „Kolej+” był wielką szansą na zmianę tego stanu rzeczy. Okazuje się, że obiecane przez premiera Morawieckiego tysiące kilometrów linii kolejowych nie powstaną, albo - przepraszam - powstaną, ale tylko na papierze. Bardzo mi przykro, ale nie daliście rady. Przez deformę oświaty, walkę z pandemią, inflację oraz rosnące koszty budowy linii kolejowych budżety samorządów są w dramatycznej sytuacji. Jak rząd zamierza pomóc tym samorządom, których nie stać na 15-procentowy wkład własny do programu „Kolej+” Co zamierzacie zrobić, by ten program nie był tylko pretekstem do teatralnej sesji zdjęciowej Andrzeja Dudy na dworcu w miejscowości Końskie?

Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Wspomniano tu dzisiaj kolej dużych prędkości, choć po wyjaśnieniach przedstawiciela rządu należałoby to nazwać kolejami nieco mniejszych prędkości. Niestety na pytanie o to, ile kilometrów nowych linii kolejowych wybudowano w ciągu ostatnich 4 lat, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury odpowiedź przedstawiciela rządu brzmiała: zero. W związku z tym trudno ocenić, jak sobie państwo poradzicie z tak ambitnym zagadnieniem. Ale zostawmy na chwilę kolej. Jedną z nowych inwestycji jest budowa brakującego odcinka drogi S7 między węzłami lotnisko Okęcie - Grójec. Z tą trasą ma się krzyżować droga wojewódzka nr 721. Niestety pomimo zabezpieczenia przez marszałka województwa mazowieckiego środków na budowę tej drogi jej budowa, rozpoczęcie tej inwestycji się opóźnia. Dlaczego? Bo od 2 lat Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie jest w stanie rozpatrzyć odwołań od decyzji środowiskowej, a wyznaczone kolejne terminy nie zostały dotrzymane.

Nie można blokować inwestycji drogowych tylko dlatego, że są realizowane przez nielubiany przez rząd samorząd. Takie działanie to jest brak szacunku dla mieszkańców regionu.

żeby do tego nie doszło. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Barbarę Bartuś. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Powtórzę: nie od razu Kraków zbudowano. Ale bez kartek, bez wypisywania kartek możemy stwierdzić: daliśmy radę, dajemy radę i damy w przyszłości radę. Co było za waszych rządów, to już tyle razy było wspominane, ale wystarczy przypomnieć samych waszych przedstawicieli ocenę, którą daliście u Sowy, chyba tak się nazywała ta restauracja. Kamieni kupa. I tak można te rządy, 8 lat koalicji ocenić. I to tak tragicznie bankrutowali, że niektórzy popełniali samobójstwa, tracąc majątek, wcześniejszy dorobek. To za waszych czasów likwidowano połączenia, o których już była tutaj mowa. To za wcześniejszych czasów dochodziło do zwijania Polski, bo to nawet nie tylko za czasów PO, koalicji PO - PSL, bo przecież tory w Polsce likwidowano wcześniej. Miał pan czas, w tej chwili jest mój czas. Ja pragnę podziękować wszystkim tym posłom, którzy wzięli udział w tej debacie. Wzięli udział w debacie, którą zorganizowaliśmy my - na nasz wniosek jest informacja bieżąca, bo my chcemy. Szanowni Państwo! Dzisiaj debatujemy o sprawie, która dotyczy wszystkich Polaków, o sprawie bardzo ważnej, o infrastrukturze drogowej, ale też debatujemy w dobie pandemii, jaką mamy, o polskich przedsiębiorcach, czy będą mieli dalej pracę, czy te inwestycje, które dotąd były realizowane, są realizowane, czy będą realizowane. I powiem coś bardzo ważnego, ale nie odkrywczego. Wszystko da się zrobić, jeżeli będzie współpraca. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociażby poprzez Fundusz Dróg Samorządowych, tę rękę, a dokładniej mówiąc, miliardy złotych, wyciąga, żeby budować Polskę. I tutaj było kilkakrotnie podkreślane, że niektóre inwestycje nie są realizowane, nie są o czasie realizowane. To jest prawda i przywołana sądeczanka jest jakby najlepszym przykładem.

Szanowni Państwo! Jeszcze raz pragnę podziękować za wszystkie te inwestycje, które tutaj zostały przywołane. I tak jak mówiłam na wstępie, liczę na to, że panowie ministrowie na te pytania wszystkie odpowiedzą, uspokoją inwestorów miejscowych, uspokoją wykonawców, zapewnią, że mogą być spokojni o swoją przyszłość, uspokoją podwykonawców, którzy faktycznie mieli też ostatnio problemy. Ale też apeluję do wszystkich: zacznijcie myśleć o Polakach, a nie tylko o swoim happeningu, który tutaj dzisiaj urządziliście, bo taka destrukcja, takie wasze działania nie doprowadzą do niczego dobrego. W 2015 r. straciliście władzę i teraz tylko sztuczkami próbujecie tę władzę odzyskać. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem na plus, nie polityczne schetynówki czy inne nazwy, tylko jest rządem na plus, i Polska jest na plus. Daliśmy radę i damy radę. I liczę na to, że Polska dalej będzie się budować. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę dyskusję, bardzo żywą. Cieszę się bardzo, że inwestycje i drogowe, i kolejowe wzbudzają tak duże zainteresowanie wśród parlamentarzystów wszystkich opcji. Dziękuję też za krytykę. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi i my też się tej krytyki nie boimy, tylko dzisiaj ze strony opozycji nie było krytyki, były kłamstwa i insynuacje. Gdyby pan poseł Cezary siedział dwa rzędy niżej, to dostałbym jego nosem w twarz, tak nakłamał.

Te prace zostały wznowione za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to funkcję ministra piastuje pan minister Andrzej Adamczyk. Żeby porównać skalę inwestycji drogowych oddanych podczas pierwszej kadencji Platformy Obywatelskiej i pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, podam liczby. Liczby to jest coś, co powinno przemawiać do wszystkich. Jeżeli chodzi o drogi szybkiego ruchu, pierwsza kadencja Platformy Obywatelskiej - dokładnie 705 km nowych dróg szybkiego ruchu. To wszystko służy polskim kierowcom, to wszystko służy transportowi osób i rzeczy, to wszystko służy polskiemu społeczeństwu.

Skończymy z fragmentarycznością A1. Ta autostrada będzie niedługo służyła jako połączenie osi północ - południe wszystkim Polakom, wszystkim tym, którzy tą autostradą przemierzają Rzeczpospolitą. Kończymy z najdłuższymi schodami Europy.

Tak że te drogi po tym, jak zostaną przygotowane w pracach przedprojektowych, zostaną zrealizowane. W tym roku co najmniej 2300 zadań. To jest coś, co działa nie tylko na korzyść komunikacji, ale również na korzyść polskiej gospodarki. Bardzo proszę pana ministra Andrzeja Bittela o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To ogromne zainteresowanie infrastrukturą niezwykle cieszy, tyle że mamy do czynienia czasami z takimi ciekawymi stwierdzeniami, np. zajechaliście Y. To jest pierwsza rzecz. Czym się różnią rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u od rządów PiS-u?

Pani poseł Milczanowska wspomniała o ogromnym sukcesie rządu związanym z negocjacjami na poziomie unijnym. I my do tych wyzwań będziemy przygotowani, bo już w tej chwili mamy studia wykonalności na inwestycje o wartości 40 mld zł. Nie było studiów wykonalności. Była wielka ofensywa kolejowa, przetargi dwuetapowe, w tej chwili już niemożliwe w tym porządku prawnym, po wdrożeniu dyrektywy unijnej. Skutkiem było to, że w roku 2016 i na początku 2017 firmy biły się o zamówienia. Stąd taka firma Astaldi, która wyłożyła się na postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji. To prawda, ale potrafiliśmy szybko przywrócić tam realizację działań. Przede wszystkim potrafiliśmy rozwiązać problemy z wypłaceniem pieniędzy dla podwykonawców. Państwo tego nie potrafiliście robić. Pan poseł ma taką nieznośną manierę, by dopowiadać. Ale ja ją przyjmuję, rozumiem. Kiedyś się tego nauczę. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeśli pani marszałek pozwoli, krótko. Linia 190, wspominana, na południu. Jeden poseł coś powiedział, drugi powtórzył i mamy klasyczną manipulację. To jest linia regionalna. Ocena jej wagi należy do samorządu terytorialnego, do instytucji zarządzającej. Kropka.

W trybie sprostowania pan poseł Cezary Grabarczyk i zamkniemy ten punkt. Panowie Ministrowie! Pan poseł Matusiak minął się z prawdą.

To jest efekt starań pana ministra Nowaka, który dojechał właśnie do tego miejsca, że jest obowiązującym prawem europejskim.

Rozumiem, panie ministrze, że na część tych pytań, na które odpowiedzi nie było, posłowie będą mogli dostać odpowiedzi na piśmie. Słyszałam, że posłowie o to prosili. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 270 i 384) Proszę pana posła Kazimierza Smolińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Ma przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 270, sprawozdanie to druk nr 384.

W załączonym projekcie uchwały jest zmiana regulaminu, która dostosowuje regulamin do wymogów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15. roku życia.

Dodatkowo do komisji wpłynął wniosek, żeby dostosować zakres działania komisji do aktualnej ustawy o działach administracji państwowej w związku z tym, że powstało Ministerstwo Klimatu, a żadna z komisji takiego działu administracji nie ma w swoim zakresie działania. Komisja zdecydowała, żeby ten zakres działania, czyli klimat oraz sprawy klimatu, przekazać do zakresu działania Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która po przyjęciu zmiany regulaminu będzie nazywała się Komisją do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Kwestia połączenia klimatu i energii jest związana przede wszystkim z tym, że jest tam bardzo duża i ważna sprawa dotycząca energii odnawialnej oraz narodowego funduszu ochrony środowiska, który dysponuje ogromnymi środkami przeznaczanymi na ochronę środowiska, ale chodzi również o kwestie związane z energią odnawialną, dlatego zapadła taka decyzja. Wobec tego jeszcze raz proszę Wysoki Sejm, aby zgodnie ze sprawozdaniem komisji przyjął załączony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu zmiany regulaminu Sejmu dotyczącego dostosowania tego regulaminu do ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko seksualności i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15. roku życia, zwanej potocznie, tak funkcjonuje w opinii publicznej, komisją pedofilską. Spośród siedmiu członków tej komisji trzech członków jest zobowiązany powołać Sejm, a procedura powołania tych członków, wyłaniania ich oraz odwoływania nie ma odzwierciedlenia w regulaminie Sejmu, wobec tego należy to wprowadzić. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera przedłożony projekt zmiany regulaminu, łącznie z kwestią zmiany zakresu działania komisji sejmowej do spraw energii i aktywów państwowych, która powinna zajmować się też sprawami klimatu.

Takie wymogi w regulaminie trzeba zawrzeć. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni popierane przez klub Prawo i Sprawiedliwość. Należało również przedstawić, w jaki sposób mogą oni być odwoływani, bo jest procedura powoływania, ale również trzeba rozstrzygnąć kwestię odwoływania członków komisji. To również znalazło się w przedłożonym rozwiązaniu, jak również kwestia wyboru przewodniczącego komisji. Sejm musi dokonać wyboru takiego przewodniczącego. Jest propozycja, aby to przedstawiało Prezydium Sejmu, w którym znajdują się przedstawiciele wszystkich klubów i koła parlamentarnego.

Była również ożywiona dyskusja w zakresie tej zmiany dotyczącej zmiany zakresu działania komisji. Wiem, że będą poprawki w tym zakresie złożone, dlatego chciałbym też w imieniu klubu złożyć na ręce pani marszałek wniosek, aby nie odsyłać tych poprawek do czytania na posiedzeniu komisji, ponieważ była bardzo ożywiona dyskusja w komisji, tylko przejść do trzeciego czytania już na sali obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Ten projekt uchwały to jest jeden wielki, ogromny wstyd.

Ten projekt jest ogromnym wstydem ze względu na to, kto i kiedy go składa. Wróćmy do historii. Rok temu po emisji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” były krokodyle łzy, było bicie się w piersi. PiS zapewniał nas, że zrobi wszystko. Był projekt ustawy, przyjęliśmy ustawę zgodnie, wszyscy. Powołujemy komisję. I nic. Marszałek Kuchciński nie robi nic, marszałek Witek nie robi nic. A dzisiaj marszałek Witek kryje się za grupą posłów, którą reprezentuje człowiek od specjalnych zadań, pan poseł Marek Suski, którego zresztą - zdaje się, że nie wytrzymał - nie ma na dzisiejszej debacie. To jest problem co do tego projektu, że od września, kiedy ustawa obowiązuje, nie zrobiliście absolutnie nic w kwestii powołania tej komisji. Ale w kwestii pedofilii, owszem, zrobiliście. Bo przecież przez ten rok dowiedzieliśmy się, że oto Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez ministra Ziobrę pisze pismo do prokuratur podległych ministrowi Ziobrze, żeby w specjalny sposób traktować pedofilów w sutannach. To samo ministerstwo później pisze instrukcję: sprawy, które prokuratury rejonowe i okręgowe prowadzą przeciwko pedofilom w sutannach, należy natychmiast przekazywać do Prokuratury Krajowej, żeby tu, w Warszawie, pod okiem ministra Ziobry były rozpatrywane. To zrobiliście. Kilka tygodni temu przy ustawie COVID 3.0 dotyczącej epidemii i gospodarki, kryzysu w gospodarce zrobiliście wrzutkę, która powoduje, że praktycznie każdy może być członkiem tej komisji. Bo przecież to bardzo charakterystyczne, że wrzuciliście taki oto przepis, iż członkiem tej komisji może być ktoś, komu nadano medal lub order, i wymienia się te ordery. Za długoletnią służbę, nienaganną - to wystarczy, żeby zajmować się pedofilią? Za to, że się walczyło w Iraku i Afganistanie? O co chodzi? Co wy z tym robicie? Nie wyjaśniacie, zamiatacie pod dywan. To wszystko pokazuje, że zamiatacie pod dywan. Pana posła Suskiego tutaj dzisiaj nie ma, bo zdezerterował, ale w komisji mówił o tym, że nam zależy na tym, żeby ścigać tylko pedofilów w sutannach. Nie, nam zależy na tym, żeby ścigać wszystkich, nam zależy na tym, żeby każdy pedofil był ukarany, żeby uchronić polskie dzieci. Wy zasłuchaliście się w Toruń, w Radio Maryja i Telewizję Trwam. Wy w TVN. ...i nie słyszycie głosu prawdziwych księży, nie słyszycie głosu papieża Franciszka, nie słyszycie głosu prymasa Polaka. Co więcej, nie słyszycie nawet głosów kapłanów z diecezji kaliskiej, którzy odmówili jednoznacznie poparcia dla bpa Janiaka, bohatera drugiego filmu braci Sekielskich. To jest rok bezczynności z jednej strony, a z drugiej strony minister Ziobro wykonuje rzeczy, które mają zamieść te wszystkie sprawy pod dywan. Nie zrobiliście nic. Przez rok przez was, przez PiS cierpiały polskie dzieci.

My tutaj chcemy, aby powstała nowa komisja sejmowa do spraw klimatu. Nie może być tak, że sprawami klimatu zajmują się ci sami ludzie, którzy odpowiadają za energetykę i którym tak bardzo zależy, żeby jak najwięcej węgla w polskich elektrowniach było spalane. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Rzeczywiście ten projekt pokazuje, jak działa Prawo i Sprawiedliwość, jak działa rząd, jak działa parlament.

Od tego czasu rzeczywiście nic się nie działo. Można powiedzieć, że reagujecie dzisiaj na to, co dzieje się w mediach, na kolejny film braci Sekielskich i nagle wrzucacie temat zmiany regulaminu i, mówiąc krótko, wykonania tej ustawy, którą ta większość sejmowa przyjęła w sierpniu ub.r. Co robiliście przez ten czas? Zauważcie, co się dzieje w ogóle tutaj, na tej sali. Dyskutujemy o projektach ustaw, które np. wprowadzają przepisy i rozporządzenia Unii Europejskiej z 2009 r., jak to miało miejsce chociażby wczoraj w sprawie ustawy dotyczącej zakładów ubezpieczeń. Działacie na takiej zasadzie, żeby nie robić nic, żeby nie realizować tego, co jest wpisane w tych projektach ustaw. Ja wiem, że zaraz powiecie: rzeczywiście pandemia, rzeczywiście kryzys, było dużo ważniejszych rzeczy, dużo ważniejszych tematów, tylko że w tym czasie, przypomnę, kilkanaście razy spotykaliśmy się tutaj, na tej sali, i od 6 marca do dzisiaj, do 28 maja można było spokojnie ten projekt przeprocedować. Tego oczywiście nie zrobiono i znowu ten projekt jest procedowany po 2 miesiącach leżakowania w zamrażarce. Co się w tym projekcie pojawia? Otóż pojawia się kwestia dotycząca komisji, a więc poszerzenia, jeżeli chodzi o komisję energetyki i o sprawy związane z klimatem, ale oczywiście pojawia się też kwestia wprowadzenia do regulaminu zapisów wynikających z tej ustawy z 30 kwietnia. Tylko co się znowu dzieje? Jest oczywiście dyskusja, i tu bym apelował o to, bo akurat Lewicy bardzo zależy na wyjaśnianiu tego typu spraw, to jest jeden z fundamentalnych punktów naszego programu, zresztą w tej sprawie swój projekt ustawy Lewica również zgłosiła, w związku z czym pewnie będziemy się starali, również jeżeli chodzi o ten projekt, tzn. o tę ustawę, w jakiś sposób ją nowelizować i namawiać was do tego, drogi PiS-ie, żebyście w tym względzie pomogli, żebyście już nie zamiatali tego pod dywan. Ale widać wyraźnie, że w tych zapisach regulaminowych znowu chcecie, mówiąc krótko, trzymać wszystko w swoich rękach, bo kwestię chociażby przewodniczącego tejże komisji pozostawiacie w gestii Prezydium Sejmu. Rodzi się pytanie, czemu tylko Prezydium Sejmu ma podejmować decyzję o tym, kto będzie przewodniczącym komisji. Jeżeli chodzi o kwestię zapisów dotyczących odwołania, to tam już posłowie mogą, 35 posłów, czy powołania, czy odwołania członka komisji, to 35 posłów ma inicjatywę, ale już w przypadku przewodniczącego nie wpisujecie tego, żeby 35 posłów mogło również wskazywać kandydata na przewodniczącego. Kolejna rzecz to kwestie, które przy okazji regulaminu. I od razu sygnalizuję, że klub Lewicy za chwilę złoży te poprawki, które chcielibyśmy wprowadzić, a mianowicie chcemy wreszcie skończyć z tym bardzo złym zwyczajem, że pan marszałek Terlecki wychodzi tutaj, na tę mównicę, i mówi: To dzisiaj mam taki pomysł, blokujemy te uwagi i blokujemy poprawki senackie w dwa bloki, i sobie wszystko będziemy głosowali w dwóch krótkich głosowaniach. Chcemy to zmienić i chcemy również zaproponować przy okazji zmian w regulaminie, żeby nie można było robić tego typu rzeczy, żeby po prostu poprawki senackie były rozpatrywane na posiedzeniach plenarnych i żeby były dyskutowane, bo to jest bardzo istotna sprawa, żeby tutaj nie dochodziło w tym zakresie do manipulacji. Dlatego wnosimy te poprawki i prosimy o to, ażeby rzeczywiście przyjąć te rozwiązania, które proponujemy, i żeby ta komisja [[Dzwonek]] wreszcie po prostu zaczęła działać. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Wysoki Sejmie! Zacznę od cytatu. To jest cytat z ustawy, która została przyjęta prawie rok temu, o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Ten cytat, preambuła do ustawy, brzmi tak: Kierując się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, mając na uwadze ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu, uwzględniając powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci mimo upływu lat nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu - dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych stanowi się, co następuje. I dalej są regulacje o powołaniu komisji. Mocne słowa, wzniosłe słowa, puste słowa, tak charakterystyczne dla was, dla Prawa i Sprawiedliwości, formacji, która rządzi Polską już od 5 lat. Pamiętam, jak mówiliście 5 lat temu o tym, że państwo jest z tektury czy z dykty, państwo, które wy zbudowaliście. Celowo używam tego słowa, bo w znaczeniu słownikowym mówi ono o czymś, co jest byle jakie, kiepskie i niskiej jakości. A najlepszą ilustracją tego, jak paździerzowe jest to państwo, jest nie tylko praktyka braku tej komisji przez 9 miesięcy od przyjęcia ustawy, ale również pożałowania godny wpis jednego z waszych prominentnych ludzi, Jacka Kurskiego, który miał czelność w Internecie napisać: Nasza pedofilia jest lepsza od ich, bo nasz film oglądało więcej niż ich.

W PRL istniało takie powiedzenie: jak chcesz zamieść problem pod dywan, to powołaj komisję. Wy jesteście spadkobiercami PRL-u dokładnie w tym wymiarze. Druga sprawa związana z regulaminem ma charakter bardziej techniczny, ale jest również poważna politycznie.

Czyżby dlatego że dla was ochrona klimatu ciągle jest funkcją polityki przemysłowej, a w szczególności wydobycia, tzn. nawet nie wydobycia, tylko spalania węgla w Polsce? W planach rozwoju górnictwa w roku 2030 planujecie utrzymać je na poziomie dzisiejszym, czyli 30 t, przy czym, raz jeszcze chcę podkreślić, 20 t z tych 30 to jest węgiel importowany w największym stopniu z Rosji, ale też z Mozambiku i Ameryki Południowej. A może dlatego, że komisją środowiska kieruje polityk opozycji, a komisją energii kieruje polityk koalicji? Chcecie ukryć przed opinią publiczną, przed polskimi obywatelami, przed tak często przywoływanym przez was suwerenem prawdziwe intencje związane z polityką klimatyczną, mimo że 80% Polaków, na co wskazują najnowsze badania, domaga się radykalnego obniżenia emisji zanieczyszczeń, a rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi traci życie z powodu zanieczyszczeń, smogu i powietrza, którym nie da się oddychać.

Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Polscy politycy zrezygnowali już z mówienia rzeczy rozsądnych na rzecz ścigania się na demagogię obliczoną na łatwe podbijanie chwilowo nośnych tematów. Co więcej, w rytm kolejnych medialnych nagonek zaczęto już pisać ustawy. Legislacja to nie jest zajęcie dla ludzi o temperamencie pismaków jakiegoś brukowca, tylko dla takich, którzy potrafią chłodno analizować dane, mieć chłodny ogląd problemów i myślą na 10, 20, 100 lat do przodu, a nie o sondażu w przyszłym tygodniu. Z ubolewaniem więc stwierdzam, że Sejm raczej jest wolny od tego typu ludzi i że za ustawodawstwo zabrali się u nas raczej politykierzy, a nie mędrcy, propagandziści, demagodzy, a nie legislatorzy, czego skutkiem jest właśnie chwiejna, humorzasta mediokracja, której doświadczamy. Taka mediokracja powoduje, że ustawy w Sejmie są przyjmowane w rytm emisji kolejnych filmów w telewizji. W zeszłym roku po pierwszym filmie dostaliśmy ustawę, teraz po kolejnych dwóch filmach o pedofilii przypominamy sobie o niej i uchwalamy zmiany w regulaminie, które pozwalają na realizację tej ustawy. Jeśli kinematografia przemawia do rządzących bardziej niż fakty, to naprawdę boję się, co będzie dalej, jaką ustawę uchwalimy, jeśli np. wypuszczona zostanie kolejna część „Gwiezdnych wojen” Chciałbym się dowiedzieć, jakie liczby, statystyki powodują, że powołujemy specjalną inkwizycję poświęconą zwalczaniu akurat tego jednego rodzaju przestępstw.

Jeśli zdaniem rządzących jakiś typ przestępstw jest po prostu zbyt słabo ścigany, to należy.

Postrzeganie tego problemu jest napompowane medialnie tak jak.

To pokazuje, że media i postrzeganie subiektywne mają większe znaczenie dla państwa niż dane.

Jeśli szczerze zależałoby nam na obronie dzieci przed agresją dorosłych, to obradowalibyśmy tutaj właśnie nad zmianami w prawie, które uniemożliwiłyby bezkarną turystykę aborcyjną. Według naszego prawa wyrodna matka wydająca na śmierć swoje dziecko jest całkowicie bezkarna w tym kraju, nie ponosi żadnej kary. Przymykanie oczu na morderstwa i jednocześnie epatowanie takimi nadzwyczajnymi komisjami, trybunałami do spraw walki z pedofilią spełnia niestety wszystkie znamiona hipokryzji. Szczęść Boże! Tak jest, to hipokryzja, której Konfederacja stara się nie dzielić i nie mnożyć. Jako reżyser dokumentalista powinienem być właściwie zadowolony z tego, że emisja filmu dokumentalnego może skłonić Wysoką Izbę do tego, żeby procedowała, i to w trybie pilnym, no bo tu natłok, nawał, walka z mniemaną pandemia, a ta zmiana regulaminowa została przez prezydium skierowana na dość szybką ścieżkę. Ja się jednak z tego nie cieszę, bo właśnie słowo: hipokryzja jest najlepszą diagnozą tej sytuacji.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Ja zadam jedno pytanie. To proszę się zapisać. A teraz bardzo proszę, pierwsza jest pani poseł Monika Falej, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wprowadzenie zmiany regulaminu Sejmu podyktowane jest obowiązkiem powołania przez Sejm członków i przewodniczącego komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej 15. roku życia. Wiem, że problem pedofilii jest złożony i wymaga głównie troski o ofiarę. Zgadzam się z tym, że pedofilia nie jest. Zgadzam się z tym, że pedofilia nie jest udziałem żadnej konkretnej grupy zawodowej. To, kim jest sprawca, nie jest istotne. Istotne powinno być skuteczne przeciwdziałanie zjawisku, samym czynom i karanie ich oraz wsparcie ofiar. W tym procesie jednak dochodzi do patologii. Do komisji, o której mowa, z uporem maniaka wciąż powołuje się ludzi Kościoła, chociażby Błażeja Kmieciaka, prawnika Ordo Iuris, czyli radykalnej organizacji powiązanej z Kościołem katolickim. Fakt ten niepokoi z kilku względów.

Kolejny problem, jaki rodzi się w momencie powołania do tej komisji ludzi związanych z kościołem, to problem. Powszechnie wiadomo, że Kościół katolicki jest instytucją chronioną, jeśli chodzi o postępowania karne wobec jej członków oskarżonych o pedofilię.

Pani poseł Katarzyna Kotula, Lewica. Wysoka Izbo! Od czasu ustawy o komisji do spraw pedofilii minął prawie rok. To długo.

To projekt napisany przez prawników, konstytucjonalistów, projekt konsultowany, ale przede wszystkim projekt, który jasno i wyraźnie mówi o tym, że priorytetem jest dobro ofiar, a członkowie komisji powinni być specjalistami. Minął rok. Za nami także zmanipulowany w wielu aspektach film pana Latkowskiego, ale tak czy siak ofiary w nim ukazane były prawdziwe. O tej sprawie wiedzieli państwo od ponad 5 lat, bo było o niej głośno, a sprawcy wciąż są na wolności. Minął rok. Ponad 16 tys. ofiar pedofilii to dużo, a wy, zamiast pomagać ofiarom pedofilii (Dzwonek), skupiliście się na umieszczaniu chrześcijańskich fundamentalistów w komisji. Do tego w tarczy antykryzysowej robicie wrzutki, a przecież gdyby Prokuratura Krajowa pod rządami Zbigniewa Ziobry działała dobrze, to nie potrzeba by było żadnej specjalnej komisji. Bardzo proszę, pan poseł Marek Rutka, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z grona 38 mln obywateli i obywatelek poszukujemy zaledwie 7 osób do komisji do spraw pedofilii. W zmianach regulaminu pojawiły się zapisy, że kandydaci to osoby, które otrzymywały m.in. order lub odznaczenie, takie jak Krzyż Walecznych lub order czy medal za walkę z ustrojem PRL. Z tego katalogu wykreślono jednak osoby, które otrzymywały Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tego rodzaju zapisy noszą znamiona tworzenia ustawy pod konkretne osoby, co wzbudza nasz istotny niepokój. Dlaczego w katalogu wymogów nie uwzględniono osób o kierunkowym wykształceniu i doświadczeniu psychologicznym oraz osób, które mają bardzo wielkie doświadczenie terapeutyczne, które pracują i pracowały z ofiarami czynów pedofilskich. Pani poseł Wanda Nowicka, Lewica. Wysoka Izbo! Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego temat pedofilii znalazł się w specustawie antykryzysowej. Dlaczego w trzeciej tarczy anty-covid-owej wprowadzono art. 44, zgodnie z którym zmienia się katalog osób, które mogą otrzymać, mogą być w składzie komisji? A więc osoby, które dostaną order bądź odznaczenie, mogą być w tej komisji, ale np. straciły to prawo osoby, które mają, prawda. Można by odnieść wrażenie, że zasiadanie w tej komisji to forma synekury dla osób nagradzanych przez obecną władzę. A jeżeli połączymy to z art. 14 ustawy o państwowej komisji, który mówi, że członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją (Dzwonek) działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji komisji, wychodzi na to, że tak naprawdę chodzi o to: będzie duża kasa, niejasne obowiązki, żadnych konsekwencji. czyli innymi słowy: żyć, nie umierać w państwie PiS, oczywiście dla krewnych i znajomych władzy. Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Przed wyborami parlamentarnymi PiS przystał, uchwalił ustawę o powołaniu tej komisji, speckomisji. Przed wyborami prezydenckimi finalizujemy poprzez zmiany w regulaminie. Całe szczęście, że ten festiwal wyborczy się kończy, bo nie wiem, co by było w trzeciej kolejności, może byście państwo to wszystko odwołali zgodnie z sugestią Konfederacji. tego gmachu wyprowadziło prawo. To, jak w tej chwili procedujemy te ustawy, jest nie do przyjęcia. Ta wrzutka, ktoś tu powiedział: techniczna, to nie jest techniczna wrzutka. Do ustawy, którą większość chce, wrzuca się poprawkę, która jest z zupełnie innej parafii i czego innego dotyczy. Więc coś wam damy, trochę drobnego, trochę marchewki, ale damy też kija, a wy się teraz martwcie, jak będziecie głosowali. Chciałabym powiedzieć: Jak można (Dzwonek), jak można tak w komisji regulaminowej z łamaniem regulaminu procedować? Naprawdę, dość dużo tutaj widziałam już porządków w tej Izbie, ale takiego jeszcze nie. Pani marszałek, niejako zobowiązuję panią, bo nie jest tu pani w ogóle adresatem tego. żeby pani ten temat podniosła na następnym posiedzeniu Prezydium Sejmu. Tak nie może być. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Zbrodnia pedofilii to jedna z najobrzydliwszych zbrodni, to jedno z najobrzydliwszych przestępstw. Najlepiej świadczy o tym fakt, jak pedofilów traktuje się nawet w więzieniu. My wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jakie nieszczęście, jaka trauma pozostaje w dziecku, które jest ofiarą takiego działania. Natomiast u was jest gęba pełna frazesów, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że ustawa została przyjęta 8, 9 miesięcy temu, 8 miesięcy temu weszła w życie, a dopiero teraz robicie cokolwiek, żeby powołać tę komisję. Ja wiem, wy macie wśród siebie, nawet mieliście wśród siebie ludzi, którzy usprawiedliwiali pedofilów, jak księdza z Tylawy, pamiętamy pana posła Piotrowicza, obecnie waszego sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Dlaczego pokazaliście, że dopiero był potrzebny nowy film państwa Sekielskich, panów, braci Sekielskich, żebyście w ogóle ruszyli sprawę? Tak naprawdę nie chcecie zrobić nic. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo!

Czy my jeszcze jesteśmy normalnym parlamentem? Powstają ustawy w 2 dni, inne powinny być tworzone, powinny być tworzone bardzo szybko. I teraz pytanie do osób odpowiedzialnych: Jak ta komisja powstanie, a my ją oczywiście poprzemy, bo każdy sposób na walkę z takimi przestępstwami jest ważny, poprzemy ten projekt, czy jeśli ona powstanie, to powstanie po to tylko, żeby stworzyć kolejny pozór? Czy dalej będziecie państwo udawać, że rozwiązujecie problem i mataczyć w tej sprawie, czy wreszcie zajmiecie się rozwiązywaniem jednego z najbardziej bulwersujących problemów, które bulwersują wszystkich Polaków i Polki? Apeluję do państwa, [[Dzwonek]] byśmy zaczęli działać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

I nie chodzi mi tu za bardzo o rozszerzenie kompetencji komisji energii i skarbu państwa pod kierownictwem imperatora Marka Suskiego, którego carskie ambicje są powszechnie znane. Bardziej się martwię o komisję ochrony środowiska, którą najpierw okrojono o sprawy gospodarki wodnej, a teraz o klimat. A przypomnę, że w tym dziale, zgodnie z ustawą, są też odpady. Komisja, może dlatego, że w nazwie ma jeszcze ochronę pozostała żałosną atrapą, pozostała taką atrapą jak Ministerstwo Środowiska - do spraw myśliwych i drwali, bo tylko tyle tam zostało. Chodzi o spojrzenie przez pryzmat eksploatacji li tylko jego zasobów. Obrazują to zresztą poglądy ministra.

Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście nie ma w słowniku ludzi kulturalnych wystarczająco mocnego słowa, żeby określić w sposób adekwatny przestępstwo pedofilii.

Sprawa została odłożona na półkę i w sposób haniebny wykorzystana podczas okresu wyborczego. Została zostawiona aż do momentu, kiedy pojawił się kolejny film. Tego nie można określić żadnym słowem, które znajduje się również w słowniku ludzi kulturalnych. Po prostu nie można. Na dodatek dzisiejsza wrzutka. Wrzucacie do regulaminu Sejmu przepis, który spowoduje, że przewodniczącego komisji wybierze de facto PiS. Kogo wy tam chcecie postawić? Przez rok daliście nam wszystkim świadectwo, że waszym jedynym celem jest to, żeby tę sprawę rozmasować, ukryć, rozpuścić, [[Dzwonek]] żeby pozostawić ofiary same, a tych, którzy byli sprawcami, przykładnie odsunąć od oczu opinii publicznej. Kogo chcecie postawić na czele tej komisji? Proszę tu przyjść i powiedzieć Polakom: Kogo? bardzo, panie pośle. Pan poseł Michał Szczerba.

Myślę, że miejsce na zabranie głosu jest przede wszystkim na mównicy sejmowej, więc do tego zachęcam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Niestety ten projekt trafił do niechlubnej sejmowej zamrażarki, mimo naszych próśb i apeli.

Ten niezwykle ważny i wielowątkowy temat, który obejmuje swoim zakresem zarówno kwestie energii, jak i rolnictwa, ochrony środowiska, a także infrastruktury i gospodarki, potraktowano tak naprawdę jak kwiatek do kożucha. Dlatego składamy odpowiednie poprawki. I tu moje pytanie do wnioskodawców:

Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Tu padło pytanie o kandydatury na przewodniczącego tej komisji. Wtedy bracia Rysicz i przyjaciele mogliby być zawezwani jako eksperci w tej dziedzinie. Pytanie: Kiedy ruszycie ze sprawą projektu „Stop pedofilii” Czy ukonstytuowanie się tej komisji w takim trybie akcyjnym będzie znamionować otwarcie nowego rozdziału i przejście do działań realnych ze strony służb prokuratorskich, policyjnych, ale także ze strony parlamentu, który powinien projekt „Stop pedofilii” wyjąć z tej de facto zamrażarki i skierować na normalną ścieżkę legislacyjną? Czy wśród ekspertów tutaj już z góry odsądzanych od czci i wiary znajdą się i tacy, którzy nie będą się wahali wskazać związku łatwego do wykazania poprzez nadreprezentację statystyczną osób hołdujących innym zboczeniom o charakterze homoseksualnym w grupie nazywanej pedofilami?

Pani Marszałek! Mam zasadnicze pytanie dotyczące omawianej dzisiaj komisji do spraw pedofilii, która dopiero zostanie powołana. Mam nadzieję, że nie jest to tylko przykrywka. Powinna ona nastąpić natychmiastowo. Widzieliście państwo wszyscy twarze tych cierpiących dzisiaj mężczyzn, te zniszczone życiorysy i poszarpaną psychikę, a ofiar jest zapewne dużo więcej. Dlatego pilnie dopytuję o opracowanie harmonogramu pracy komisji, ustalenie jej członkostwa oraz dokładnego terminarza jej pracy. Mam nadzieję, że nie będzie ona, tak jak każda powoływana w tej Izbie komisja, słono opłacana ze środków podatników. Mam również nadzieję, że presja społeczna, która dzisiaj jest przecież ogromna, doprowadzi do tego (Dzwonek), że wreszcie winni zostaną ukarani, a sprawiedliwości stanie się zadość. Bardzo proszę sprawozdawcę komisji pana posła Kazimierza Smolińskiego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szkoda, że większość tej debaty niestety nie skupia się na przedmiocie przedłożenia, czyli zmianie regulaminu, tylko na ustawie, która została już przyjęta przez Sejm i nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Ale w związku z tym, że tyle było wokół tego pytań różnego rodzaju i dywagacji, pozwolę sobie też do tego się odnieść. Lewa część sali niestety ma usta pełne frazesów, ale jak przedłożyliśmy rozwiązanie, które niewątpliwie pomaga w walce z pedofilią, czyli rejestr pedofilów, państwo byliście przeciwni. Nie zagłosowaliście za tym. I ciągle mówicie tylko: 8 miesięcy, 8 miesięcy. A ja mówię: 8 lat. Co przez 8 lat zrobiono w zakresie walki z pedofilią? Następnie rozpowszechnialiście państwo nieprawdziwe informacje związane z tym, że w tym rejestrze nie są uwzględnieni księża. Przecież to jest nieprawda. Od początku ten rejestr w tym zakresie był jawny i obejmuje wszystkich - wszystkich. Oczywiście. To jest kwestia właśnie zrozumienia i czytania ze zrozumieniem ustawy, każdej, i tej zasadniczej, w postaci konstytucji, którą nie trzeba wymachiwać, tylko trzeba stosować, i każdej innej ustawy. Ta ustawa stanowi dla nas obowiązek, żebyśmy wybrali trzech przedstawicieli, nie tylko przedstawicieli Sejmu, bo będą tutaj kandydaci zgłoszeni przez Naczelną Radę Adwokacką, naczelną radę radców prawnych i wszystkie inne organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw dzieci czy ochroną osób poszkodowanych. Każda z tych organizacji może złożyć propozycję co do swojego kandydata. Po to jest regulamin. Proszę państwa, pani marszałek powiedziała czy też pan marszałek Terlecki powiedział, że w tym tygodniu. Niestety w tym tygodniu nie zdążymy tego zrobić, ponieważ dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj, przegłosujemy tę zmianę regulaminu, a gdy zostanie ogłoszona, gdy wejdzie w życie, niezwłocznie, następnego dnia pani marszałek musi ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej, że organizacje uprawnione z tej ustawy mogą zgłaszać kandydatów, i wyznaczy termin na zgłaszanie tych kandydatów.

Jestem przekonany, że to będą osoby o dobrym przygotowaniu, o właściwych kompetencjach, osoby, które będą chciały walczyć z pedofilią, którą, myślę, wszyscy na tej sali oceniamy jednoznacznie - tak jak tu niektórzy powiedzieli, brak słów na ocenę tych przestępstw. Tak że nas nie trzeba przekonywać do tego, że to ohydne przestępstwo musi być ścigane. Tu przede wszystkim komisja ma wspierać organy państwa, prokuraturę. I w tym zakresie nie ma żadnych świętych krów. Czy to będzie środowisko kościelne, czy to będzie środowisko polityków, czy to będzie środowisko nauczycieli, obojętnie, wszyscy są tak samo traktowani. Nie ma świętych krów w tym zakresie.

Dzisiaj nawet padły te słowa, że w tym filmie to już są manipulacje, że w tym zakresie są manipulacje. A statystyka jest właśnie inna. Nie chodzi tu o statystykę, bo każde przestępstwo jest takim samym dramatem jak tysiące innych. I będą wszystkie te przestępstwa zwalczane, jestem przekonany co do tego, w taki sam sposób. To jest kwestia tylko tego, ile czasu pani marszałek da tym organizacjom na zgłaszanie kandydatur. Myślę, że nie będzie to długi czas. Organizacje są przygotowane do tego, żeby zgłaszać te kandydatury, więc teraz czekamy.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Przypominam, że był pan sprawozdawcą komisji. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania po doręczeniu zestawienia poprawek. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej panią Barbarę Sochę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Przepraszam bardzo. Ale tutaj miałam napisane.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Opieka nad dziećmi do lat 3 to jest jeden z ważniejszych kierunków działań rządu, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Program „Maluch+” to jest obok innych wiodących programów rządu Zjednoczonej Prawicy ważny element. W tej chwili pracujemy nad strategią demograficzną i mogę powiedzieć, że po pół roku pracy jesteśmy bardzo na bieżąco ze wszystkimi badaniami naukowymi dotyczącymi wpływu różnych czynników na dzietność.

Ustawa „Maluch+” jest właśnie realizacją takiej polityki.

Jedną z zasadniczych zmian, które już w 2018 r. obowiązywały, była możliwość zakładania żłobków przez podmioty prywatne, nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego. To bardzo wpłynęło na dynamikę liczby miejsc.

Podnieśliśmy również standardy co do wyżywienia dzieci. Jak wspomniałam, została poszerzona lista podmiotów, które mogą tworzyć i prowadzić żłobki, i było szereg innych zmian. Myślę, że jedną z najważniejszych były zwiększone nakłady na tego rodzaju inwestycje i wprowadzenie różnych modułów, zgodnie z którymi szczególnie gminy czy obszary, w których nie było do tej pory takich placówek, mogły korzystać z uprzywilejowanych form wsparcia na tworzenie żłobków, co powoduje, że znacząco wzrasta liczba gmin, gdzie te żłobki się pojawiają, rośnie liczba miejsc.

To jest bardzo duży wzrost na przestrzeni poprzednich kilku lat. Oczywiście nadal program „Maluch+” będzie rozwijany. Pracujemy nad kolejnymi zmianami, które spowodują, że jeszcze więcej żłobków będzie powstawało. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, myślę, istotny w momencie, kiedy rozmawiamy o opiece nad dziećmi do lat 3. Żłobki są ostatnim preferowanym przez polskie rodziny sposobem opieki. W moim przekonaniu zbliżamy się do.

Myślę, że szczególnie gdy rozpoczyna się debatę, liczę na taką debatę nad strategią demograficzną, będzie okazja, żeby rozmawiać o rozwijaniu innych form opieki nad dziećmi, jako że te inne formy opieki są bardziej preferowane przez rodziców w Polsce. Posługuję się tutaj nie swoimi przekonaniami, tylko danymi statystycznymi i badaniami prowadzonymi przez różne jednostki. Z tych najświeższych dysponujemy badaniami CBOS-u na ten temat. Kolejne badania, przygotowywane dokładnie pod konkretną operacjonalizację strategii demograficznej, są w tej chwili w trakcie i myślę, że do końca roku będą zrealizowane. Witam serdecznie państwa. Pan poseł Borowiak, zapraszam. Pani poseł, przepraszam. Proszę bardzo. W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiam sprawozdanie o sprawozdaniu Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r., druk nr 83. Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 223. Na posiedzeniu 11 lutego 2020 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła przedłożony dokument. Przeprowadzono dyskusję, posłom zadającym pytania zostały udzielone odpowiedzi. W efekcie prac nad tym dokumentem za przyjęciem sprawozdania głosowało 17 posłów, przeciw - 1, wstrzymało się 4. Wobec powyższego Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wnosi do Wysokiego Sejmu o przyjęcie sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Zapraszam serdecznie panią poseł Teresę Wargocką z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. Priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy jest prowadzenie polityki nakierowanej na wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Obok wsparcia finansowego rodzin w programach 500+, 300+ dużą wagę przykładamy do rozszerzenia zakresu wsparcia w formie organizacji instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Formy tej opieki są bardzo zróżnicowane.

W dyskusji na temat opieki i wychowania dzieci najmłodszych spotykamy się z różnymi poglądami. Środowiska lewicowo-liberalne promują model pełnej opieki instytucjonalnej, a środowiska skrajnie prawicowe przekonują o szkodliwości dla rozwoju dzieci powierzania opieki nad nimi osobom innym niż członkowie rodziny. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku absolutnego poszanowania autonomii rodziny. Chcemy, by wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci do lat 3 było adekwatne do oczekiwań rodziców i nie stanowiło bariery przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu potomstwa. Jesteśmy społeczeństwem, w którym wartości rodzinne są stawiane na najwyższym miejscu, jednocześnie potrzeba samorealizacji, aktywności zawodowej, niezależności finansowej jest cechą postaw podzielanych przez wiele kobiet. Z badań wynika, że młodzi małżonkowie oczekują od władzy publicznej stwarzania jak najlepszych rozwiązań godzących pracę zawodową z macierzyństwem. Stanęliśmy po stronie rodziców w sprawie wprowadzanego przez Platformę i PSL obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Znieśliśmy obowiązek edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich. Tutaj też rodzice mogą wybrać i chętnie tę edukację wybierają. Ale wybór jest najważniejszy. Prawo i Sprawiedliwość szanuje autonomię rodziny, jednocześnie wsłuchuje się w oczekiwania rodziców. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 jest dobrą ustawą. Przyjęta w 2011 r. ponad politycznymi podziałami jest sukcesywnie realizowana poprzez rządowe programy „Maluch”, a obecnie „Maluch+” Ten „+” pozwolił bardziej zdynamizować rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Trzykrotne zwiększenie środków finansowych na program, do kwoty 450 mln, poszerzenie zakresu podmiotów, które mogą z tego programu korzystać poprzez sektor prywatny, dofinansowanie kosztów utrzymania miejsca w żłobku - to są zmiany, które w 2018 r. pozytywnie przyczyniły się do osiągnięcia dobrych rezultatów i powiększenia liczby miejsc w żłobkach o ok. 19%. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w dużej mierze realizowana jest przez podmioty prywatne, a nie jednostki samorządu terytorialnego. W 2018 r. samorządy utworzyły 760 żłobków, co stanowi 24%, i tylko 46 klubów dziecięcych, co stanowi 7% wszystkich utworzonych klubów. 62% samorządów nie ma zorganizowanej jakiejkolwiek opieki nad dziećmi do lat 3. Dane te świadczą o dużej rozbieżności pomiędzy polityką prorodzinną państwa a realizacją zadań własnych przez samorządy. Tak jak wspomniałam na wstępie, liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powinna być skorelowana z potrzebami społecznymi rodziców na danym terenie - ani większa, ani mniejsza. To samorząd terytorialny powinien diagnozować te potrzeby i adekwatnie je zaspokajać, korzystając z rządowego wsparcia, chociażby takiego jak program „Maluch+” Z danych ministerstwa rodziny, które zebrało informacje o liczbie osób oczekujących na listach rezerwowych na miejsca w placówkach opieki nad małymi dziećmi, wynika, że to zapotrzebowanie jest nadal duże i na koniec 2018 r. wynosiło ponad 70 tys. miejsc. Tak więc zadanie wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3 jest zadaniem ciągłym. Oczekiwane jest większe zainteresowanie samorządów prowadzeniem polityki prorodzinnej na szczeblu gminy. Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał wszystkie propozycje rządu mające na celu wsparcie rodzin (Dzwonek) zgodnie z ich oczekiwaniami. Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za przyjęciem informacji. Zapraszam panią poseł Aleksandrę Gajewską z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo też muszą wybrać, w jaki sposób pojmują politykę prorodzinną: czy państwo stoją za tym, żeby Polska była Polską socjalną, czy Polską społeczną. To jest zderzenie pewnych wizji.

Tak, jest program 500+, to jest ważny program, ale to jest program, który nie stanowi systemowego rozwiązania prorodzinnego. On przede wszystkim nie spełnia założenia demograficznego, bo to, że zostały przekazane te środki, w żaden sposób nie wpłynęło na zwiększenie dzietności w Polsce. Program, na temat którego słuchamy dzisiaj sprawozdania, też nie jest państwa systemem, tylko to jest system, który został wprowadzony przez rządy Prawa. Państwo dodali do tego słowo „plus” Państwo to kontynuują, co ja pochwalam, ale nie w sposób doskonały. Nie w sposób doskonały, właśnie dlatego że państwo zmienili te standardy, które były wprowadzone przez PO i PSL. Państwo je zmienili w taki sposób, że protestowali rodzice, protestowali pracownicy.

To pozwalało na godzenie obowiązków zawodowych z bardzo ważnym życiem rodzinnym. Wprowadziliśmy też dofinansowanie dla niań, państwo to potem obcięli o połowę. Ja się zastanawiam, co państwo traktują w tym programie jako plus. Bo państwo sobie w pewien sposób tutaj też przypisują zasługi samorządów. To polskie samorządy tę ciągłą funkcję realizują i to samorządy robią to właśnie w sposób najlepszy. I za te działania tym samorządom należy podziękować, zwłaszcza że wczoraj obchodziliśmy 30-lecie polskiej samorządności. Ja byłam prawie 9 lat radną Warszawy i Warszawa jest najlepszym przykładem, że można realizować taką politykę prorodzinną dobrze, mądrze i skutecznie. 13 tys. miejsc. jeżeli pani pyta, już pani odpowiadam, opieki nad dziećmi do lat 3. W zeszłym roku utworzono 5252 nowe miejsca. Warszawa wydaje na ten cel więcej niż rząd w skali kraju. 344 mln na politykę prorodzinną. Co to jest? 160 mln dajecie dotacji dla brata pana ministra Szumowskiego, 214 mln dostaje Radio Maryja. Państwo wspierają rodziny, ale rodziny ministrów i rodziny Radia Maryja, a nie rodziny, które rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Tylko co dzieje się. Bo my możemy mówić o większych miastach, ja akurat mam takie doświadczenie z Warszawy, w której prezydent, zarząd miasta, urzędnicy doskonale radzą sobie z tymi zadaniami, ale co z biedniejszymi, mniejszymi gminami?

Właśnie na tym polega różnica między nami a państwem, że my te samorządy traktujemy po partnersku. Badamy usługi żłobkowe, w klubikach itp. i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców, tak żeby było coraz bardziej elastycznie i żeby rodzice mogli się realizować. A więc państwo powinni przekazywać więcej środków samorządom i odejść od tych złych przepisów, które pozwalają na to, żeby coraz więcej dzieci upychać w [[Dzwonek]] coraz mniejszych salach. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią posłankę Darię Gosek-Popiołek z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Pani Minister! Rozmawiamy dziś o tym, jak państwo wywiązuje się ze swojego obowiązku zapewnienia opieki nad rodzinami, nad dziećmi do lat 3. A więc takie szybkie pytanie: Kiedy możemy liczyć na to, że ten raport, sprawozdanie za rok 2019 trafi do naszych rąk? Ale wróćmy do tego sprzed 2 lat już tematu. Chwali się pani minister wzrostem liczby miejsc w żłobkach, ale powiedzmy uczciwie, z czym się to wiąże. Od 2018 r. wystarczy, że w żłobku będzie jedno pomieszczenie dla dzieci. Zmniejszono także wymaganie, jeżeli chodzi o metraż, jaki przypada na jedno dziecko.

Te białe plamy to są samorządy, w których nie ma żłobków - ani państwowych, ani prywatnych. Po prostu ich nie ma. Oczywiście, ale spójrzmy na te liczby. Zaledwie 22% gmin zgłaszało potrzebę utworzenia większej liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, ale te gminy to są generalnie gminy, w których już te żłobki i przedszkola są, więc jest tam sytuacja całkiem niezła. To oznacza, że na wsiach, w mniejszych miastach, w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich po prostu żłobków i klubów dziecięcych nie ma. Tam rodzice, matki są pozostawieni sami sobie. i jeżeli ktoś chce łączyć życie zawodowe z wychowywaniem dzieci, właściwie nie może liczyć na wsparcie państwa. Z tego sprawozdania nie dowiemy się także o sytuacji żłobków dziś i o tym, co będziemy robić.

Nie wiemy, co będzie, gdy zmuszone brakiem finansów gminy zmniejszą dotacje na żłobki. Nie dowiemy się, co będzie z dziećmi, które do żłobków nie pójdą, nie wrócą do nich bądź w ogóle tam nie pójdą, dlatego że ich rodzice albo stracili pracę, albo muszą borykać się z tak radykalnym zmniejszeniem zarobków, że ich po prostu na to nie będzie stać. A więc teraz widzimy, że ten system, który państwo opracowali wiele lat wcześniej, po prostu nie działa. O tym, że nie działa, mówią nam rodzice, ci rodzice, którzy z nami się kontaktują i mówią, że dla ich dziecka nie ma miejsc w żłobku publicznym, a prywatny kosztuje 1200 zł. O tym, że system nie działa, wiemy od rodziców, których państwo polskie zmusza, aby kalkulowali, czy w obliczu pracy na śmieciówce bądź pracy za najniższą krajową opłaca się im posłać dziecko do żłobka. O tym, że system nie działa, wiemy od kobiet, od matek, które nie mogą wysłać swoich dzieci do żłobka, ponieważ nie mogą teraz pójść do pracy, nie mogą rozpocząć aktywności zawodowej. Będą mieć głodowe emerytury. I wtedy to państwo, które wy tak ułożyliście, przyjdzie i powie im: nie, nie. Panie nie dostaną wysokiej emerytury. Panie nie pracowały. Cóż z tego, że one wykonywały ciężką pracę, skoro państwo tego nie rozpoznaje i nie chce im pomóc? To jest ten moment, kiedy widzimy, że to nie działa, i zróbmy, szanowni państwo, coś, czego to państwo nigdy w życiu jeszcze nie zrobiło: wyciągnijmy wnioski. Wyciągnijmy wnioski. Skoro pomimo milionów, pomimo silnych samorządów, które starają się zapewnić miejsca w żłobkach, to nie działa, zmieńmy ten system. Państwo powinno w znaczący sposób wesprzeć gminy w tworzeniu żłobków czy klubów dziecięcych za pomocą subwencji, tak, subwencji, na kształt subwencji oświatowej, nie jakichś tam dotacji, które raz są, a raz ich nie ma. Żłobki to nie luksus, to nie biznes, by powstawać tylko tam, gdzie to się komuś opłaca. Są potrzebne także w mniejszych gminach. To element systemu, tak samo jak szkoły czy przedszkola. Zadbajmy o pensje i warunki zatrudnienia osób, które zajmują się naszymi dziećmi w żłobkach. To trudna i wymagająca praca. Zupełnie nie widzę powodu, dla którego praca opiekunek w przedszkolach, w żłobkach ma być inaczej wynagradzana (Dzwonek) niż praca nauczycielek w przedszkolach czy szkołach. Żłobki to nie tylko dobrze zaopiekowane dzieci. To szczęśliwe rodziny, to matki, które mogą się realizować, to ojcowie, którzy mają spokój w głowie. Dobrze urządzona, zaopiekowana i mądra Polska zaczyna się w żłobku. Dziękuję serdecznie.

Ale przyznam się szczerze, że mam ogromny niedosyt i być może nawet pretensje do siebie, że szło to tak wolno.

Państwo mówicie o tym, pani minister dzisiaj, że opieka żłobkowa nie jest preferowana przez rodziców i że są jakieś inne formy opieki, które są jakoby lepsze, co wynika z badań, które państwo przeprowadziliście, natomiast w strategii do 2030 r. mówicie, że liczba tych miejsc ma wzrosnąć do 30%. To, proszę państwa, jest naprawdę bardzo, bardzo mało.

Chciałabym zwrócić uwagę na to, że kiedyś konserwatywne wychowanie to było wychowanie dzieci w wielodzietnej rodzinie. Dzieci wychowywały się wśród licznego rodzeństwa. Dziś, kiedy mamy jedno dziecko w rodzinie, naprawdę absolutnie dobrze mu zrobi, jeżeli na jakiś czas będzie ono zaopiekowane właśnie w takich formach, gdzie będzie miało towarzyszy zabaw. To będzie dla niego bardzo dobre i nie ma to nic wspólnego z tym, czy mówimy tu o konserwatywnym, czy lewicowym sposobie wychowywania. Dlatego bardzo jestem rozczarowana tym, że idzie to tak wolno. Chciałabym zwrócić jednak uwagę, że być może idzie to tak wolno dlatego, że te formy opieki, które państwo w tym sprawozdaniu umieszczacie, są po prostu zbyt, powiedziałabym, trudne dla tego dziecka, zbyt niedoskonałe, mianowicie sporo dzieci pod opieką wychowawczyni, niewielkie sale, oszczędności na dzieciach.

Chciałabym też zwrócić uwagę na samo sprawozdanie.

Dlatego dziwi to, że państwo opóźniacie przedstawienie tych sprawozdań.

Chciałabym zwrócić uwagę, że polityka prorodzinna powinna być absolutnie priorytetem państwa, ponad wszelkimi podziałami. Dlatego cieszę się, że ten program „Maluch+” lepiej czy gorzej jest dalej realizowany. Mam nadzieję, że liczba miejsc w żłobkach, i to dobrych miejsc, takich miejsc właśnie, które będą dobre dla dzieci, będzie po prostu większa, czego sobie i państwu życzę. Dziękujemy za życzenia. Prosimy w tej chwili pana posła Krzysztofa Tuduja z koła Konfederacji. Pan poseł nadchodzi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po pierwsze, w tej debacie warto ukłonić się wszystkim rodzinom, dzielnym Polakom, którzy nie rezygnują z posiadania dzieci, nie rezygnują dla kariery, dla jakiegoś pędu ekonomicznego.

Rolą państwa jest nie przeszkadzać. Dobrze, że w tym przypadku tych opcji jest kilka, jest wiele.

Nie punkcik, nie żłobki, tylko kompleksowy programu polityki prorodzinnej, który szeroko, mocno i skutecznie odpowie na wyzwania związane z demografią. Trzeba pamiętać, że to jeden z dwóch, trzech najważniejszych problemów, przed jakimi stoimy. Tak że zachęcam i apeluję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Panie Marszałku Czcigodny! Kontynuując wątek podjęty przez mojego kolegę posła Tuduja, powiem wyraźnie i zdecydowanie: żeby w ogóle były jakieś dzieci w Polsce, o których los można by się troszczyć, broniąc je przed przestępczością zorganizowaną i niezorganizowaną - przez przestępczość zorganizowaną rozumiem oczywiście gangi pedofilów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest przestępczość zorganizowana, działanie na szkodę dzieci wspólnie i w porozumieniu przez rozmaite mafie, służby i loże, które dokonały już dawno wrogiego przejęcia projektu polskiej państwowości - żeby w ogóle można było dzieci bronić, troszczyć się o nie, to one się muszą urodzić. W związku z tym sprawozdania tego typu, ta sprawozdawcza radosna twórczość biurokratyczna to jest jeden nieustający pokaz hipokryzji w sytuacji, gdy życie, samo życie, bezpieczeństwo życia ludzkiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest prawnie gwarantowane.

Pierwszy raz w najnowszych dziejach politycznych Rzeczypospolitej, bo za dawnych czasów o takich oczywistych oczywistościach na szczęście na forum publicznym nikt nie dyskutował, dzieciobójstwo było dzieciobójstwem i tyle. Ale od kiedy się o tym dyskutuje, pierwszy raz w dziejach Rzeczypospolitej trzeciej i pół mamy, zdawałoby się, oczywistą, gotową, gwarantowaną większość parlamentarną za życiem. Bo kto z was, koleżanki i koledzy z tej strony sali, ze strony jedynie słusznej większości, Prawo i Sprawiedliwość z przystawkami, publicznie wyprze się, zaprze i wykręci w tej sprawie? Kto z was powie otwarcie, że nie jest za życiem? Głosy Konfederacji są gwarantowane. 11 głosów za. Kiedy trzeba było tutaj głosować w sprawie projektu przeciwko aborcji eugenicznej, naszych 11 dłoni podniosło się w górę. Ale także i w sąsiednich klubach znajdą się tacy, co może lekko się konspirują, może się z tym nie afiszują, ale przecież nie będą przeciw. I otóż wyłącznie wola polityczna, a raczej jej brak, zaniechanie po stronie aktualnego układu rządzącego, sprawia, że bezpieczeństwo życia ludzkiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest gwarantowane. Wykorzystuję te chwilę, żeby wezwać was, władzo, rządzie, prezydencie belwederski, i was, większości parlamentarna z prezesem, premierem i naczelnikiem żoliborskim na czele: zagwarantujcie bezpieczeństwo życia ludzkiego, a potem zajmijcie się spisywaniem raportów, w których. Tam jest mowa o kwalifikacjach, jakie muszą mieć te osoby, które się zajmują dziećmi. I tam jest wszystko: jest wyższe wykształcenie, aż do tytułów naukowych, tam są kwalifikacje, doświadczenie.

Zagwarantujcie bezpieczeństwo życia ludzkiego. To przejdzie do historii, to otworzy nową kartę w dziejach Polski. Dziękuję w imieniu dziadków, panie pośle. Proszę państwa. Dziękuję serdecznie, panu też tego życzę. Wcześniej czy później dojdzie pan do takiego stanu. Proszę państwa, zaczynamy. Pracuje pan? Gdyby pan chciał wiedzieć, jak to się robi, służę pomocą. Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań.

Zapraszam pierwszą osobę, panią posłankę Wandę Nowicką z klubu parlamentarnego Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministro! Program rządowy, który jest opisany w sprawozdaniu, dalece nie satysfakcjonuje.

W związku z tym trudno się dziwić, że efekty tego programu rządowego są, jakie są. Panie marszałku, mogę prosić o interwencję? Ja przepraszam, przepraszam. Ja mam do pani taką prośbę, pani poseł. Nie przerywajmy sobie, bo pójdę po marszałek Witek, a ona panią ukarze. Tak mi dzisiaj powiedziała, [[Dzwonek]] że jak ktoś będzie przerywał, to mam po nią pójść, ona przyjdzie i będzie karała.

Proszę bardzo, pani posłanka Nowicka. Dziękuję, panie marszałku, za interwencję. Tak, trudno być zadowolonym z programu, na który przeznaczyliśmy tak małe pieniądze. I to wynika oczywiście ze sprawozdania rządowego. Natomiast czego brakuje w tym sprawozdaniu? Jakiejkolwiek analizy, dlaczego jest tak źle, kiedy niby jest dobrze. Proszę państwa, w województwie śląskim dostępność miejsc w żłobkach jest na poziomie 17%. To jest naprawdę bardzo niewiele. W Gliwicach - miasto w końcu duże - też są ogromne problemy z opieką żłobkową. Proszę państwa, ja nie kupuję takiej opowieści, że winne są temu samorządy. Od rządu oczekuję, żeby przedstawił analizę, dlaczego np. samorządy nie są w stanie zbudować więcej żłobków. Widocznie dajecie za mało pieniędzy albo te pieniądze są źle adresowane. Zastanówcie się nad tym, co możecie zrobić, żeby tę sytuację poprawiać. Bo to, że jest dobry rząd, który daje, i zły samorząd, który celowo nie chce budować żłobków, to jest nieprawda. To jest obraźliwe stwierdzenie pod adresem samorządów i takich argumentów nie możemy przyjąć. A zatem weźcie się do roboty i zróbcie wszystko. Przede wszystkim dajcie więcej pieniędzy, dobrze adresowanych.

Dziękuję serdecznie.

Nie wyłącza mikrofonu. Wszyscy będą mówili. Proszę o cudowne zgłoszenia.

Pani Minister! Wysoki Sejmie!

Bo jeśli popatrzymy na ten raport, z którego wynika, że w 21% gmin wiejskich mamy tylko jedną z instytucji opieki nad małymi dziećmi. To jest podstawowy problem. Po drugie, mamy też zróżnicowanie terytorialne.

Ci, którzy chcą, wiedzą, jak to zrobić, i mają pieniądze, chcą uruchomić.

A co dalej? A co z wieloletnią prognozą finansową? Dziękuję. Pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że w rządowych opracowaniach jako barierę utrudniającą podejmowanie decyzji o powiększeniu rodziny i posiadaniu dzieci wskazano niemożność łączenia życia rodzinnego z pracą. Zauważenie kwestii oczywistych dla Lewicy to postęp umożliwiający wprowadzenie rozsądnych polityk interwencji.

Dla samorządów niepubliczna opieka nad dziećmi do 3. roku życia jest tańsza niż budowanie i utrzymywanie nowo budowanych żłobków publicznych. Pytam zatem o wnioski ze sprawozdań. Jak chcecie zapewnić stałość wsparcia tych podmiotów niepublicznych, które nie raz i nie dwa doświadczały wycofywania wsparcia umożliwiającego zachowanie płynności finansowej?

Czy planujecie zmiany w rozliczaniu programu „Maluch+” Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Katarzyna Kotula, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo!

Podobnie wygląda to w Krakowie i we Wrocławiu. To oczywiście koszty z uwzględnieniem posiłków.

Opłata za wyżywienie to jest 7 zł. Łatwo policzyć, że nawet 500+ na opłatę nie wystarczy. Chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam dorosłą już córkę, bo mogę powiedzieć z całą stanowczością, że na żłobek nie byłoby mnie stać. Martwię się faktycznie, co będzie, kiedy zostanę babcią, i czy nie będę musiała jednak do tego dokładać. Oczywiście mamy świadomość dotacji, innych programów socjalnych i wszelkiej pomocy, którą oferujecie. Chciałabym jednak zapytać, czy macie świadomość - bo nie znalazłam nic o tym w raporcie - że dofinansowanie nie pokrywa opłaty wpisowej w żłobku, która wynosi między 300 a 500 zł. Jest to dosyć wysoka kwota. Może okazać się, że będzie potrzebna pożyczka na zapisanie dziecka do żłobka. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Paulina Matysiak, klub parlamentarny Lewica.

Pani Minister! Wysoka Izbo! Zgodnie z raportem liczba miejsc w żłobkach wzrasta, ale dlatego że większość nowych miejsc to miejsca prywatne. Przedstawicielka ministerstwa mówiła wprost, że utworzenie miejsc w żłobkach prywatnych jest tańsze niż w państwowych, dlatego rządzący idą w tę stronę. To nie jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza w okresie kryzysu, gdy dochody wielu rodzin drastycznie spadły bądź drastycznie spadną i nie będzie ich stać na prywatną placówkę. Nieodpłatne miejsce w publicznym żłobku powinno czekać na każde dziecko, powinno być prawem, a nie towarem, i to już nawet nie ze względu na rodziców, ale ze względu na prawa dzieci. Konsekwencje prywatyzacji doskonale widać teraz w wielu branżach. Dostępność usług publicznych staje się przywilejem prywatnym, kiedy w związku z obostrzeniami wiele dzieci nie może wrócić do żłobka, bo brakuje miejsc. Skoro jest tak dobrze, jak przedstawia to raport, to czemu dzieci z Bródna, czemu dzieci z Żoliborza czy z innych zakątków Polski ciągle nie mogą wrócić do żłobka (Dzwonek), tylko muszą zostać z rodzicami w domu? Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po raz kolejny rozmawiamy o raporcie za 2018 r. w maju 2020 r. Bo niby dlaczego mamy czekać praktycznie 2 lata na to, żeby rozmawiać o takim raporcie? W moim rodzinnym mieście, w Jeleniej Górze, jest jeden żłobek prowadzony przez samorząd.

Jestem tego przeciwnikiem i uważam, że powinniśmy wesprzeć samorządy po to, żeby te samorządy mogły budować żłobki, ale też je utrzymywać. Myślę, że to nie przypadek, że 7 października były minister ochrony środowiska (Dzwonek), już niestety nieżyjący, podsumował politykę w stosunku do żłobków. Powiedział, cytując: Nie trzeba pomagać w sposób sztuczny w budowie żłobków, przedszkoli, tych innych rzeczy. To są sprawy chwilowe, jako spuścizna po poprzednim systemie komunistycznym. Dziękuję. Pan poseł Paweł Krutul, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do przedstawionego raportu można mieć wiele zastrzeżeń: co do jakości, co do sposobu prezentowanych liczb, co do ostrożności autorów w ich prezentacji. Jednak to, co rzuca się w oczy, to fakt, że rząd, ten sam, który mówił tyle o bezpieczeństwie rodzin w 2018 r., przeznaczył na żłobki 500 mln zł. Tak jak pani marszałek powiedziała, tyle samo państwo przeznaczyliście na obraz „Dama z łasiczką”

Mamy przygotowane rozwiązania i zachęcamy do korzystania z nich. Na początek możecie państwo zrezygnować z zakupu przykładowo samolotów szturmowych F-35 i zainwestować w naszą przyszłość, w nasze dzieci. Dziękuję serdecznie. Proszę panią posłankę Monikę Falej z klubu parlamentarnego Lewica. A jeżeli jej nie ma, to poproszę panią posłankę Karolinę Pawliczak. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Nie twierdzę, że w sprawie opieki żłobkowej przez lata nic nie zrobiono, bo sytuacja na pewno się poprawiła.

Pozostaje jednak pytanie: Czy można zrobić coś więcej? Opublikowany raport GUS o sytuacji opieki nad dziećmi do lat 3 pokazuje, że w Polsce na ponad 1 mln dzieci przypada 150 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. To są często dramaty tych rodzin. Proszę zatem o informację: Jakie programy dzisiaj są w przygotowaniu w celu (Dzwonek) zwiększenia liczby miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach publicznych? Co robi ministerstwo w tym zakresie?

Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Jana Szopińskiego, klub parlamentarny Lewica. Pani Minister! Wysoka Izbo!

Chciałbym się dowiedzieć, jakie środki z programu „Maluch+” wpłynęły do mojego województwa, kujawsko-pomorskiego, i ile w związku z tym nowych miejsc opieki, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, powstało w moim województwie i ile miejsc pracy powstało w ramach tych środków w gminach naszego województwa. Jak rząd ocenia współpracę z moim regionem w kwestii opieki nad dziećmi do lat 3? Czy są jakieś szczególne pozytywne przykłady tej współpracy? Czy rząd zamierza w przyszłości zwiększyć (Dzwonek) finansowanie programów opieki ze środków unijnych? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister!

Tym zasadniczym problemem będzie zorganizowanie opieki dla ich dziecka, ponieważ większość z nich będzie chciała wrócić do pracy. Otóż proponujecie im państwo albo pozostanie w domu i rezygnację z pracy, albo posłanie dziecka do żłobka prywatnego, w którym, jak to już było przed momentem mówione, opłata wynosi 1000 zł, 1200 zł, 1500 zł, 1700 zł albo więcej. Zdecydowanej większości polskich rodzin na takie opłaty nie stać. Faktycznie, liczba żłobków, liczba miejsc w polskich żłobkach wzrasta, ale są to miejsca w żłobkach niepublicznych, za które trzeba ponosić ogromne opłaty, chyba że dopłacają do tego samorządy. A więc znów mówimy o partycypowaniu samorządów w kosztach, które powinno (Dzwonek) ponosić państwo. W 70% gmin nie ma w ogóle żadnego żłobka. A więc proponuję i proszę bardzo o to, aby zwiększyć środki w programie „Maluch+” i zmienić sposób finansowania, bo części tych biedniejszych gmin nie stać na wkład własny. I jeszcze, panie marszałku, jeśli pan pozwoli, 2 sekundy na jedno pytanie. Kolejny raz jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, jak kilka tygodni temu, kiedy zajmowaliśmy się informacją rządu na temat sytuacji osób starszych, że zajmujemy się raportem, w którym są przeterminowane dane.

Przecież to jest kompletnie niepoważne. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Marta Wcisło, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.

Szanowni Państwo! Debatujemy, tak jak kolega powiedział, nad sprawozdaniem z 2018 r. Jest rok 2020, więc te dane, które podała pani minister, nie dość, że są nieaktualne, to jeszcze są nieprawdziwe. To jest po prostu nieprawda i oczekujemy od pani minister prawdziwych danych. Te prawdziwe dane podała chociażby pani koleżanka: średnio to jest 19%. Są to głównie duże miasta, dzięki nim te wskaźniki są przyzwoite, a w dużych miastach na szczęście nie rządzicie wy, tylko rządzą prawdziwi samorządowcy. Szanowni Państwo! To nieprawda również, że wzrosła liczba żłobków. Wzrosła liczba miejsc w żłobkach, ponieważ zmieniliście państwo parametry.

Chciałabym wiedzieć, jakie środki ministerstwo wydało na własne, że tak powiem, potrzeby finansowe przez te pół roku, kiedy to debatowaliście o wskaźnikach i parametrach, o czym pani minister mówiła. Dziękuję serdecznie. Z niecierpliwością będziemy czekali na odpowiedź pana ministra.

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Bardzo się cieszę, że pani minister powiedziała, iż preferowane są również inne formy opieki nad dziećmi do lat 3 niż opieka żłobkowa, że trwają prace nad zmianami w ustawie, dlatego że chciałabym się odnieść do zatrudnienia niani, która przysługuje rodzicom dopiero od 20. tygodnia życia dziecka. Państwo gwarantuje pomoc dla rodziców w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia, ale nie rozróżniacie państwo sytuacji rodzin wielodzietnych, kiedy rodzi się jednocześnie więcej niż jedno dziecko.

Miałam też taką sytuację. Spotkałam się z mamą trojaczków, wcześniaków, które urodziły się chore. Rodzice muszą wyjeżdżać do lekarza, muszą wyjeżdżać na rehabilitację. Jedno dziecko zostaje w domu, z dwójką muszą wyjechać. Nie mają opieki nad tymi dziećmi, ponieważ rodzina czy bliscy nie są w stanie tej opieki zabezpieczyć. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na pytanie, pani minister, czy może przygotowujecie państwo zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania, jeżeli chodzi o sytuację matek, które urodziły jednocześnie więcej niż jedno dziecko.

Dziękuję serdecznie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam taki apel w imieniu warszawianek i warszawiaków. Rozmawiamy o roku 2018, ale chciałbym przejść do roku 2019. Wysoka Izbo!

Jedna prośba jest taka, żeby dofinansowanie dla Warszawy do bezpłatnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 było co najmniej takie jak dofinansowanie w roku 2019 spółek powiązanych z panem ministrem Łukaszem Szumowskim. W roku 2019 to dofinansowanie spółek wyniosło ponad 22 mln zł.

Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Oczywiście problem opieki nad dzieckiem to jest problem nie tylko dużych miejscowości, ale także, powiedziałbym, Polski powiatowej, tych mniejszych miejscowości, gdzie bardzo często brakuje miejsc opieki, brakuje miejsc, gdzie rodzice mogą zostawić swoje pociechy. I pytanie do ministerstwa, do rządu, czy planowany jest w związku z tym program, który w szczególny sposób będzie traktował te małe społeczności lokalne w małych miejscowościach, ale nie tylko na ścianie wschodniej, bo rząd przyzwyczaił nas, że tam idą te fundusze, ale np. w takich województwach jak województwo śląskie, gdzie ta liczba miejsc na jedno dziecko należy do najniższych w kraju.

Ci rodzice zostali pozostawieni bez środków, bez możliwości opieki. Czy rząd przewiduje jakieś wsparcie finansowe właśnie dla tych pracujących zazwyczaj obojga rodziców? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Tomasz Olichwer, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ze sprawozdania Rady Ministrów dotyczącego opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynika, że w Polsce jest zdecydowanie za mało żłobków i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Jestem tym faktem bardzo zaniepokojony. W sprawozdaniach przekazywanych przez gminy oraz podmioty niepubliczne, tj. ok. 22% wszystkich gmin w Polsce, zadeklarowano potrzebę utworzenia nowych miejsc opieki, określając to na ok. 71 tys. miejsc. To są dane tylko z części Polski. Bardzo zmartwiło mnie również stwierdzenie w sprawozdaniu, że nie można wykluczyć tego, że dane są zaniżone ze względu na brak środków finansowych w gminach, np. na zakładanie żłobków. Smutna refleksja. Czy samorządy muszą uciekać się do ukrywania potrzeb mieszkańców, bo nie mogą liczyć na pomoc rządu? W związku z tym mam pytanie: Jakie działania zamierza podjąć rząd, żeby te gminy wróciły do warunków, na jakie zasługują wszyscy rodzice i dzieci? Oni też są Polakami. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Opieka nad dziećmi do lat 3 jest niezwykle istotna, ważna co najmniej z dwóch względów: po pierwsze, trzeba zapewnić dzieciom właściwą opiekę, merytoryczny nadzór, a z drugiej strony - umożliwić rodzicom podjęcie zatrudnienia. Bardzo się cieszę z tego, że zarówno nakłady na tę opiekę, jak i poziom użłobkowienia rosną, natomiast trzeba powiedzieć że jest to poziom absolutnie niewystarczający. Bardzo dużo mówiono tutaj o tym, że rodzice powinni mieć wybór. Oczywiście powinni mieć wybór, natomiast niestety go nie mają, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że nadal w ok. 70% gmin nie ma żadnego żłobka samorządowego, po drugie, nawet jeśli jest, to koszt, który ponoszą rodzice, jest kilkukrotnie wyższy niż koszt opieki przedszkolnej. Co należałoby zrobić? Nie wystarczy zbudować żłobek, trzeba zapewnić systematyczne wsparcie na wzór subwencji oświatowej. Dziękuję serdecznie.

Bardzo dziękuję, panie marszałku, szczególnie za ten spokój w prowadzeniu tak ważnej debaty. Po pierwsze, nie chce mi się ścigać z Prawem i Sprawiedliwością i mówić, kto ile dokonał.

To pokazuje, ile musimy wspólnie zrobić.

Chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy sytuację dramatyczną. Dramatyczną, dlatego że tysiące żłobków, pani minister, może nie przetrwać. Jedno zdanie, panie marszałku. 54% wszystkich żłobków to żłobki otworzone przez osoby fizyczne. Jeżeli dzisiaj kryteria COVID-owe pozwalają na przyjęcie tylko 50% dzieci, to większość tych żłobków może nie przetrwać następnych tygodni i miesięcy.

Nie odtworzymy tego, co zrobiły tysiące osób podejmujących na co dzień trud wychowania najmłodszych. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Adama Szłapkę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Pani Minister! Pani minister, to jest prehistoria, to jest czas, rzeczywistość Prawdziwa rzeczywistość jest tu i teraz. Chcę wykorzystać obecność pani minister, żeby zapytać o tę rzeczywistość tu i teraz, o to, co najbardziej martwi Polaków. Bardzo proste, konkretne pytanie. I pytanie: Jak zabezpieczyliście żłobki? Czy samorządy otrzymały wsparcie w wykonaniu testów dla personelu? Nie. Odpowiedź jest prosta: Nie zrobiliście tego. Zostawiliście samorządy, zostawiliście ten personel, zostawiliście rodziców. To jest odpowiedź, my znamy tę odpowiedź, ale żeby ta odpowiedź została dla potomnych, poproszę panią minister o przygotowanie odpowiedzi na to pytanie na piśmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią posłankę Katarzynę Kretkowską z klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo!

Żłobki funkcjonują głównie w dużych miastach, ale nawet w tych dużych miastach, takich np. jak Poznań, 2/3 żłobków to są żłobki niepubliczne, gdyż samorządów nie stać na zorganizowanie tylu miejsc w żłobkach, na ile jest zapotrzebowanie.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Te 2/3 żłobków nawet w tych dużych miastach, które (Dzwonek) zabezpieczyły organizacje pozarządowe, w tej chwili są zagrożone z uwagi na te obostrzenia i 2-miesięczny, 3-miesięczny przestój.

Jakie państwo przewidujecie nowe zabezpieczenia, żeby opieka żłobkowa prowadzona przez organizacje pozarządowe i przez samorządy w ogóle przetrwała? Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Grzegorza Brauna z koła Konfederacja. Wysoka Izbo! Kontynuuję wątek hipokryzji w postępowaniu władzy tak wykonawczej, jak i ustawodawczej. Skoro już powstaje raport na temat opieki, a zatem i bezpieczeństwa dzieci, skoro już uważacie za pożądane i słuszne ingerowanie państwa w tę sferę życia Polaków nieletnich, świeżo urodzonych, to czy nie czujecie państwo odpowiedzialności za bezpieczeństwo tychże najmłodszych w przestrzeni publicznej, która - jak sama nazwa wskazuje - będąc publiczną, podlega bezpośrednio jurysdykcji, a dziś jest pod coraz baczniejszym okiem władzy policyjnej administracji? Otóż w tej przestrzeni publicznej w ostatnich latach, właśnie już po tym czasie, którego dotyczy raport (Dzwonek), mamy do czynienia z radykalną, rewolucyjną inwazją w postaci manifestacji zboczeńców i promotorów zboczeń. W ubiegłym roku, którego ten raport już nie dotyczy, przez ulice większości dużych polskich miast przetoczyły się, przedefilowały parady dewiantów i promotorów dewiacji.

Proszę pana, zgłaszam się obrażony, oczywiście, w imieniu ludzi, których nie należy obrażać. Dziękuję panu serdecznie. Do widzenia panu. Jeszcze chciałem panu powiedzieć jedną rzecz: nie życzę sobie, żeby w polskim Sejmie obrażał pan ludzi. I bez względu na to, czy prowadzi te obrady pani marszałek Witek, czy ktokolwiek z marszałków, i bez względu na to, jakie ma poglądy, to nie dopuszczę do obrażania kogokolwiek w polskim Sejmie. Pani posłanko, proszę bardzo.

Może pan usiąść? Dyscyplina czasami pomaga w myśleniu. Wysoka Izbo! Panie Pośle Braun! Ale to jest czas na zadanie pytania. W odróżnieniu od pana posła Brauna ja to pytanie zadam. Statystyki można przedstawiać w różny sposób. Gdy mowa o raporcie, oczekujemy obiektywnych danych.

Wszyscy wiemy, że te koszty są znacznie wyższe.

I chciałam jeszcze zapytać o środki wydatkowane z programu „Maluch+”

Dziękuję bardzo. Zapraszam, pani poseł. Proszę bardzo, pani poseł. Pani Minister! Chciałam panią prosić o ewentualne potwierdzenie informacji, które zebrałam odnośnie do utworzenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w Warszawie.

Jeżeli mówimy o samorządach, o za małym zaangażowaniu w tworzenie miejsc opieki żłobkowej, to bardzo proszę nie mówić w ten sposób, że rząd nie daje i nie robi, ponieważ mamy wspólną pracę do wykonania (Dzwonek) To praca polegająca na tym, że posłowie w swoich samorządach lobbują na rzecz rodziny, rozmawiają z mieszkańcami i z samorządami, zachęcają, żeby może zrobić 1 km drogi mniej, a zaopiekować się rodziną. Chciała pani zadać sobie pytanie. Proszę bardzo. Wysoki Sejmie! Rzeczywiście nie zamierzałam tego pytania stawiać, ale zostałam do tego zainspirowana przez panią poseł z Platformy Obywatelskiej. Proszę pozwolić, że przytoczę kilka zdań: podejmowane do 2015 r. działania nie przełożyły się na rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Liczba żłobków i klubów dziecięcych pozostawała daleko niewystarczająca.

Sami państwo tak oceniliście siebie, a zatem pani teza, że nie wiadomo, jak było dobrze, jest nieuprawniona. Dla porównania: w 2017 r., jeśli chodzi o liczbę gmin, w których takie instytucje funkcjonowały, to 805, 32%, w 2018 r. - 930 gmin, 38%. Pani Minister! Moja uprzejma prośba, czy mogłaby pani wskazać progres, jaki dokonał się od 2015 r. w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 do roku bieżącego, żeby uzmysłowić posłom opozycji, jak wygląda sytuacja, jak wiele zostało zrobione. Ubolewam bardzo nad tym.

Różnica między Platformą Obywatelską a PiS-em jest taka, że my nigdy nie byliśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy.

Wysoki Sejmie! Chciałabym zaprotestować przeciwko słowom pana posła Brauna. Oczywiście zgadzam się z krytyką pana marszałka, że nie wolno w polskim Sejmie obrażać ludzi, ale chciałabym odnieść się jeszcze do wcześniejszych słów. Otóż pan poseł Braun z tej mównicy powiedział, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to organizacja przestępcza.

że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jest instytucja, która od 85 lat dba o to, żeby polscy seniorzy dostawali emeryturę. I na świecie nie ma innego (Dzwonek) powszechnego systemu emerytalnego niż taki, że młodzi pracujący płacą składkę, żeby starzy nie umierali z głodu. Rozumiem, że jak Konfederacja, nie daj Boże, kiedyś doszłaby do władzy, to do polskiego emeryta nie zapuka listonosz, nie przyniesie mu emerytury, bo organizacje przestępcze trzeba likwidować, to wie chyba każdy rząd.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Paszyk, klub parlamentarny PSL-Kukiz15. A, przepraszam serdecznie, przepraszam, pani poseł. Dziękuję, panie marszałku.

Powiedziałam już w trakcie swojego wystąpienia: państwo pozwolili na upychanie dzieci w mniejszej liczbie sal i są bardziej zapełnione placówki. To nie jest państwa dokonanie, to jest obniżenie standardów, to jest to, czego my w Warszawie nie chcemy i na to nie pozwalamy. A jak już życzy pani sobie, żeby uzupełnić dane dotyczące Warszawy, to pani powiem.

Państwo doskonale zdają sobie sprawę - panią minister chciałabym prosić, żeby pani odpowiedziała na to na piśmie - bo wynika to z danych samorządów, że dotacje rządowe pokrywają 10, maksymalnie 20% rzeczywistych kosztów budowy oraz utrzymania miejsc żłobkowych. Pozostałe koszty są na barkach samorządów, na barkach przedsiębiorców, a my uważamy, że to jest państwa zadanie. Nie wspieranie telewizji, nie wspieranie swoich, a opieka nad dziećmi. I nie nakładanie na samorządy nowych zadań, za którymi nie idą środki, bo te samorządy będą musiały teraz te żłobki.

Proszę bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Na wstępie bardzo mocno zaprotestuję przeciwko temu, żebyśmy tu w historycznych sporach, analizach się zakręcili. Dzisiaj, myślę, ważna jest refleksja na przyszłość, to co w opiece nad dziećmi do lat 3 państwo polskie może zrobić. Jest potrzebna błyskawiczna refleksja o działaniach do przodu, wyprzedzających tę sytuację. Bo czy w Poznaniu, w Warszawie czy w wielu innych mniejszych miejscowościach - problem jest ten sam, tzn. mamy zbyt mało miejsc. Nie dam się pani poseł wmanewrować w licytowanie, kto więcej, kto lepiej. Dzisiaj wszyscy powinniśmy, państwo jako ci, którzy sprawują władzę, postawić na dobre programy, które będą tę bazę żłobkową rozwijały. Pytanie na koniec. Pani minister, jakie resort (Dzwonek) planuje podjąć działania?

Dziękuję. Nie ma już żadnych osób zapisanych do zadania pytań, więc pan poseł Braun w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Oszczercza insynuacja padła z tej trybuny, pani poseł Leszczyna zasugerowała, niezgodnie z rzeczywistością, jakoby Konfederacja nie opowiadała się za wypełnianiem zawartych umów. Wręcz przeciwnie, Konfederacja bardzo skrupulatnie chciałaby wyegzekwować wywiązywanie się państwa, Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jej agendach, ze zobowiązań zaciągniętych wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Jednak to nie ma nic wspólnego z godziwością czy niegodziwością takiej instytucji, takiej piramidy finansowej, jaką jest bismarckowski z genezy ZUS.

A takie słowa, panie marszałku, jak zboczeńcy, sodomici, dewianci, to są słowa należące do słownika języka polskiego i nie sądzę, żeby były obraźliwe. Dziękuję serdecznie. Zapraszam podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej panią minister Barbarę Sochę.

Wysoka Izbo! Pierwsza uwaga, wstępna: z pewnym zdumieniem obserwuję, że duża część pytań dotyczy liczb i danych, które są zawarte w sprawozdaniu. A więc zachęcam państwa przede wszystkim do czytania. Oczywiście nie odniosę się teraz szczegółowo do każdego z tych pytań. Chętnie tej odpowiedzi udzielimy, częściowo też powtarzając informacje zawarte w sprawozdaniu. Natomiast do kilku stwierdzeń, które tu padły, chciałabym się odnieść. Po pierwsze, jeśli chodzi o liczbę żłobków, które powstały przez ostatnich 5 lat, to ja może odczytam dane: w 2015 r. było 2990 żłobków, w kolejnym roku - 3451, w kolejnym - 4271, w 2018 r. - 5080.

Rzeczywiście padły tu z mojej strony słowa, że użłobkowienie wynosi 24%. Te różnice są znaczące.

Jednocześnie zwracam uwagę, że to: za mało nie oznacza, że żłobki są jedyną formą opieki, i to nadal podtrzymuję. Opieka instytucjonalna nad dziećmi jest tylko czy aż jednym z elementów, jednym z ważniejszych, ale jednym z elementów szeroko rozumianej polityki rodzinnej. Ponieważ mamy przed sobą, na co bardzo liczę, merytoryczną, użyję jednak tego słowa, debatę nad strategią demograficzną, którą, mam nadzieję, niedługo będę miała możliwość zaprezentować, to myślę, że będzie też okazja porozmawiać o opiece nad dziećmi do lat 3 szerzej, nie tylko w rozumieniu dynamiki wzrostu liczb tych miejsc opieki, ale również w odniesieniu do różnych innych instrumentów, które tę opiekę mogą wspierać.

No ale niestety pomysły, które polegają na likwidacji, blokadach, rezygnacji.

Oczywiście nie są one dla nas zadowalające, dlatego tę politykę będziemy kontynuować, mam nadzieję, z dobrą współpracą przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, które też mają wielką rolę do odegrania. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Joannę Borowiak, sprawozdawcę komisji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Rozpatrujemy sprawozdanie Rady Ministrów o realizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 w 2018 r. Muszę powiedzieć, że z pewnym zdumieniem przyjęłam tak mocne upolitycznienie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Ministrów dotyczącym właśnie opieki nad dziećmi do lat 3. Nie spodziewałam się, że tego typu dyskusja będzie miała miejsce, dyskusja tak bardzo polityczna, w której padały tak dalece nieuprawnione tezy. Zdaje się, że sala plenarna Sejmu tak oddziałuje, wpływa na taki właśnie klimat dyskusji, ponieważ muszę powiedzieć, że na posiedzeniu komisji, mimo że dyskusja była bardzo ożywiona, dyskutowaliśmy dużo spokojniej i merytorycznie. Mam wrażenie, że niektórzy państwo posłowie z opozycji chcieli zabrać głos, ale na zupełnie inny temat. To niestety obniża rangę tej naszej dyskusji. Pojawiły się także pytania, na które odpowiedź państwo posłowie znajdą w dokumencie, nad którym teraz pracujemy. Tam państwo znajdą wszelkie informacje z podziałem na województwa, bo rozumiem, że każdego z nas interesuje, jak w naszym regionie ta opieka jest realizowana. Koniec 2018 r. - blisko 145 tys. miejsc opieki, o 70% więcej niż w 2015 r., kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejmował odpowiedzialność za Polskę. Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci do lat 3. na koniec 2018 r. wyniósł 19%. To o 60% więcej niż w 2015 r. Szczególnie cieszy wzrost liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w mniejszych gminach, w gminach wiejskich chociażby. Te dane dowodzą, że rozwój instytucji opieki nad tymi najmłodszymi dziećmi jest priorytetem polityki rodzinnej rządu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, by powstawały i działały bezpieczne miejsca opieki dla dzieci najmłodszych. Celem jest to, by do 2030 r. wskaźnik objęcia opieką instytucjonalną dzieci w wieku do lat 3 wyniósł 33%. Aby to osiągnąć, likwidowane są bariery niewystarczającej liczby miejsc opieki, powstają nowe miejsca opieki, prowadzone są również działania, by obniżyć koszty, o których mówili też państwo posłowie, prowadzenia i tworzenia miejsc opieki przy zachowaniu jakości usług i bezpieczeństwa dzieci. Szanujemy autonomię rodziny, chcemy, żeby rodzice mogli decydować, dokonywać wyboru między opieką domową a opieką instytucjonalną, także pomiędzy jej formami.

Otóż tak, są potrzebne najwyższe kwalifikacje, ponieważ dzieci są naszym skarbem i od najwcześniejszych miesięcy życia musimy się o nie jak najlepiej troszczyć, a zatem te kwalifikacje są konieczne. Jeszcze jedno. Padło tutaj takie twierdzenie, że powinniśmy dawać wędkę, a nie rybę. Nie, bo to tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć rodzicom: albo macie państwo miejsce dla swojego dziecka w żłobku czy klubiku, albo musicie je sobie stworzyć sami. Nie mylmy pojęć, szanowni państwo posłowie. Jeszcze raz dziękuję za tę dyskusję. Ona na pewno była twórcza, mówię o głosach merytorycznych, wyłącznie o tych, które się odnoszą do dzisiejszego dokumentu, nad którym pracujemy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, zamykam dyskusję. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny proponuje, aby Sejm przyjął sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r., zawarte w druku nr 83. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Dziękuję serdecznie. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, druk nr 392.

Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 383 i 392) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Nie wiem, czy mówiłem tak szybko jak pani marszałek Witek, ale strasznie się starałem. Jak pan to ocenia, panie pośle? Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z pracy Komisji Finansów Publicznych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, zawartym w druku nr 383, sprawozdanie komisji to druk nr 392. Pani marszałek Sejmu skierowała rządowy projekt ustawy do pracy w Komisji Finansów Publicznych w celu odbycia pierwszego czytania, jak również rozpatrzenia tego projektu. Projekt dotyka finansów publicznych, a właściwie dotyka reguły stabilizacyjnej, reguły wydatkowej, która jest zawarta w ustawie o finansach publicznych, a która zabezpiecza finanse publiczne państwa polskiego przed nadmiernym zadłużaniem się, przed nadmiernym wydatkowaniem. Można by powiedzieć, że ta reguła wydatkowa w sposób stabilny rozkłada równomiernie na wszystkie lata wydatki, czyli przy dobrej koniunkturze te wydatki poniekąd hamuje, przy gorszej pozwala jednak na dokonywanie tych wydatków, bo odnosi się do lat wstecz, do wydatków z lat poprzednich.

Widać bardzo wyraźnie, że zarówno reguła wydatkowa, polityka fiskalna, jak i polityka wydatkowa rządu są tutaj bardzo skuteczne.

Z drugiej strony oczywiście są ulgi w ZUS-ie, umorzenia tego typu. Chodzi także o konieczność zamrożenia gospodarki, szczególnie w dziedzinach turystyki, transportu publicznego czy usług. Faktem jest, że przychody budżetowe na pewno będą w tej dziedzinie mniejsze. Stąd widać bardzo wyraźnie, że bez zamrożenia czy zawieszenia reguły wydatkowej bardzo trudno byłoby zrealizować w roku 2020 wydatki budżetowe i zrealizować ambitny, zrównoważony budżet. To jest problem, który jest powszechny w całej Europie. Na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej wszystkie kraje mogą te wydatki poluzować.

Wręcz pokazuje się ścieżkę powrotu do reguły wydatkowej. To jest niezwykle cenne. Komisja finansów rozpatrzyła ten projekt ustawy. Dyskusja była bardzo długa, merytoryczna. Często schodziło na dyskusję o poziomie długu publicznego.

W imieniu Komisji Finansów Publicznych wnioskuję, aby Wysoka Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych w przedłożonym zakresie, druk nr 392. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dowiemy się, co ma w tej sprawie do powiedzenia Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, bo poprosimy pana Zdzisława Sipierę. Zapraszamy, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Natomiast chodzi o skalę tego problemu. I ta reguła, poluzowanie tej reguły, dopisanie w ustawie tego elementu, który do tej pory nie był przewidywany, czyli epidemii, jest tym właśnie zamysłem ustawowym wprowadzającym możliwość czasowego poluzowania tych wydatków. Proszę państwa, głównym zadaniem, tym, czym się będziemy zajmowali, jest cały czas ochrona rynku pracy, miejsc pracy oraz miejsc, gdzie ta praca jest podawana, gdzie są przedsiębiorstwa.

Minister finansów o tym mówił.

To jest czas na decyzje. To nie jest czas na debaty. Często spotykamy się z takim zastrzeżeniem, że klub Prawa i Sprawiedliwości niektóre ustawy przeprowadza sprawnie i szybko. Pozwolą państwo, bo jest okazja, żeby o tym powiedzieć. To nie są małe pieniądze, przyznacie państwo. Tarcza antykryzysowa.

To są konkrety. Dobre zarządzanie polega na tym, żeby przewidzieć i wcześnie reagować, a nie czekać na efekty. Tak to traktujemy i uważamy, że to idzie w tym kierunku. Dlatego też klub Prawa i Sprawiedliwości w całej rozciągłości będzie popierał tę ustawę. Mamy nadzieję, że również opozycja się przychyli - przynajmniej takie głosy słyszeliśmy w komisji, zobaczymy, jak to będzie podczas głosowania - bo to, proszę państwa, jest wymiar odpowiedzialności za polskie państwo, odpowiedzialności za to, co będzie nas czekało w najbliższych miesiącach i latach. Ustawa jest określona. Żadne bezpieczniki konstytucyjne nie są naruszone. 3% i 55% są nienaruszalne. To jest gwarancja, że nie będzie żadnych problemów z przekroczeniem tych elementów, które są zapisane w prawie, i bezpiecznikiem finansów publicznych. Uważamy, że to, co będzie w najbliższym czasie możliwe do zrealizowania poprzez działania rządu, będzie stabilizowało sytuację w Polsce. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam serdecznie pana posła Janusza Cichonia z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Omawiamy zmianę ustawy o finansach publicznych, której kluczowym elementem jest od 2013 r. stabilizująca reguła wydatkowa. To reguła antycykliczna, której istota sprowadza się do tego, że w latach chudych, czyli w latach spadku tempa wzrostu gospodarczego, możemy wydawać nieco więcej, natomiast w latach tłustych, kiedy to tempo wzrostu gospodarczego jest odpowiednio wysokie, budujemy poduszkę i wydajemy. W nieco mniejszym tempie wzrosną wydatki, niż wynikałoby to z tego wzrostu gospodarczego.

W tle była też zmiana dotycząca sposobu kalkulowania działań dyskrecjonalnych. Uwierała was bardzo, obchodziliście ją, przypisywaliście tym działaniom dyskrecjonalnym np. wzrost dochodów podatkowych, mimo że zdawaliście sobie sprawę z tego, że ten wzrost w dużej mierze wynika z tego, że rośnie gospodarka i że te dochody mają procykliczny charakter. To wam w dalszym ciągu nie wystarczało. Wobec tego zaczęliście wyprowadzać wydatki poza budżet. Przykład Funduszu Solidarnościowego - wypłata trzynastek to jest klasyk, jeśli chodzi o tego typu działania, nie pierwszy i nie jedyny. O tyle byłaby dzisiaj lepsza sytuacja polskich finansów publicznych i większa swoboda reakcji, niż mamy dzisiaj, w tych naprawdę bardzo trudnych czasach. Przy czym my rozumiemy, że sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna. Mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym, stanem klęski żywiołowej, i to z pewnością uzasadnia klauzulę wyjścia, która w tej ustawie, nawiasem mówiąc, jest zapisana. Ale wy kluczycie. Proponujecie rozszerzenie warunków wykorzystania klauzuli wyjścia o stan epidemii i w ten sposób próbujecie tę regułę zawiesić. To naprawdę jest dziwne rozwiązanie, żeby o klauzuli wyjścia, zawieszeniu reguły decydował minister zdrowia. Na szczęście wpisaliście w ten projekt spadek tempa wzrostu gospodarczego jako dodatkowy warunek. 2 punkty procentowe to nie jest za wiele. Wiemy, że ta elastyczność dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki, jest nam bardzo potrzebna. W obliczu recesji niezbędne jest wsparcie systemu ochrony zdrowia, ochrony ludności, także ochrony gospodarki. Pozwala na to także Unia Europejska.

Chcemy też mieć pewne miejsce dla impulsu fiskalnego w kolejnych latach. Ta nadmierna swoboda może w tym niestety przeszkadzać. Inna kwestia, czy to będą inwestycje publiczne, jak wam się wydaje (Dzwonek), czy np. nie lepiej byłoby przejściowo obniżyć podatki. No zobaczymy.

To jest ograniczenie pokusy obchodzenia reguły wydatkowej w przyszłości, po powrocie tak naprawdę do niej, a jednocześnie kontrola parlamentu, kontrola w demokratycznym procesie tego, jak wykorzystujecie to narzędzie i zawieszenie tej reguły. Żeby wyeliminować te mankamenty, składamy poprawki. A pan marszałek z przyjemnością je przyjmie. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam panią posłankę Hannę Gill-Piątek, klub parlamentarny Lewicy. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś zdejmujemy zabezpieczenia z wydatków państwa, bo trzeba sfinansować walkę z kryzysem. Gdybyście posłuchali państwo Lewicy i wprowadzili stan klęski żywiołowej wtedy, kiedy o tym mówiliśmy, moglibyśmy w sposób adekwatny zareagować, bez tej dyskusji, którą toczyliśmy dzisiaj, bo ta ustawa przewiduje takie postępowanie w stanach nadzwyczajnych. Teraz trzeba dodawać stan epidemii jako powód luzowania reguły wydatkowej. Czy może być lepszy dowód na to, że faktycznie mamy do czynienia w Polsce ze stanem nadzwyczajnym? Pojawia się kilka ważnych pytań. Jaką mamy gwarancję, że nie zostaną złamane progi ostrożnościowe? Po tej dyskusji nie jestem do tego przekonana. Nie jesteśmy do tego przekonani jako Lewica, ponieważ relacja długu do PKB, wiadomo, nie powinna przekroczyć 55% zgodnie z ustawą, a 60% - zgodnie z konstytucją. Obecnie do tego ostatniego brakuje nam zaledwie 12 punktów procentowych. Wobec spadku PKB o 4,3%, jak szacuje Komisja Europejska, przekroczenie tych progów jest bardzo realne. Jak rząd zagwarantuje, że realizacja tej ustawy nie sprawi, że za kilka miesięcy nie będziemy zbierać się tu, by zmieniać konstytucję, bo za dużo wydacie? A ile już w tej chwili państwo wydaliście? Do kogo tak naprawdę trafiły te pieniądze? Gdybyście dbali o ludzi tak samo jak o banki, kryzys byłby mniej dotkliwy. Zagwarantujcie, że pieniądze z poluzowania reguły wydatkowej trafią tam, gdzie powinny. Zamiast hojnie rozdawać nasze fundusze na Kościół, media publiczne, podratowanie budżetów rodzin ministrów, premie w spółkach, zrealizujcie po prostu postulaty Lewicy służące zwykłym ludziom. Przypomnę tutaj trzy z nich: świadczenie kryzysowe - 1800 zł dla wszystkich, którzy stracili źródło utrzymania w kryzysie, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zagrożonych firm - 3/4 wynagrodzeń finansowane przez państwo, koszty stałe przedsiębiorców - połowa kosztów najmu, opłat za prąd dla małych przedsiębiorstw w kryzysie. To są proste postulaty, które mogłyby być tutaj sfinansowane. Lewica będzie za tym projektem, ale chcemy mieć pewność, że te pieniądze trafią tam, gdzie trzeba, że realnie pomogą.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Mianowicie mimo że mamy do czynienia z projektem rządowym, znowu uniknięto nawet najbardziej podstawowych konsultacji. Gdyby te konsultacje się odbyły, to na pewno w ich ramach uwzględniono by stanowisko Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a w tym stanowisku bardzo ciekawie zostały wyłuszczone istotne problemy, które, jak myślę, byłyby bardzo ważne. Ano na to, że co najmniej od 4 lat mamy problem, jeśli chodzi o przejrzystość finansów publicznych w Polsce.

To jest pierwsza sprawa. Panie ministrze, nie da się debaty nad tym projektem oddzielić do tego, co obserwowaliśmy w ostatnim czasie.

A to, jeśli chodzi o finanse samorządów gminnych związane z reformą oświaty.

Tylko, panie pośle, proszę nie prezentować tych danych tak, jakby to były pana pieniądze czy pana środowiska politycznego. To są pieniądze przedsiębiorców, to są pieniądze Polaków, które tworzą budżet państwa, tworzą finanse publiczne. To jest też refleksja, która się w toku tej debaty sama nasunęła. Zdaniem Koalicji Polskiej, którą mam przyjemność reprezentować, oczywiście ten szczególny czas wymaga rozwiązań nadzwyczajnych i takowe w tej ustawie są zawarte, ale też wymusza, i na to chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę, porządki w finansach publicznych i dopracowanie pewnej przejrzystości, która niestety w ostatnim czasie gdzieś tam się rozjeżdża.

Ale nie możemy tego rozdzielić z ogólną sytuacją finansów publicznych i działaniami, które w ostatnich latach wokół finansów publicznych dokonywał rząd. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Jakuba Kuleszę z koła Konfederacji. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Żaden rok rządów Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji dobrej światowej koniunktury nie skończył się nadwyżką budżetową. Żaden. Wszystkie kraje naokoło, Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Dania, miały nadwyżki budżetowe, tylko nie Polska. Przez 5 ostatnich lat Polki i Polacy byli przez rząd Prawa i Sprawiedliwości opodatkowywani i, co gorsze, zadłużani. Przyszedł kryzys, choć, jak powiedział Stefan Kisielewski, to nie kryzys, to rezultat, rezultat państwa fatalnych, szkodliwych decyzji. W związku z tym kryzysem czeka nas z jednej strony eksplozja długu publicznego, a z drugiej strony spadek albo przynajmniej stagnacja PKB. Oczywiście możecie majstrować przy stosowaniu stabilizacyjnej reguły wydatkowej, ale co zrobicie, jak dług osiągnie konstytucyjny limit 60% PKB? Powiedzcie szczerze: Co zrobicie? Zmienicie konstytucję? Zmienicie definicję zadłużenia? Może zmienicie definicję PKB? Czy widzicie twarz ministra Rostowskiego, twarz tej właśnie kreatywnej księgowości rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zmiany definicji po to, żeby nie przekraczać tego konstytucyjnego progu? Żeby nie było, że tylko państwa krytykuję, powiem państwu, co należy zrobić. Muszą państwo zacisnąć pasa. Nie chodzi mi o pas obywatela, chodzi mi o państwa pas. Odpowiedzialny gospodarz przez 7 tłustych lat oszczędza na lata chude, a nawet jak nie oszczędzi, to w czasie kryzysu w pierwszej kolejności szuka oszczędności, a nie leci z językiem na wierzchu po chwilówkę, po siano do Bociana. Zapytacie, jak macie zacisnąć ten swój pas. Po pierwsze, głęboka deregulacja, czyli likwidacja tysięcy zbędnych, szkodliwych, kosztownych przepisów. Po drugie, debiurokratyzacja, likwidacja setek zbędnych, szkodliwych i kosztownych urzędów i instytucji. Jeśli natomiast chcecie stymulować gospodarkę, to w żadnym razie nie za pomocą nieefektywnej urzędniczej redystrybucji pieniędzy zagrabionych przyszłym obywatelom. To nie zadziała. Proponuję obniżkę opodatkowania pracy albo najlepiej likwidację opodatkowania pracy. To zatrzyma nadciągającą falę bezrobocia, to wyciągnie ludzi z szarej strefy, to sprawi, że obywatelowi wreszcie zacznie się opłacać zatrudnienie, pracowanie, a przedsiębiorcom zacznie się opłacać większe zatrudnienie. I te obietnice kandydatów, dyletantów ekonomicznych, prezydenta Dudy czy prezentera Hołowni, o tym, by zwiększyć zasiłek dla bezrobotnych powyżej płacy minimalnej, włóżcie między bajki, najlepiej pomiędzy „Kapitał” Marksa a „Ogólną teorię zatrudnienia, procentu i pieniądza” Keynesa. Bardzo się cieszę, że pana widzę. Apeluję do pana: proszę nie iść drogą ministra rządu PO-PSL, ministra Rostowskiego, drogą kreatywnej księgowości. Wiem, że często jest pan do tego ministra porównywany. Proszę nie słuchać też tych socjalistów z ław poselskich, i tych pobożnych z prawej strony, i tych bezbożnych z lewej strony.

Gdy uzasadniałem poprawkę Krzysztofa Bosaka wprowadzającą do artykułu o zawieszeniu kredytów automatyzm, czyli żeby nie było tych wniosków, bez zbędnej biurokracji, szybko i sprawnie, to przedstawiciel rządu bez słowa uzasadnienia powiedział: przeciw. No i słusznie oburzona posłanka Lewicy zapytała: Dlaczego? Na to wchodzi on, cały na biało, prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, wyjaśniając: bo skorzystają z tego bogaci. Na co posłanka Lewicy: no to przeciw. I tak właśnie wyglądają wspólne rządy socjalistów, i tych pobożnych, i tych bezbożnych. Niestety te rządy, ta pogarda wobec bogatych, wobec dobrobytu skończy się katastrofą biedy. Jak dobrze wiemy, socjalizm wszystkim równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze. Dziękuję serdecznie. I ci pobożni, i ci bezbożni dali to, panie pośle, że może pan w demokratycznym kraju wygłaszać swoje poglądy, za które serdecznie dziękuję. Proszę państwa, otwieram zadawanie pytań. Minuta na pytanie. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska, klub parlamentarny PSL - Kukiz15. Panie Ministrze! I pański zespół, który jest dzisiaj obecny! To jest pewna wyjątkowa okazja, ale ustawa o finansach publicznych sprawia, że to dobrze, że tak jest.

W uzasadnieniu państwo napisaliście, że dotyczy to 90% sektora finansów publicznych, zarówno jednostek państwowych, jak i samorządowych. Chciałbym w związku z tym zapytać, jaką projekcję państwo przewidują jako resort finansów, jeżeli chodzi o te problemy samorządowe, które samorząd aktualnie przeżywa? Czy to mieści się, że tak powiem, w rozumieniu tej nowej regulacji, którą w dniu dzisiejszym omawiamy i która za chwilę ma być uchwalona (Dzwonek), z tej racji, że wpływy podatkowe spadły od 30 do 40% w zależności od rodzaju podatku w jednym miesiącu? Niektóre samorządy sygnalizują, że rosnące koszty i spadek wpływów mogą sprawić, że będą miały kłopoty z realizacją budżetu już w listopadzie obecnego roku, przy utrwalającej się dynamice. Mówił pan tak fantastycznie, że byśmy słuchali i słuchali. Pan poseł Robert Obaz z klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo!

Jak państwo zagwarantują tymi wszystkimi rzeczami, o których tu mówił poseł przede mną, że te samorządy przetrwają i na koniec roku będą mogły utrzymywać szkoły, żłobki, przedszkola oraz zapłacić pensje swoim urzędnikom, których chcecie zwolnić? Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Krutul, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jeszcze parę miesięcy temu, kiedy rząd pracował nad budżetem, ogłaszał, że to najlepszy budżet od 30 lat, budżet, który miał być zrównoważony i bezpieczny. Prezes NBP mówił, że dysponujemy nieprzebranymi ilościami gotówki. W marcu wasi urzędnicy byli już ostrożniejsi. Twierdzili, że gotówki jest wystarczająca ilość, a PKB będzie na poziomie 2%. Recesja. Co się stało, panie premierze? Czy państwo polskie, podobnie jak Agencja Rezerw Materiałowych, było przygotowane na każdą ewentualność, z wyjątkiem pandemii? Dzisiaj mówicie, że chcecie pomóc m.in. służbie zdrowia.

Zamiast pomagać Polkom i Polakom, zaczęliście finansować interesy swoich ministrów. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiemy, że koalicja rządowa uwielbia komplikować i gmatwać. Gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej, nie musielibyśmy toczyć dzisiaj tej dyskusji i się przekonywać. PiS uwielbi wszystko ukrywać i działać pod osłoną nocy. Lewica będzie nieustannie nawoływać i domagać się, aby wydatki państwa były jawne i przejrzyste. Chcemy wiedzieć, komu i ile dajecie. Dlatego pytam, gdzie my, obywatele i obywatelki, gdzie my, parlamentarzyści, znajdziemy szczegółowe sprawozdania z wydatków budżetowych mających wyciągnąć z kryzysu nasze państwo, mających pomóc naszemu krajowi w zwalczaniu skutków pandemii. Komu i ile? Proszę o odpowiedź na piśmie.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Izabela Leszczyna, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! 4 lata rekordowych dochodów podatkowych, świetnej koniunktury gospodarczej, 4 lata uszczelniania systemu podatkowego. Wystarczyły niespełna 3 miesiące epidemii, z którą rząd PiS, jak twierdzi, poradził sobie najlepiej na świecie, żeby okazało się, że jesteśmy bankrutem. Mamy katastrofę finansów państwa. Chciałabym, żeby pan minister z mównicy, przed Wysoką Izbą, potwierdził, że szacowany deficyt sektora finansów publicznych w tym roku ma wynieść 13% PKB, 200 mld zł. To znaczy, że zostawiliście Polaków na tę ostrą zimę na bosaka, w dodatku, jak się przeziębią i będą chorzy, to nie będzie nawet na system ochrony zdrowia, żeby ich leczyć. To zrobiliście każdej Polce i każdemu Polakowi, bo przez 4 lata przehulaliście [[Dzwonek]] ich pieniądze. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Dariusza Rosatiego, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. A jeżeli go nie ma, a nie ma, to zapraszam panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W czasach, gdy powinniśmy szczególnie oszczędzać, w czasach, gdy powinniśmy każdą złotówkę oglądać dwa razy, żeby wydać ją jak najbardziej efektywnie, wy po prostu wzięliście 70 mln zł i wyrzuciliście je w błoto, drukując ulotki wyborcze, bo pakietami wyborczymi tego nie nazwałabym. Dziś chcecie, by z powodu epidemii zamrozić regułę wydatkową, ale reguła nie jest żadną regułą, jeśli się z nią postępuje, jak wy postępujecie z nią od paru lat. Najpierw ją zmienialiście, potem ją obchodziliście.

Panie ministrze, pan dobrze zdaje sobie z tego sprawę (Dzwonek), że to nie jest koszt naszej epidemii i lockdownu, i zamrożenia gospodarki, bo gros z tych pieniędzy było już w deficycie, który był przez was założony przez obchodzenie reguły finansowej i wydawanie pieniędzy na lewo i prawo w czasie dobrej koniunktury. Czy pozwolicie uszczelnić regułę finansową, regułę stabilizującą? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, bijący sobie brawo na wejście. Wspaniale podsumowała te absolutnie nieodpowiedzialne niemalże 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo wszyscy wiemy, że pomimo dobrej koniunktury, pomimo tego, że firmy pracowały, pracownicy pracowali, rząd hulał, rozdawał, prowadził absolutnie nieodpowiedzialną politykę finansową. Okazuje się, że pomimo tylu lat dobrej koniunktury, pomimo tego, że mogło być dzisiaj tak, że zaoszczędzone wtedy pieniądze mogłyby służyć rozruszaniu gospodarki, budowaniu różnych impulsów i stawianiu polskich firm na nogi, dzisiaj tych środków nie ma. Dzięki Unii Europejskiej, znowu dzięki Unii Europejskiej, dzięki przepisom europejskim, przychodzicie dzisiaj do Sejmu z pomysłem na kolejne środki, które będziecie pożyczać. Dzwonek Panie ministrze, jeżeli mamy pracować tutaj, współpracować, przyjąć tę ustawę, to proszę stanąć w prawdzie i powiedzieć, jaki jest deficyt, rzeczywisty deficyt budżetu państwa, który niedawno Sejm przyjął, bo to, że ten deficyt poukrywaliście w różnego rodzaju funduszach, jest faktem. Proszę mieć cywilną odwagę, stanąć tutaj przed Wysoką Izbą i powiedzieć, jaki jest rzeczywisty deficyt w budżecie państwa, poukrywany w różnego rodzaju funduszach. Pani poseł Zofia Czernow, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałabym w pytaniu kontynuować to, co rozpoczęli posłowie wypowiadający się przede mną, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w okresie prosperity i ile zaoszczędzono na okres dekoniunktury, ale z nieco innego punktu widzenia, bowiem chciałabym dojść do tego, dlaczego tak się stało. Z jednej strony niewątpliwie przyczyną było to, że rząd nie szanował tej reguły, obchodził ją, wyprowadzał pieniądze poza budżet i rozdawał więcej, niż powinien. Myślę, że trzeba zapytać o rolę ministra finansów. Przecież minister finansów powinien stać na straży finansów publicznych. I proszę mi powiedzieć, panie ministrze, czy nie sądzi pan, że jedną z przyczyn jest to, że obecnie, tak jak nigdy dotąd nie było, minister finansów znajduje się na bardzo niskim szczeblu hierarchii w rządzie. Wszyscy inni się wtrącają, pan minister o niczym nie decyduje. I po drugie, panie ministrze, czy pan będzie miał na tyle cywilnej odwagi, żeby pilnować finansów publicznych?

Jeszcze pana nieraz do ściany przykują. Pan Krzysztof Piątkowski, pan poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Luzujecie stabilizacyjną regułę finansową, i słusznie, należy tak postępować w czasie kryzysu gospodarczego, należy tak robić, ale warto przypomnieć przy tej okazji, że ten kryzys zaczął się znacznie wcześniej niż epidemia COVID-19, jeszcze przed waszym pseudozrównoważonym budżetem. Należy jasno powiedzieć, że niestety wprowadzacie te ograniczenia w oparciu o niezgodną z konstytucją ustawę. Jednocześnie, i to muszę powiedzieć jako były samorządowiec, zaciskacie pętlę na szyi samorządów, które mają coraz mniejsze dochody z powodu epidemii, a jednocześnie - coraz większe koszty z powodu waszych decyzji. Dlatego pytam: Kiedy wreszcie zabierzecie się państwo za tarczę dla samorządów? Pan Piotr Borys, poseł Koalicji Obywatelskiej i mój dobry kolega.

Jest pan obecny na posiedzeniu Sejmu bodajże drugi raz, po raz pierwszy ze swoim zastępcą. Chciałbym, żeby pan odpowiedzialnie, pod rygorem powiedzenia prawdy powiedział, jaki dzisiaj mamy deficyt w finansach publicznych. Istnieją oczywiście przesłanki, o czym mówi Unia Europejska, dotyczące klauzuli wyjścia, ale nie mogą one być stosowane pod rygorem zagrożenia średniookresowego rozwoju, średniookresowej stabilizacji. Tymczasem w czasach naprawdę największej prosperity nie przygotowaliście Polski na czas trudny, wydawaliście po prostu za dużo. Pan doskonale o tym wie. Dzisiaj większość pomocy dla przedsiębiorców zlokalizowana jest w dwóch funduszach, które nie obciążają deficytu państwa. To jest blisko 200 mld zł. Żądam informacji, jaki jest dzisiaj prawdziwy deficyt w finansach publicznych. I chcę powiedzieć, że musi pan za chwilę przystąpić do nowelizacji budżetu, bo w obecnie funkcjonującym budżecie mamy wzrost gospodarczy i zerowy deficyt. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Łącki, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oj, przepraszam. Tak pokrótce można streścić rządy PiS-u w Polsce. Chaos społeczny, chaos polityczny, chaos gospodarczy. A po dzisiejszych obradach jeszcze do tego można dołożyć chaos prawny, bo te ustawy, które się teraz robi, robi się na kolanie po to, żeby tuszować wszystko to, co się zrobiło przez ostatnie 4 lata. Dlaczego się dopisuje stan epidemii? Ano dlatego, że się nie ogłosiło stanu klęski żywiołowej, który już w tej ustawie jest. Bo gdyby się ogłosiło stan klęski żywiołowej, to trzeba byłoby wypłacić przedsiębiorcom i tym, którzy stracili pracę i swoje miejsca pracy, i tym, którzy stracili firmy, odszkodowania, które by im się należały. A tak nie trzeba tego robić. Daje im się jałmużnę, a przez jałmużnę tworzy się społeczeństwo klientowskie, klientów, a nie społeczeństwo obywatelskie. I wy, proszę państwa, panowie z PiS-u i panie z PiS-u, i wy, [[Dzwonek]] panowie ministrowie z PiS-u [[Oklaski]] tworzycie państwo klientów. Mam do was jedno pytanie, fundamentalne: Kiedy przestaniecie psuć moją ojczyznę? Czy pan poseł Michał Szczerba jest na sali? Jeżeli nie ma, to poprosimy pana posła Dobromira Sośnierza z koła Konfederacja. Zabiegacie państwo o wyrwanie bezpieczników z systemu finansowego, żeby móc się dalej zadłużać, tylko że tutaj powstaje problem, kredyt nie jest narzędziem bogacenia się sam w sobie, kredyt może być dobry, kiedy ktoś ma pomysł na inwestycje, kiedy wie, w co zainwestować i jak, żeby się to potem zwróciło, natomiast kredyt konsumpcyjny jest narzędziem ubożenia tylko, bo to się przeje, przepije, a oddać trzeba z odsetkami. Dlatego jeśli ktoś przychodzi po kredyt, to trzeba sobie zadać dwa piekielnie ważne pytania, i liczę, że uzyskamy na nie odpowiedź: W co chcecie zainwestować te pieniądze, żeby to się zwróciło, i co już zrobiliście, żeby zaoszczędzić pieniądze, żeby sprawdzić, czy aby na pewno potrzebujecie tego kredytu? Ilu już zwolniliście niepotrzebnych urzędników? Ile już zbędnych programów rozrzutnego rozdawnictwa zlikwidowaliście? Czy już pożegnaliśmy się z planem budowy bezsensownego lotniska pośrodku niczego? Czy nie jest czasem tak, że właśnie chcecie zachować swój rozrzutny tryb życia i dlatego się zapożyczacie, żeby rozrzucać pieniądze z helikoptera i mówić, i wywiązać się z obietnic (Dzwonek), które teraz nieodpowiedzialnie składacie, że wszystkim na wszystko dacie? Dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Katarzyna Ueberhan, klub parlamentarny Lewica.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy tutaj do czynienia z luzowaniem stabilizującej reguły wydatkowej. Jest to w normalnych warunkach sytuacja niebezpieczna. W obowiązującej ustawie o finansach publicznych nie określono sposobu powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej. Przedłożony projekt zawiera takie warunki, które mają określić właśnie długość ścieżki powrotu, która jest określona na podstawie skali, charakteru kryzysu. W uzasadnieniu można znaleźć kolorowy graf, można znaleźć ładnie wyglądające, fachowo na papierze wyglądający wzór formuły na klauzulę wyjścia. Jednak w żaden sposób nie zwiększa to przejrzystości finansów publicznych, które w naszym kraju są niestety przykładem kreatywnej księgowości. W uzasadnieniu wskazali też państwo na granice czasowe: 2, 3 lub 4 lata, w zależności od skali załamania gospodarki. Ale co to tak praktycznie oznacza: mniejsza lub większa skala załamania gospodarki (Dzwonek) czy zła sytuacja makroekonomiczna? Takie określenia jak: większy, mniejszy, zły nie są to wskaźniki ekonomiczne, więc pytam: Jak dokładnie będą to państwo określać i uzależniać czas powrotu do wyjścia z tej klauzuli? Pani posłanka Katarzyna Kretkowska, klub parlamentarny Lewica. Zapytam się, bo był wykreślony pan poseł Jan Szopiński, a widzę pana posła: Będzie pan się zgłaszał do głosu, tak? Dziękuję. Wysoka Izbo! Jaki jest faktyczny stan budżetu państwa? Jaki jest faktyczny stan deficytu budżetowego? Ile faktycznie dotąd wydano na działania związane z ratowaniem gospodarki, z ratowaniem przedsiębiorców, z ratowaniem Polaków, Polek, pracowników, pracowniczek po nastaniu pandemii? To są podstawowe pytania, na które powinniśmy dostać wyliczenia co do drugiej pozycji po przecinku lub dalej, zanim przystąpimy do tego typu projektu, jak dzisiejszy, [[Oklaski]] czyli odstąpienie, poluzowanie stabilizującej reguły wydatkowej. Komisja Europejska w marcu tego roku dopuściła takie poluzowanie, ale po to, żeby państwa podjęły działanie na rzecz zwiększania możliwości służby zdrowia, ochrony ludności i ochrony gospodarki. Ile dotąd na to wydano i ile państwo zamierzacie wydać konkretnie na ochronę ludności? Czy zamierzacie państwo wprowadzić świadczenie kryzysowe, chociażby to, które proponuje Lewica? Czy zamierzacie państwo pokrywać koszty stałe przedsiębiorstw dotkniętych lockdownem, jak proponuje Lewica? Czy zamierzacie państwo zwiększyć wydatki na służbę zdrowia do 7,2%, jak proponuje Lewica?

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.

Szanowny Panie Marszałku! Będę miała do państwa pytania. Ale chciałabym powiedzieć, że przez ostatnią kadencję opróżniliście państwo wszystkie kieszenie, opróżniliście państwo, pieniądze wzięliście z konta Funduszu Pracy. Przecież to były pieniądze przedsiębiorców.

Dzisiaj nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia. Państwo wprowadziliście 35 podatków i danin. I dzisiaj państwo przychodzicie i mówicie, że dajecie przedsiębiorcom. I teraz pytanie, panie marszałku: Czy leci z nami pilot?

Jak my mamy państwu wierzyć?

Jeżeli chodzi o tę salę, to pilotuję ja, jakoś daję sobie radę, chociaż nie wiem, czy dalej mi tak dobrze pójdzie, bo zapraszam do głosu pana posła Grzegorza Brauna, koło Konfederacji. Czcigodny Panie Marszałku! Wysoka Pustawa Izbo! Szczęść Boże! Panie i Panowie Ministrowie! Panie ministrze, cieszę się, że widzę pana, bo my w naszym kole popadliśmy w stany lękowe, że może pan jest jakąś postacią fikcyjną, jakąś kreacją Ministerstwa Cyfryzacji, wie pan, jakimś fantomem, którego nam pokazują w telewizji.

Pan premier powiedział: nie zawahamy się.

Proszę mi odpowiedzieć: Czy pan bez lęku zwiększa dług publiczny, czy może z lekką bojaźnią i drżeniem? I ostatnia kwestia, bo może nie będzie więcej okazji. Czy dalej jest pan owładnięty myślą o odebraniu Polakom gotówki, czy to już panu przeszło, panie ministrze?

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Nie będę oryginalny. Chcę zapytać, jak na dzień dzisiejszy mają się finanse publiczne w Polsce. Jakie są wydatki?

Myślę, że udzielenie Wysokiej Izbie odpowiedzi na to pytanie nie będzie wydatnym problemem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Grabczuka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polityka fiskalna jest jedną z najważniejszych spośród wszystkich polityk. Wspieranie ludzi, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą, którzy chcą być aktywni, a jednocześnie zachęcanie ich do prowadzenia tej działalności, to sprawy szczególnie ważne. Istotne jest nieobciążanie ich w sposób nadmierny podatkami, ponieważ wcześniej czy później to się źle kończy. Mieliście państwo najlepszą od kilkunastu lat koniunkturę gospodarczą na świecie. Przyszedł kryzys i okazuje się, że z tej koniunktury gospodarczej w zasadzie nic nie zostało. To w moim przekonaniu, ale chyba nie tylko w moim, była kreatywna księgowość. Proszę państwa, kryzys obnażył wszystko, co się dzieje. Ta silna pogoń za zrównoważonym budżetem, który de facto, jak wszyscy wiemy, nie był zrównoważony, również miała miejsce. Panie Ministrze!

Dziękuję panu. Zapraszam pana posła Jakuba Kuleszę, koło Konfederacji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiele lat temu Stowarzyszenie KoLiber - taka prawicowa masoneria, której członkowie później zostają posłami, wiceministrami, ze dwóch tutaj widzę - zorganizowało akcję „Polska bez długu” Forum Obywatelskiego Rozwoju umieściło fizyczny licznik przy rondzie Dmowskiego, który już dawno temu wybił 1 bln zł. Chciałem spytać pana ministra: Jak idzie ta walka o Polskę bez długu? Dziękuję serdecznie. Niedługo już się dowiemy, panie pośle, jak to idzie. A w tej chwili pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu ustawy, nad którą w tej chwili procedujemy, czytamy: Konieczność jak najszybszego wejścia w życie ustawy wynika z potrzeby nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Dalej piszecie panowie: niewprowadzenie proponowanych zmian uniemożliwia wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami w sytuacji ogłoszenia epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej. W efekcie bez wprowadzenia proponowanych zmian uruchomienie działań w ramach tarcz antykryzysowych musiałoby zostać skompensowane ograniczeniem innych wydatków. Przecież do tej pory słyszeliśmy, że wprowadzane tarcze nie wiążą się ze zmianą budżetu. Samorządy na terenie naszej ojczyzny wołają do rządu: panie i panowie, pochylcie się nad nami. Przedstawiają wam wiele różnych propozycji, a rząd, niestety, na te propozycje nie odpowiada.

Bardzo dziękuję za te rady.

Nigdzie nie powiedziałem, że chcę wykluczyć gotówkę w Polsce. Powiedziałem, że chcę, żeby obywatele mieli prawo do płacenia, jak chcą: albo gotówkowo, albo bezgotówkowo.

To, co ja mówię, to, co państwo mówią, to są oczywiście nasze perspektywy, ale najważniejsza jest taka reguła w finansach, w sektorze finansów, że ten, który ma pieniądze, decyduje.

Myślę, że nie jest najgorzej. Co do JST wszyscy mieliśmy i mamy kłopot z finansami w tym roku podczas tej pandemii.

Dlaczego nie nowelizujemy dzisiaj budżetu?

I to jest powód, dlaczego dzisiaj przychodzimy do Wysokiego Sejmu z projektem ustawy, żeby zawiesić przez rok SRW. Wtedy będę mógł zaproponować nowy budżet, nowelizację budżetu.

Będziemy wiedzieli, ile jest mniej podatków z powodu kryzysu gospodarczego, ile jest podatków, bo siadła gospodarka. A są one potrzebne, żeby rozkręcić naszą gospodarkę, żeby mogła bardzo szybko wyjść z tego kryzysu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę państwa, zamykam ten punkt. Dziękuję serdecznie za miłą współpracę.

Wznawiam obrady. Proszę zatem wszystkich państwa posłów o naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku.

obradach bierze udział 436 posłów. Stwierdzam kworum. Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, druk nr 391. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (druk nr 391) Bardzo proszę państwa posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. Na pamiątkę tamtego dnia w 2000 roku ustanowiono Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony co roku właśnie 27 maja. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce wywodzą się jeszcze z Konstytucji 3 maja. Samorząd istniał również na wszystkich ziemiach polskich objętych zaborami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadziła go także konstytucja marcowa z 1921 roku. Zlikwidowany w roku 1950 przez komunistów i przywrócony dopiero w 1990 roku. Samorząd terytorialny stał się podstawową formą lokalnego życia publicznego, najpierw na szczeblu gminy, a od 1999 roku - także na szczeblach powiatu i województwa. Reforma samorządu gminnego z 1990 roku to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 roku. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną, polityczną i ekonomiczną. Monopol państwowej własności i system centralnej władzy zostały złamane. 30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, wyraża uznanie i podziękowania za ten wysiłek na rzecz dobra wspólnego oraz zachęca do kolejnych lat budowania wspólnoty samorządowej” Proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę przez aklamację. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Proszę - 1 minuta. Szczęść Boże! Dobry wieczór. Pani Marszałek Czcigodna! Rządzie! Wysoka Izbo! Wniosek formalny o przerwę celem zwołania Konwentu Seniorów, celem szybkiego położenia kresu reglamentacji dostępu do tej Izby, do tej sali. Bardzo proszę skończyć z tą szopką. Pod pretekstem walki z mniemaną pandemią państwo w istocie sprowadziliście parlamentaryzm Rzeczypospolitej Polskiej do fasadowości, a za fasadowością obracacie w farsowość to nasze procedowanie.

Rozumiem, że to jest powtórzenie wniosku z rana, wniosek o przerwę. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 390. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły dodatkowe sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, - o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 257-A i 354-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące trzecie czytania tych projektów ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! W czasie przeprowadzonego drugiego czytania na sali plenarnej zgłoszono do ustawy jedną poprawkę. Komisja rozpatrzyła poprawkę, sprawozdanie zawiera w druku nr 365-A i rekomenduje Wysokiej Izbie poprawkę odrzucić i przyjąć całość projektu ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 365. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 365, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 364-A. Proszę pana posła Piotra Polaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić dodatkowe sprawozdanie zawarte w druku nr 364-A dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Podczas drugiego czytania tutaj na sali plenarnej zostało zgłoszonych pięć poprawek do tego projektu ustawy.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 364. W dodatkowym sprawozdaniu komisja przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 3. do 5., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 364, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 363. Komisja przedstawia wniosek mniejszości, nad którym głosować będziemy w pierwszej kolejności. We wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują dodać art. 8a określający maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego osób określonych w tym przepisie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 363, wraz z przyjętą poprawką, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 387-A. Proszę pana posła Bolesława Piechę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić dodatkowe sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. W trakcie drugiego czytania projektu ustawy na sali plenarnej zgłoszono 14 poprawek.

W czasie rozpatrywania poprawek wnioskodawcy wycofali poprawkę 3. Jednocześnie proponuję i w imieniu komisji zgłaszam, żeby Wysoka Izba całość ustawy przyjęła. Dziękuję. Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie z PiS! Zrobiliście dobrą ustawę. Chcieliśmy ją poprzeć, chcieliśmy móc głosować za nią, ale nie rozumiem, czemu znowu wkładacie ideologię, czemu do dobrej ustawy, która ma pomagać w kształceniu lekarzy, w dbaniu o ich zawód, wkładacie wasze pomysły ideologiczne. Pomysł z dołożeniem tutaj zapisów o klauzuli sumienia jest przede wszystkim nieetyczny, jest ograniczeniem dostępu do wiedzy, jest uderzeniem w prawa pacjenta i naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia. Jeżeli nawet chcecie iść na wojny ideologiczne, robicie to kosztem praw lekarzy. Te wasze zapisy nie pozwalają nam popierać tej ustawy, a szkoda. Szkoda, że każdą rzecz, którą robicie, musicie choć troszeczkę zepsuć, że wasze ustawy muszą być takie. Dlatego proszę, pani marszałek, o wycofanie tego punktu w tej chwili z porządku obrad i danie czasu na refleksję posłom wnioskodawcom i posłom z PiS, na usunięcie ideologicznych zapisów i przeprowadzanie normalnej, rzetelnej ustawy, która nie będzie uderzała w prawa pacjenta. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 387. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 12. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zwierającego zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. W 8. poprawce do art. 29 ust. 10 wnioskodawcy proponują inne brzmienie pkt 2. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 10.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. W 11. poprawce wnioskodawcy proponują inne brzmienie art. 53. Z poprawką tą łączy się poprawka 13. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 12.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 387, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie dyskusji zgłoszono poprawki oraz wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały po doręczeniu zestawienia poprawek. Poddam pod głosowanie wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały bez odsyłania do komisji. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm skierował projekt uchwały do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za propozycją przystąpienia do trzeciego czytania projektu uchwały zawartego w druku nr 384 po doręczeniu zestawienia poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Zgłoszone poprawki zostały paniom i panom posłom doręczone do druku nr 384. Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 384. Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu uchwały nowelizującej. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 2. poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 4. poprawki. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 384, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64, 257 i 257-A) - trzecie czytanie. Proszę panią poseł Annę Kwiecień o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić państwu sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 257-A, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, druk nr 64. W dniu wczorajszym odbyło się połączone posiedzenie obu komisji. na którym to posiedzeniu była rozpatrzona jedna poprawka wniesiona przez klub Lewicy.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 257. Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm będzie głosować w pierwszej kolejności. W poprawce do art. 3a pkt 4b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wnioskodawcy proponują, aby rekomendacje, o których mowa w tym przepisie, nie były wiążące. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 257,

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 268, 354 i 354-A) - trzecie czytanie. Proszę pana posła Cezarego Grabarczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Do projektu ustawy z druku nr 268 wniesiono tylko jedną poprawkę o charakterze legislacyjnym. W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała tę poprawkę i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy wraz z poprawką. Dziękuję, panie pośle. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 354. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W poprawce do art. 47 ust. 1 wnioskodawcy proponują zmianę odesłania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 354, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

za, nikt nie był przeciw, 12 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., podmiotów oferujących papiery wartościowe członków Grupy Kapitałowej GetBack S.A. oraz firm audytorskich badających sprawozdania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A. - zgłoszony przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; - Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego wyprowadzenia z Polskiego Krzyża blisko 3 mln zł, a w szczególności możliwości przeznaczenia przez działaczy PiS wyłudzonych środków w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do parlamentu w 2015 roku oraz wskazania w jakim zakresie badany był przez prokuraturę udział w przedmiotowej sprawie prominentnych działaczy PiS, Prezesa Rady Ministrów w sprawie wiedzy jaką posiadał na temat wykrytych nieprawidłowości i czynności podejmowanych w toku prowadzonego przez prokuraturę postępowania, a także wystąpienia możliwych powiązań sprawców popełnionego przestępstwa z politykami PiS, w tym z byłymi lub obecnymi członkami rządu - zgłoszony przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni; - Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat wdrażania zmian w wymiarze sprawiedliwości - zgłoszony przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym pierwszego czytania poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa dotyczącego wyprowadzenia z Polskiego Czerwonego Krzyża blisko 3 mln zł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym informacji na temat wdrażania zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382, 382-A i 390) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Szanowna Pani Marszałek! Wczoraj na posiedzeniu plenarnym odbyło się pierwsze czytanie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów w związku z COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pani marszałek po pierwszym czytaniu skierowała projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych. Komisja Finansów Publicznych przez wiele godzin, zakończyliśmy prace o godz. 4 nad ranem, rozpatrywała projekt. Do projektu zgłoszono kilkadziesiąt poprawek.

Dotyczyły one głównie uściślenia, uporządkowania i doprecyzowania zapisów, które wspierają przedsiębiorców, ale również zapisów, które regulują życie w okresie pandemii, m.in. również, oprócz oprocentowania, dopłat do oprocentowania kredytów, Prawa restrukturyzacyjnego, które zmieniamy na czas COVID i najbliższe lata po nim, aby zabezpieczyć polskie spółki o znaczeniu strategicznym przed przejęciem przez firmy spoza Unii Europejskiej, przez kapitał spoza Unii Europejskiej.

Natomiast rozwiązania, które są proponowane w innych zapisach ustawy, oczywiście też będą miały koszty budżetowe, ale również przede wszystkim koszty organizacyjne. Dotychczasowe zapisy poszczególnych tarcz antykryzysowych spowodowały, że Polska jest jednym z liderów ochrony miejsc pracy w Europie i bardzo trudna sytuacja, która jest związana z występowaniem epidemii, nie odbiła się w sposób znaczący, jak w innych krajach europejskich, na bezrobociu. Środki finansowe, które według informacji ministra rozwoju zostały przekazane polskim przedsiębiorcom, szczególnie poprzez Polski Fundusz Rozwoju, jako pożyczki w części umarzalnej na ochronę miejsc pracy, przekraczają już 30 mld zł. Stąd jest oczywiste, że wielu przedsiębiorców zostawia pracowników, korzystając z różnych form dofinansowania.

Takich czynności również należy dokonywać, stąd m.in. takie zapisy w kodeksach się pojawiły.

Uznaliśmy, że ważność spraw i pilność rozwiązań w zamianach kodeksowych są istotniejsze niż dochowanie pełnej procedury, dlatego komisja przyjęła również te rozwiązania. Ostatecznie komisja przedstawia Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, sprawozdanie jest zawarte w druku nr 390, i wnosi o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę. Panie Premierze! Wysoki Sejmie!

Według Centrum Informacyjnego Rządu ta pomoc może wygenerować kredytowanie kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych potrzebnych na refinansowanie już występujących kredytów przedsiębiorców na kwoty kilkudziesięciu miliardów złotych. Dopłaty do oprocentowania zabezpieczone klauzulą wpisaną w tej ustawie dla małych. Subwencją, dopłatą 2% dla mikroprzedsiębiorców i 1% przy zachowaniu średniego oprocentowania jako odniesienie stosowanego w poszczególnych bankach, które zawrą umowę w Banku Gospodarstwa Krajowego dla tego typu kredytów.

Proszę państwa, mielibyśmy w istocie budżet zrównoważony po kwietniu po stronie dochodów i wydatków, gdyby nie dodatkowe wydatki podjęte w tym roku. A więc rząd w sposób bardzo odpowiedzialny, wyważony kieruje cały czas intensywnie pomoc, ale też uzyskuje wsparcie od innych instytucji. Proszę zwrócić uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej odważnie obniżała stopy procentowe, dając oddech w spłacie kredytów hipotecznych i konsumenckich.

Ile razy rozmawialiśmy o tym, czy warto przyjąć euro, czy nie. Mamy własną politykę pieniężną, doskonałe narzędzie wykorzystywane przez mądrych ludzi w sposób odważny, elastyczny. Właściwie analitycy nie spodziewali się tej obniżki, a ona spowoduje, że osoby zadłużone w kartach kredytowych, w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, na kredytach gotówkowych zostaną po raz kolejny beneficjentami takiej polityki pieniężnej. Szanowni Państwo! Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przekonali się do licznych propozycji zgłoszonych również przez klub Prawo i Sprawiedliwość, przeze mnie. W miarę upływu czasu ta nasza dyskusja była coraz bardziej merytoryczna i wiele poprawek zostało popartych, ponieważ są probiznesowe.

To jest jednak nieodzowne przy takim gąszczu przepisów, które zostały użyte do wygenerowania pomocy publicznej.

Bardzo proszę, teraz pan poseł Dariusz Rosati, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Pani Premier! Szanowny pan poseł Janczyk dokonał świetnego podsumowania tarczy 4.0. Powiedział, że jest to gąszcz przepisów podlegający ciągłym korektom. Rzeczywiście dostajemy co 2 tygodnie, co 10 dni, co 3 tygodnie kolejne akty prawne, które są głównie poświęcone poprawianiu poprzednich aktów prawnych. Niestety muszę powiedzieć, że jeśli państwo posługujecie się nazwą „tarcza” w stosunku do tego dokumentu, to jest to nazwa mocno na wyrost. Powiedziałbym, że to raczej taka pokrywka, która, jeśli chodzi o wpływ na sytuację przedsiębiorstw, prawdopodobnie nie przyniesie specjalnych efektów. Był pan również łaskaw powiedzieć, że świetnie, że mamy własną walutę, wszyscy się z tego cieszymy, bo Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe do 0,1. Szanowni Państwo! Po pierwsze, dlatego że znowu otrzymujemy na ostatni moment projekt aktu prawnego liczący prawie 100 stron, który tylko w niewielkiej części dotyczy dopłat do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw, a w ogromnej części stanowi takie przyczynkarskie propozycje zmian do rozmaitych aktów prawnych, często niemających kompletnie nic wspólnego z epidemią COVID-19. Podam jeden przykład. W ramach tych poprawek, które zostały przegłosowane, mieliśmy np. poprawkę dotyczącą wynagrodzeń członków państwowej komisji do spraw zwalczania pedofilii, która miała być powołana w ubiegłym roku przez pana premiera, ale do tej pory nie została powołana.

W efekcie otrzymaliśmy coś w rodzaju grochu z kapustą i nawet posłowie partii rządzącej wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą, nie bardzo mieli orientację, w jakim właściwie kierunku zmierzają te zmiany i dlaczego poszczególne zapisy tej ustawy w ogóle znalazły się w tym głównym projekcie. Muszę powiedzieć, że główny zarzut, jaki stawialiśmy w przypadku tej ustawy, że ona jest procedowana za szybko, że jest przygotowana na kolanie, w sposób niechlujny, został wczoraj udokumentowany i potwierdzony, choćby takim faktem, że biuro analiz, przepraszam, biuro prawne, Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło, już nie pamiętam, kilkadziesiąt czy nawet więcej poprawek do tego tekstu. Chciałbym z tego miejsca podziękować prawnikom z Biura Legislacyjnego, bo wykonali rzeczywiście wspaniałą robotę. Jednocześnie ujawnili, jak niestarannie, jak nieprofesjonalnie, w jak amatorski sposób była przygotowywana ta ustawa. Dodatkowym dowodem na to, że to był bubel, który do nas trafił, był fakt, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zgłosili kolejne poprawki, czterdzieści kilka poprawek liczących ponad 60 czy 70 stron.

Jeszcze raz z tej trybuny chcę powiedzieć, że stanowczo protestujemy przeciwko tej formie i temu trybowi pracy Sejmu. Również pana marszałka chciałbym poprosić, aby pan na ręce pani marszałek przekazał wyrazy naszego oburzenia sposobem, w jaki traktuje się Sejm, izbę ustawodawczą w naszym kraju, rzucając nam projekty ustaw i dając 24 godziny, żeby się tymi prawami zajmować. Nie możemy oczekiwać pozytywnych efektów, jeśli chodzi o walkę z pandemią i skutkami kryzysu, nie możemy oczekiwać tego, że wszyscy będą zadowoleni w sytuacji, kiedy te akty prawne są przygotowywane na kolanie. Chciałbym w związku z tym, panie marszałku, poinformować, że klub Koalicji Obywatelskiej złoży poprawki do tej ustawy.

Pan poseł Adrian Zandberg, klub Lewicy.

Parę tygodni temu modne było, także tutaj, nagrywanie sobie filmików, na których politycy klaskali. Klaskał pan minister Szumowski, klaskała pani marszałek Kidawa, klaskali różni politycy partii rządzącej. Chcieli w ten sposób wyrazić szacunek dla pielęgniarek, dla rejestratorów medycznych. Muszę państwu przyznać, że nie brałem udziału w tej akcji, bo miałem poczucie, że my, politycy, jesteśmy ostatnią grupą, która powinna brać w niej udział, bo z naszej strony nie są potrzebne oklaski, tylko porządne pensje w budżetówce, nie oklaski, tylko dobre wyposażenie, nie oklaski, tylko bezpieczne warunki i godna praca. I bez tego, bez realnych działań te oklaski brzmiały po prostu fałszywie. Dlaczego o tym dzisiaj mówię, proszę państwa? Bo dzisiaj to klaskanie ze strony rządu się skończyło i rząd uderza w dokładnie tych samych pracowników budżetówki. Dzisiaj tym ludziom rząd chce poobcinać płace. Dzisiaj tych ludzi rząd straszy zwolnieniami. Dzisiaj kosztem tych ludzi, jak to ktoś ujął z ław rządowych wczoraj, cytuję: będziemy się ratować. Jeżeli z tych polskich szpitali nie wywozi się dzisiaj setek czarnych worków ze zwłokami, to nie jest to zasługa ani pana premiera, ani pani premierki, ani pana ministra Szumowskiego, tylko jest to zasługa ludzi, którzy często za psi grosz pracują dla polskiego państwa: ratowników medycznych, pielęgniarek, ale też pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, pracowników sanepidu i szeregowych urzędników, pani premierko. To dzięki nim właśnie Polska się nie zawaliła, a dzisiaj grozicie im zwolnieniami, dzisiaj grozicie im obniżaniem pensji. Proszę państwa, co macie dla tych ludzi? Macie dla nich arogancję, którą było widać w wypowiedziach pani minister pracy, która powiedziała, że jeżeli ktoś nie dostał postojowego, to może sobie iść do sądu. Dla pracowników handlu, dla kurierów, dla pracowników logistyki macie obniżkę pensji na kolejny rok. Zaproponowaliśmy wykreślenie tych antypracowniczych przepisów. Usłyszeliśmy, że te poprawki zostaną odrzucone. Usłyszeliśmy też po raz kolejny kłamstwa, że podobno te rozwiązania są popierane przez stronę związkową. Muszę powiedzieć, że mój telefon się wczoraj zagotował od połączeń od związkowców, którzy pytali mnie, czy wiem, kto to niby popiera, bo nie znają żadnego związkowca, który byłby za obcinaniem pensji, który byłby za ta ustawą. Żeby nie być gołosłownym, proszę państwa, trzy opinie. Największe związki. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: Ten projekt został stworzony właściwie wyłącznie z myślą o pracodawcach, z dążeniem do zagwarantowania korzyści wyłącznie dla biznesu. To jest zachwianie relacji pomiędzy pracą a kapitałem, nie tylko rażąco niesprawiedliwe, ale też grożące długotrwałym utrzymywaniem się kryzysu społeczno-gospodarczego. Za szczególnie niekorzystne uważamy zwolnienia w kolejnych jednostkach sektora finansów publicznych, niższe świadczenia dla zwalnianych pracowników, zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy, likwidację świadczeń społecznych. Nie ma na to zgody OPZZ. Drugi związek, mniejszy, Inicjatywa Pracownicza: Zapisy wynikające z projektu tarczy pokazują, że PiS uderza w interesy pracowników. Metody stosowane przez rząd to nic innego jak działanie na zasadzie kopiuj-wklej z czasów, kiedy Polską rządziła Platforma. Koniec cytatu. I wreszcie związek, który, zdaje się, powinien być wam bliski, NSZZ „Solidarność”: Prezydium Komisji Krajowej wyraża stanowczy protest przeciwko art. 58 ustawy. Propozycja ta jest dla „Solidarności” całkowicie nie do zaakceptowania. Niedopuszczalne jest, aby cenę zahamowania pogarszającej się sytuacji budżetu państwa miały ponieść osoby zatrudnione w sferze finansów publicznych. Koniec cytatu. Z tym się, proszę państwa, nic nie da zrobić. Skoro odrzucacie poprawki, które wykreśliłyby te złe, antypracownicze przepisy, to tę ustawę trzeba po prostu wyrzucić. A więc to właśnie zróbmy. Proszę państwa, przestańcie kłamać, przeproście związkowców i po prostu wycofajcie te antypracownicze przepisy. A jeśli poczta przeciążona przez pana Sasina nie działa dobrze i opinie związków zawodowych, OPZZ-tu i „Solidarności”, do rządu nie dotarły, to mam je tutaj dla państwa wydrukowane i niniejszym przekazuję pani premierce Emilewicz, zachęcając ją do lektury.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Państwo Ministrowie! Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zacznę od przytoczenia Wysokiej Izbie kilku cyfr. Według opublikowanych dzisiaj danych BCC 48%, 46% firm dostało jedynie jakąkolwiek pomoc w ramach dotychczasowych tarcz, 30% firm otrzymało tylko pomoc z PFR-u, 40% przedsiębiorstw, które złożyły wnioski o pomoc, nawet nie dostały do dnia dzisiejszego decyzji. Zza kolejnej, czwartej tarczy antykryzysowej rządu, dzisiaj trudno nie odnieść takiego wrażenia, wyłania się biała flaga, biała flaga rządu Zjednoczonej Prawicy. Te skandaliczne zapisy dotyczące pomocy osobom, które pozostaną bez pracy, najlepiej tego dowodzą.

Tej zapobiegliwości, pani premier, w dotychczasowych trzech tarczach i tej czwartej nie bardzo widać. Lepiej ratować mniejsze, małe, mikrofirmy i te większe, niż dzisiaj leczyć skutki czy za chwilę, za kilka tygodni, kilka miesięcy leczyć skutki w postaci rosnącego bezrobocia. Niezwykle dziwi nas jako Koalicję Polską to, z jaką niechęcią państwo podchodzicie od kilku tygodni, kiedy procedujemy nad kolejnymi tarczami w tej Izbie, do projektu dobrowolnego ZUS-u, projektu Koalicji Polskiej. To jest to rozwiązanie, które leczyłoby, nim przyjdzie choroba w postaci masowego wzrostu bezrobocia i lawinowego wzrostu liczby osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem.

Mówiąc o projekcie dobrowolnego ZUS-u, który jest niezwykle dobrze przez przedsiębiorców, i tych mikro-, i większych, i dużych, odbierany, dzisiaj trzeba powiedzieć jedno, że za kilka dni kończy się zwolnienie z ZUS-u, które państwo zagwarantowaliście przedsiębiorcom jedynie na 3 miesiące. Pani premier, co dalej? Co dalej? To właśnie obarczenie każdej działalności gospodarczej składką na ZUS może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach pracowników.

Bardzo byśmy prosili, żeby na to w ten sposób zwrócić uwagę. Oczywiście jako Koalicja Polska również, po raz czwarty, chociaż już nieco zrezygnowani, jesteśmy otwarci na to, żeby o dobrych rozwiązaniach w ramach tych tarcz rozmawiać. I pozwolę sobie pakiet kilku propozycji ze strony naszego klubu złożyć, licząc na to, że może nie do trzech razy sztuka, ale do czterech razy sztuka, i da się wspólnie porozmawiać o dobrych rozwiązaniach, nie dzieląc tej Izby na tych lepszych i tych gorszych, którzy też mają coś do powiedzenia w sprawie przeciwdziałania skutkom koronawirusa.

Dobry wieczór. Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Pustawa Izbo! Za pamięci - poprawki. 45 poprawek koła Konfederacja. Tak jest, tak jest. Jak sami nie będziemy siebie oklaskiwać, to kogóż to wzruszy, że i te wyrzucicie pewnie do kosza? Wystąpi tu pewnie sam marszałek z takim wynalazkiem, żeby poprawki zblokować na te słuszne, te niesłuszne. Tak to będzie. Ale my solidnie odrabiamy lekcje, przychodzimy tutaj do roboty, zakontraktowani przez naród dla Rzeczypospolitej, piszemy, składamy, głosujemy. Między młotem a kowadłem, między Scyllą a Charybdą, między specjalistami od księgowości kreatywnej i rolowania długu publicznego. Rozumiem, że dziś lotów wielkim helikopterem z dużymi pieniędzmi już nie będzie, więc pani premier ma czas, żeby tutaj nam się przysłuchiwać. A z drugiej strony właśnie nie wiem, czy młot, czy kowadło. Panie Przewodniczący Zandberg!

Ta maska, jedna z ostatnich już tutaj, w tej Wysokiej Izbie, ona akurat pasuje, bo właśnie tu się roluje dług, a tu jest inna perspektywa. Oddajcie portfele, Polacy. Lewica będzie lepiej wiedziała, jak wydać wasze pieniądze. No i cóż, między tymi ekstremami Konfederacja musi się jakoś odnaleźć. Staramy się odnajdywać merytorycznie.

Wysoka Izbo! Koniec maja. Koniec maja to znaczy, że epidemia w Chinach trwa 5 miesięcy, na świecie - 4 miesiące, w Polsce - 3 miesiące. A my mamy czwartą tarczę, mamy sprzeczną politykę ministra Szumowskiego, który najpierw w lutym ogłaszał, że w ogóle nie ma żadnego problemu, jesteśmy świetnie przygotowani, potem była trwoga i głupie kroki w stylu zamykania parków i lasów, później mamy wzrost zachorowań i pomimo tego wzrostu zachorowań rozmrożenie. Bo co? Bo sondaże. Sondaże was dopadły i zmęczenie rodaków kwarantanną was dopadło. Nie macie żadnego, najmniejszego, sensownego, konsekwentnego, przemyślanego, przepracowanego i własnego planu na walkę z tą epidemią. Nie posiadacie go, bo słuchacie np. skompromitowanego WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, która raz mówi: maseczek nie zakładać, drugiego dnia mówi: maseczki zakładać. I wy jak te barany posłusznie realizujecie to, co oni wam każą. Nie macie żadnego planu, bo jeśli mielibyście plan, to nie działalibyście pod dyktando globalnych organizacji lub sondaży, które dzisiaj wam mówią: trzeba w panice wszystko rozmrażać, bo się naród oburzył. Bo naród się oburza, jak widzi, że prezydent Duda robi tłok i ścisk po miejscowościach w Polsce, a łowicka pielgrzymka jest aresztowana. Taka jest prawda o tym, jaką hipokryzję reprezentujecie. I to widzi również chrześcijańska opinia publiczna w naszym kraju. 2 miesiące temu Krzysztof Bosak z tej mównicy apelował o to, żeby ulżyć kredytobiorcom, żeby obciążyć instytucje finansowe, a wy za czwartą tarczą poszliście po rozum do głowy i cokolwiek w tej sprawie robicie.

Teraz głos ma wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na początek chciałam tylko zrobić uwagę formalną. Ja rozumiem, że mój rozmiar nie jest zbyt znaczący, ale jednakowoż na każdym posiedzeniu Sejmu, na którym prezentowany jest projekt ustawy, który przygotowuję, zawsze jestem obecna, zawsze odpowiadam na pytania, co więcej, uczestniczę również w obradach komisji, a także podczas posiedzeń komisji odpowiadam. Ale odpowiadając na pytania i wątpliwości, które się pojawiły, przede wszystkim chciałabym podziękować za to komisji, za wytężoną pracę nad tym projektem ustawy, który, tak, zgodzę się, nie był prosty, nie był krótki, był wymagający, ale z całą pewnością był potrzebny. Odpowiem na pytania dotyczące złożoności, skomplikowania czy też kolejnej odsłony tarczy gospodarczej, dlaczego jest kolejna, dlaczego nie przygotowaliśmy od razu kompletnego, pełnego projektu. Tak, panie pośle, wszyscy zapewne się zgodzimy, że chcielibyśmy stworzyć kompletną architekturę legislacyjną adresującą wszystkie potrzeby wszystkich poszkodowanych, wszystkie potrzeby związane z epidemią, która rozpoczęła się w Polsce 13 marca. Tak chcielibyśmy zrobić i pewnie już dzisiaj po 2,5 miesiąca mielibyśmy gotowe rozwiązania zarówno dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego, jak i dla dużych firm, które utraciły płynność.

Tym wszystkim setkom tysięcy miejsc pracy, które dziś jeszcze są na rynku, a których zapewne za sprawą tej doskonałej legislacji wypracowywanej przez kolejne miesiące po prostu by nie uzyskali i po prostu dziś byliby kolejnymi zarejestrowanymi bezrobotnymi.

I za to państwu bardzo serdecznie dziękuję, przyznając, że na pewno wszystkie rozwiązania nie były doskonałe, przyznając, że musieliśmy je poprawiać. Ale zdecydowaliśmy się na taką inicjatywę legislacyjną, bo to po raz pierwszy, gdy.

Przypomnijmy, że w 2009 r., w czasie ostatniego kryzysu, ówczesny polski rząd zaproponował dość skromny pakiet wsparcia dla gospodarki, zdecydowanie za mały, biorąc pod uwagę skalę ówczesnego kryzysu. Uzasadniano wówczas, że bardziej ambitny pakiet spowodowałby kryzys na polskim rynku walutowym, skok inflacji i utratę wiarygodności. I dlatego po ówczesnym kryzysie znacznie więcej osób rejestrowało się w rejestrze bezrobotnych.

Tak, robimy wszystko, aby ci wszyscy, którzy kwalifikują się do tej pomocy, tę pomoc uzyskali. Dlatego wiele elementów uprościliśmy, teraz opierają się one na prostych formularzach, które sprawiają, że ta pomoc trafia naprawdę tak szybko, jak to możliwe. A tam, gdzie jest to niemożliwe, staramy się upraszczać procedury. Czy wówczas chcielibyśmy mieć sytuację włoską bądź hiszpańską, panie pośle? Odpowiadając, rozjaśniając jeszcze raz wątpliwości, które tutaj się pojawiły, w zakresie ochrony rynku pracy, jeszcze powtórzę, panie pośle, że te działania, które podejmujemy w każdej z naszych ustaw, są po to, aby utrzymać miejsca pracy.

I wówczas oczywiście moglibyśmy powiedzieć: nie pozwalamy, moglibyśmy powiedzieć: nie dajemy szansy przedsiębiorcom na to, aby byli w stanie udźwignąć koszty kryzysu, utrzymując miejsca pracy, jednocześnie przenosząc odrobinę tych kosztów na pracowników. My dajemy rozwiązanie, które, tak jak powtarzam, pozwala utrzymać miejsca pracy, obniżając pensje, ale jednocześnie dając nadzieję na to, że te miejsca pracy zostaną utrzymane, i dając szansę na wypłatę pensji przy wsparciu z budżetu państwa. Jak można ten pakiet nazywać pakietem antypracowniczym? To jest właśnie taka sytuacja, w której my podejmujemy działania na rzecz ratowania miejsc pracy. A zatem dziękując państwu za tę ogromną pracę dziś do wczesnych godzin porannych, jeszcze raz proszę Wysoka Izbę o przyjęcie tego projektu, bo na ten projekt czekają pracownicy, pracodawcy i samorządowcy. Pan poseł Grzegorz Braun w trybie sprostowania, ponieważ jego nazwisko było wymienione.

Chociaż mogą zaistnieć jakieś okoliczności łagodzące, jeśli proceder rozsypywania wirtualnych pieniędzy z wielkiego helikoptera będzie jakoś mitygowany, ograniczony. Dziękuję bardzo. Teraz w trybie sprostowania pan poseł Krzysztof Paszyk.

Panie Marszałku! Pani Premier!

Jeszcze raz powtarzam: tylko jedna trzecia przedsiębiorców skorzystała z PFR-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Dwa zdania. Pani zarysowała fałszywą alternatywę: albo można robić to, co wy, czyli ciąć pensje, albo można nie robić nic. I zasugerowała pani, że Lewica wolałaby nie robić nic. Otóż nieprawda. My uważamy, że robicie zbyt mało. Zaproponowaliśmy konkretne ustawy, wzorowane na rozwiązaniach duńskich, z dopłatami, które zagwarantowałyby utrzymanie wysokości pensji. To jest możliwe przy dzisiejszych kosztach obsługi długu zagranicznego. Nie zdecydowaliście się na przyjęcie gotowych rozwiązań, które wam przynieśliśmy. Pani Premier! Proszę w końcu powiedzieć, ile jest dzisiaj w Polsce zwolnień, ile jest w tym momencie już zwolnień grupowych, bo związki zawodowe od tygodni nie mogą się doczekać na uczciwe i niezafałszowane informacje na ten temat. A fala zwolnień grupowych w wielu branżach po prostu idzie. Więc o zwolnieniach, pani premier, naprawdę, kto jak kto, ale wy nie powinniście mówić. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina (druki nr 375 i 385) Proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Borysa Budkę o przedstawienie uzasadnienia wniosku. Wysoka Izbo! Cóż, nie ma nawet pana premiera Morawieckiego. Nie dziwię się, że nie przychodzi bronić skompromitowanego ministra Sasina. Nie dziwię się, bo to olbrzymi wstyd mieć kogoś takiego w rządzie. Żałuję, że nie mogę spojrzeć prosto w oczy panu ministrowi, jego wprost zapytać, czy nie wstydzi się tego, co zrobił, czy nie wstydzi się tego, w jaki sposób wyrzucił w błoto ponad 70 mln zł. Czy wiecie państwo, na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wynagrodzenie minimalne dla ponad 26 tys. osób, które straciły pracę. To wypłata postojowego dla ponad 33 tys. pracowników. To 138 tys. testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia czy oświaty. To 850 respiratorów, które mogły znaleźć się w polskich szpitalach. To ponad 1600 tys. maseczek - ale to po tej zawyżonej cenie od kolegi pana Szumowskiego, [[Oklaski]] bo po normalnej cenie to by było 17 mln maseczek. Ale co wolał zrobić rząd PiS? Co wolał zrobić rząd PiS rękami ministra Sasina? Wolał te 70 mln przeznaczyć na pseudowybory. Wolał je przeznaczyć na coś, co się nie odbyło. Co więcej, chciał to zrobić waszym kosztem, kosztem waszego zdrowia i życia, kosztem zdrowia i życia tych, którzy mieli te pakiety dostarczać, kosztem listonoszy, kosztem członków obwodowych komisji wyborczych. To nie doszło do skutku, ale do dziś nie wiemy, gdzie są te karty. Obiecuję, panie ministrze, że panu pomożemy znaleźć te 30 mln kart. Wie pan dlaczego? Bo w tej ustawie zapisaliście, że za zgubienie jednej karty można iść na 3 lata do więzienia. Zamiast 90 mln lat więzienia będzie pan odpowiadał tylko [[Oklaski]] za przekroczenie uprawnień i za wyrządzenie szkody majątkowej, a za to się idzie do więzienia na kilka lat. Wiecie, ile drzew wycięliście? Prawie 30 tys. drzew, tylko dlatego, żeby przeprowadzić te pseudowybory. Ale pan minister Sasin ma wiele takich dokonań. On jest, jak to niektórzy mówią, jak ten przysłowiowy król Midas, tylko w drugą stronę: za co się nie zabierze, to. A, nie będę mówił, w co się obraca. Nie wyszło. Chciał być metropolitą warszawskim, przeprowadzał referenda. Nie wyszło. Dopłaty dla Polaków do prądu miały być. Nie wyszło, nie ma tych dopłat, a prąd podrożał. Miały być sukcesy w górnictwie. Zapraszam na Śląsk, do kopalni, które pan premier ma nadzorować, a w których są ogniska koronawirusa, bo woleliście się zajmować wyborami.

Co pan by powiedział swoim przełożonym w Irlandii czy w Hiszpanii, gdy nadzorowali pana działalność w banku, gdyby pan spowodował straty 30 mld zł? Wiecie, co to są za straty, szanowni państwo? Przez 6 miesięcy nadzoru pana ministra Sasina nad spółkami Skarbu Państwa 13 kluczowych giełdowych spółek w akcjonariacie Skarbu Państwa straciło 31 mld zł. O tyle mniej wart jest majątek polskich podatników w spółkach nadzorowanych przez pana Sasina. Te 70 mln to jest taki pikuś. Panie Premierze! Czy pan bierze to na siebie? No bo pan premier Sasin dzisiaj się broni. Mówi, że to nie on wydawał te decyzje, to pan. Więc pytam: Czy państwo dzisiaj będziecie bronić pana Sasina, poświęcając pana premiera Morawieckiego? A może prezydenta Dudę? Bo o ile się nie mylę, to ósmego, w piątek, po wielkich naradach na Nowogrodzkiej, dziewiątego udaliście się w grupie kierownictwa PiS-u właśnie do Pałacu Prezydenckiego. A może poświęcicie pana premiera Gowina, który dotrzymując danego mi słowa, spowodował, że wyborów nie było w maju? Zdecydujcie się. To jest gigantyczna kompromitacja. Ale to jest pytanie o uczciwość, to jest pytanie o to, czy wreszcie zaczniecie ponosić konsekwencje za to, że wydajecie bezkarnie pieniądze polskich podatników. Okradliście podatników na 70 mln. I za to pan premier powinien podać się do dymisji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Bardzo dziękuję za aplauz opozycji. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posiedzenia. Niech pan się wstydzi, rzeczywiście, za to, co pan robi. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji Skarbu Państwa dotyczące tego wniosku, który został złożony w sprawie odwołania pana premiera Jacka Sasina.

Ale jako sprawozdawca - co prawda czas jest bardzo krótki - mam obowiązek przedstawić nie tylko wynik głosowania.

Ale po kilku minutach, po 2 czy 3 minutach, pan poseł przerwał i zaczął dyskutować z którymś z posłów i go strofować. Zapytałem, o co chodzi. No jak to? Tutaj pan poseł bezczelnie rozmawia przez telefon, zamiast słuchać wiekopomnego wystąpienia opatrznościowego męża stanu, który miał swoje życiowe przemówienie.

To jest sprawozdanie. Opowiadam po prostu, jak to wyglądało. Po czym po następnych 2 minutach pan premier Jacek Sasin odpowiedział na te wszystkie zarzuty, przedstawiając po prostu stan prawny i to, jak to wyglądało. zostawiając swoje wojsko bez dowództwa, można powiedzieć, na polu walki, przegranej bitwy, bo ta bitwa była przegrana. Szanowni Państwo! Po pierwsze, że wybory były przygotowywane. A drugi zarzut? Że tych wyborów nie było. Były zarzuty takie, że. No właśnie usłyszeliśmy tutaj, że pan premier nie zajmował się walką z COVID i na Mazowszu panowała zaraza. Rzeczywiście boskie przymioty ma pan premier, bo gdyby się zajmował, to nie byłoby pandemii.

Nie, spółki, które podlegały ministrowi aktywów.

że nawet część opozycji uznała, że ten wniosek był kuriozalny i całkowicie nieuzasadniony. Rekomenduję w imieniu komisji odrzucenie tego wniosku [[Oklaski]] jako skandalicznego, politycznego i przerzucającego wasze winy na premiera, który chciał.

Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję.

Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. Bardzo proszę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pan poseł Wojciech Zubowski. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera Jacka Sasina, dodajmy: najbardziej kuriozalnego wniosku, jaki pojawił się w ostatnim czasie, opartego wyłącznie na doniesieniach medialnych i wyrwanych z kontekstu fragmentach wypowiedzi. W uzasadnieniu Koalicja Obywatelska pisze wprost, że przed niebezpieczeństwem związanym z organizacją wyborów oraz głosowaniem uchronił obywateli wyłącznie wyraźny i stanowczy sprzeciw społeczny i konsekwentna praca opozycji. Wiemy już więc, komu możemy zawdzięczać to, że te wybory się wtedy nie odbyły. Ale mało tego, powszechnie wiadomo, że sprzeciw wobec wyborów 10 maja podyktowany był chęcią podmiany kandydata. Gdyby nie to, opozycja poniosłaby sromotną porażkę, a tak po prostu odsuwacie ją w czasie. Panie pośle, spokojnie. Ten wniosek nie pojawił się w związku z przygotowaniami Poczty Polskiej do doręczenia pakietów wyborczych obywatelom i przekazania ich do Państwowej Komisji Wyborczej, ale dlatego, że wicepremier Jacek Sasin okazał się skuteczny jako minister aktywów państwowych. Teraz zamiast skoncentrować się na walce ze skutkami epidemii, Platforma Obywatelska chce nadal destabilizacji sytuacji. Jeżeli państwo nie potraficie pomóc, bo wiem, że nie potraficie, to przynajmniej spróbujcie nie przeszkadzać tym, którzy wiedzą, jak to zrobić. Wbrew faktom okłamujecie Polaków, że Poczta Polska i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych organizowały wybory 10 maja. A te miały być przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, do której poczta miała dostarczyć wypełnione przez obywateli pakiety wyborcze. w ramach głosowania korespondencyjnego, co nie jest niczym nowym w polskim systemie prawnym. Mało tego, sami przecież państwo postulowaliście rozszerzenie tychże rozwiązań. Rozwiązanie to jest skutecznie stosowane w innych krajach. Jest czymś oczywistym, że skoro ustawa mówiła o przeprowadzeniu wyborów w trybie korespondencyjnym, należało podjąć odpowiednie przygotowania. Za czasów waszych rządów oczywiście nie byłoby to możliwe, ponieważ Poczta Polska była w ruinie. Irytuje was. Irytuje was, że mieliśmy rację, podejmując działania repolonizacyjne, wzmacniając pozycję spółek Skarbu Państwa. Dzięki skutecznej polityce właścicielskiej podmioty nadzorowane przez wicepremiera sprawnie i szybko włączyły się w walkę z epidemią. Ponad 173 mln zł wsparcia finansowego przeznaczono na zakup sprzętu medycznego i ochronnego dla szpitali, DPS-ów, laboratoriów. Przeprowadzono ogromne operacje logistyczne dostarczenia tych materiałów do potrzebujących ośrodków. Spółki udzieliły też wsparcia rzeczowego.

Mamy jeden z najniższych wskaźników ofiar śmiertelnych epidemii w Europie, ale to nie wzięło się znikąd, proszę państwa, to takie działania pomogły utrzymać go na tak niskim poziomie. To pokazuje, że kapitał ma narodowość i że jest to dla was niewygodne. Przypomnijmy, że przez lata usprawiedliwialiście swoją politykę kryzysem z roku 2008. Proszę państwa, dla przypomnienia, kiedy kryzys wybuchł w roku 2008, wy ustawę, która miała pomóc zwalczać jego skutki, wprowadziliście dopiero w lipcu roku 2009. Proszę państwa, okazuje się, że skutecznie można walczyć o polskie interesy, co nie podoba się też rosyjskim koncernom energetycznym, tak łaskawie traktowanym za waszych czasów, oczywiście kosztem polskich podatników. W czasie ostatniego półrocza, gdy ministrem aktywów państwowych był pan Jacek Sasin, PGNiG wygrał spór z Gazpromem, dzięki czemu mamy odzyskać ponad 6 mld zł. Wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie zmienił formułę cenową, która służy do ustalania ceny w kontrakcie jamalskim. Połączono Orlen z Energą, tworząc polską firmę energetyczną o europejskiej skali. Do tego za czasów rządów obecnej opozycji oferowano prezesom przekraczające granice zdrowego rozsądku i przyzwoitości milionowe odprawy. My ścięliśmy te kominy płacowe, dotrzymaliśmy słowa, pensje menedżerów są uzależnione od wyników finansowych spółek. Proszę państwa, obecne działania pokazują prawdziwe intencje Koalicji Obywatelskiej, która chce odwołania wicepremiera wzmacniającego pozycję narodowych przedsiębiorstw, ministra, który przeciwstawia się obcym wpływom w sektorze energetycznym i buduje (Dzwonek) niezależność Polski na arenie międzynarodowej. czyim interesie działacie? Dlatego też wnosimy o odrzucenie tego bezsensownego wniosku, mającego ukryć odpowiedzialność opozycji za brak wyborów prezydenckich 10 maja. które zablokowaliście, bo wymiana kandydata była dla was ważniejsza niż konstytucja, na którą tak często się powołujecie. Wnosimy o odrzucenie wniosku, bo chcecie odwołać ministra, który w przeciwieństwie do niektórych polityków opozycji w czasie epidemii nie uciekł na L4, tylko twardo stawił czoła wyzwaniu przeprowadzenia spółek przez ten trudny okres.

Panie Premierze!

Tyle wesołych rzeczy powiedzieć w jednym momencie, w jednej wypowiedzi. A, może do wesołości, takiej smutnej, tragikomicznej. Na przełomie lat 70. i 80. Wojciech Młynarski napisał świetną piosenkę: Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? To była piosenka, która krytykowała komunistów epoki Gierka, początków Jaruzelskiego. Ale mistrz Młynarski chyba nie przewidział, że będą takie czasy, że będzie rząd PiS-u i będzie taki mistrz świata od spieprzania jak premier Sasin. Nie będę powtarzał tego, co pan przewodniczący Borys Budka już mówił na temat pseudowyborów, głosowania korespondencyjnego. Dzisiaj poseł Kierwiński z posłem Tomczykiem pokazali, że gdyby te wszystkie pakiety wyborcze, które zostały wydrukowane, ułożyć jeden na drugim, to tzw. wieża Sasina miałaby 29,7 km. chciałem wystawić rachunek.

Tu, panie premierze Sasin, pan krzyczał, z tej mównicy, że zostanie ujawniony majątek żony premiera Morawieckiego. Wtedy mówiliśmy panu, że ta ustawa, której pan tak pilnował, zawiera błędy konstytucyjne i skończy w trybunale. Oprócz problemu żony pana premiera Morawieckiego mamy jeszcze problem z panią Szumowską.

Zastanawiam się, czy za chwilę nie będzie kłopotu z panią Sasin, bo problemy z oświadczeniem majątkowym pana premiera Sasina trafiły do CBA. Nie słyszałem, żeby ta sprawa się skończyła, panie ministrze.

Co by tu jeszcze, panowie, co by tu jeszcze? To jest jak z tym anty-Midasem, o którym mówił pan przewodniczący Budka. Nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej - pierwsze zdanie. Będą bardzo niskie - po jakimś czasie. Minęło kilka miesięcy - będą rekompensaty. Nic, tylko wzrosty. Raport Klubu Jagiellońskiego mówi wyraźnie: o 20 mld polska gospodarka miała wyższe koszty przez wzrost cen energii. A to jest tabela, jak rządzi pan Sasin. Rekordziści: 42% - PGE, 42% - PKP Cargo. Mój ojciec mówił, że chłopca od mężczyzny odróżnia tylko jedna rzecz: mężczyzna bierze odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Panie premierze Sasin, najwyższa pora wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.

Wysoka Izbo! Pan minister Sasin wydrukował karty wyborcze bez żadnego trybu, bez żadnej podstawy prawnej, a na końcu je zgubił. Nie wie, gdzie jest 30 mln kart do głosowania. To wszystko kosztowało nas 68 mln zł. Za te 68 mln można by dopłacić kilku tysiącom pielęgniarek do pensji, można być kupić 40 tys. komputerów do nauczania zdalnego. 30 tys. drzew poszło pod topór, żeby zorganizować wybory, których nie było.

Dziś mamy ponad 3 tys. zarażonych górników. Gdyby te 68 mln wydał pan na sprzęt ochronny dla górników, to chorych byłoby mniej. Panie Premierze! Na to są paragrafy: art. 231 i art. 296 Kodeksu karnego. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego i wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Zawiadomienie do prokuratury już poszło, a Trybunał Stanu czeka. Tyle faktografii. Zastanawiam się od pewnego czasu, jak to jest, że ludzie racjonalni zachowują się nieracjonalnie, jak ten wasz system działa. W wiem: „Cesarz”, Kapuściński, Etiopia, Hajle Sellasje: wszystkie zmiany od monarchy tylko pochodzić mogły, jego zgody i poparcia wymagały, bo inaczej przeniewierstwem się stawały. Trzy były grupy ludzi zabiegających o cesarza. Ci, którzy uważają, że wszystko mogą, lizusi i ci, którzy wiedzą, że albo będą rządzić, albo będą siedzieć. Zacznę od tych, którzy wszystko mogą. Pan premier je obiad, maseczki nie ma. Nie ma również rodziny. Lata w jedną i w drugą stronę z rodziną. Nie płaci za to. Dlaczego? Bo może. Całe Śródmieście zamknięte. Dlaczego tak się dzieje? Bo mogą. Kaczyński i cmentarz. Pan prezes Kaczyński jedzie na cmentarz. Inni nie mogą. Nie mogą. On może. Pokazała fucka całej Polsce, całej opozycji, wszystkim, wszystkim uczciwym ludziom. A wiecie, dlaczego jej nie ukarała? Bo mogła. Bo należy do kasty ludzi, którzy mogą. Trójka. Wiecie, proszę państwa, jak ten chłopak musiał się namanipulować i wymyślać, żeby temu prezesowi się podlizać? Znalazł tę piosenkę i sobie pomyślał: przecież prezes, jak to usłyszy, kiedy to będzie jedynka w Trójce, i jak ja to zdejmę, to może muśnie mnie wzrokiem, może się do mnie uśmiechnie, może mi powie „cześć”, może mnie w ogóle dostrzeże. Im większa kasa, tym większa wazelina. Policja - dobrze, spełnia swoją rolę, poza tymi, którzy sprawdzają rowery. A może ktoś zobaczy, że sprawdzę rower, zobaczy, że ktoś coś ma na tym rowerze, zobaczy, że ktoś jakiś plakacik zły o prezesie napisał. Zobaczę, jak to będzie. Urzędnicy - biorą pieniądze i co uznali? Uznali, że 500+ to jest jarkowe. Tak nawiasem, nie wstyd wam za to? Jest cytat w tej sprawie. Jeśli chodzi o hojność, to lepiej być hojnym, dysponując cudzą własnością, skąpym, jeśli chodzi o własne dobra. Lepiej budzić strach niż miłość. I teraz trzecia grupa: tych, którzy albo będą rządzić, albo będą siedzieć. Pan Sasin drukuje karty, bo szybkie wybory są potrzebne. Wie, że jak Duda przegra, będzie rozkład cesarstwa, wie, że pałac siedliskiem miernoty jest, zbiorowiskiem ludzi wtórnych, a ci w chwili kryzysu zawsze tracą głowę i starają się tylko ocalić własną skórę. Szliście po władzę, wmawiając wszystkim, że reprezentujecie ludzi i przychodzicie walczyć z elitami. Dziś widać wyraźnie: to wy jesteście tą elitą, która walczy z ludźmi. To wy jesteście elitą, która napełniła kieszenie ministra [[Oklaski]] publicznymi pieniędzmi, cenzuruje piosenki, bije ludzi na protestach. Traktujecie Polskę jak swój pałac. Dlatego w tym państwie taki minister jak pan Sasin powinien być odwołany.

Koalicja Polska. Po pierwsze, zdrowia dla pana premiera Sasina. Nie będę się nad nim pastwił, bo wy z niego na końcu i tak zrobicie kozła ofiarnego. Pomimo że zawsze najdzielniejszy uczeń, najbardziej pilny, zatańczy i zagra, zatańczy zawsze tak, jak mu prezes zagra, na końcu wchodzi znów pan prezes i mówi, że nie do rytmu, kroki nie takie, a tak naprawdę to nie ta piosenka. Pan Jacek się stara. Cały czas przekazem z Nowogrodzkiej nadaje. Później dochodzi do tego, że to nie ten przekaz i gadał nie do rzeczy. Szkoda trochę człowieka, bo robicie z niego kozła ofiarnego. Nie ma wyborów - wina Sasina. Prąd drożeje - wina Sasina. Nie ma rekompensat - wina Sasina. Majątek państwowy topnieje - wina Sasina. A wy czyste rączki, zdezynfekowane. Ale to nie tak, że to jest wina tylko Sasina. Ten wniosek nie jest wnioskiem wobec tylko i wyłącznie jednego ministra, wicepremiera, dzielnego żołnierza PiS-u, to jest wniosek przeciwko systemowi rządów, który wprowadziliście. On jest tylko i wyłącznie trybikiem w tym patologicznym, zepsutym świecie PiS-u, w tej patologicznej, zepsutej machinie, w tym systemie i układzie, które stworzyliście. Z wyborów prezydenckich zrobili czeski film. Najpierw sprawa druku kart. Nie wiadomo, kto te karty wydrukował, na jakiej podstawie, na czyje polecenie. Wiadomo za to, że karty zginęły. Co prawda część w Głogowie się odnalazła na ulicy i już byli ci szczęśliwcy, którzy jako jedyni w Polsce mieliby szansę zagłosować, ale ABW zajęło się sprawą. Nie potrafiła wskazać tego miejsca ani Państwowa Komisja Wyborcza, ani Poczta Polska. No, szacun, zgubić 30 mln kart - naprawdę trzeba się postarać. Prezes wam kota do pilnowania już więcej nie zostawi. Wiadomo, że te 30 mln kart, które zostały wydrukowane, to jest koszt 70 mln zł. O tym była już mowa. To jest 1400 firm, które mogłyby dostać dotację po 50 tys., to jest 27 tys. pensji minimalnych wypłaconych pracownikom, to jest 7 mln posiłków. To wszystko, co zrobiliście z tymi kartami, z wyborami, może byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było tak straszne. Taki napis, takie zdjęcie widziałem w Internecie: „Sasin, oddaj nasze 70 baniek. Polacy” Naprawdę do tego doprowadziliście państwo polskie, do takiej śmieszności? Wyborów nie byliście w stanie przeprowadzić, teraz mówicie, że to wina opozycji? Idźmy dalej. Ta telenowela z prądem, o której była już mowa. Najpierw miało nie być podwyżek, później podwyżki tylko niewielkie, a do tego zaraz rekompensaty. Rekompensaty miały być, jako zaliczki, już w styczniu, jest maj, nie ma żadnej ustawy o rekompensatach, nie ma żadnej propozycji, nie ma pracy nad tym w Sejmie. Ale są spadki spółek Skarbu Państwa. Za ostatni rok: Pekao - 44% w dół, PKO BP - 36% w dół, Bank Ochrony Środowiska - 20% w dół. Jak spółki energetyczne? Tauron - 26%, Enea - 30%, PGE - 50%. I nie mówcie, że to są spadki na giełdzie, bo giełda średnio spadła o 15%, a JSW - o 68, PKP Cargo - o 70%. To jest efekt rządów pana premiera Sasina, ale też całej machiny obsadzania samych swoich w spółkach Skarbu Państwa. Ich nie brakuje. Wymiany zarządów co chwilę, a za chwilę nacjonalizacja. Jacek Sasin jest tylko symbolem, jest znakiem firmowym waszych rządów, a tak naprawdę znaczkiem pocztowym za 70 mln zł. To jest esencja tak naprawdę i w nim się skupia cała filozofia sprawowania waszych rządów, nieudolnych, niekompetentnych, w systemie, który niestety wam na to pozwolił. Trzeba doprowadzić nie tylko do odwołania Jacka Sasina, ale do zmian ram ustrojowych, do zmian tej patologicznej filozofii, według której funkcjonujemy.

Wysoka Izbo! Wczoraj podczas prac komisji, które jak zwykle z właściwą sobie finezją, polotem i zwrotami akcji prowadził pan przewodniczący Marek Suski, mogliśmy wysłuchać mnóstwa rzeczy na temat Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dlaczego likwidujecie to ministerstwo? Dlaczego?

Nowogrodzka zaczęła tracić kontrolę nad polityką frakcji w spółkach Skarbu Państwa. To jest powód, dla którego pan wicepremier Sasin doświadczył zaszczytu i został wysłany na ważny front polityki partyjnej. Miało być jak w „Uchu prezesa”: spokojna konsumpcja owoców władzy, a nagle przyszła epidemia, przyszedł kryzys i trzeba drukować karty. Szanowni Państwo! Trochę współczuję panu wicepremierowi. Myślę, że koledzy z rządu się z niego podśmiewają. Pan wicepremier Gliński - za 70 mln go targają? Jak krew w piach.

Przepalone miliardy złotych. Przepalone bezsensownie za tej władzy. Przepalone po to, żeby obsadzać państwo kolesiami w najgorszym, SLD-owskim i platformianym tego słowa znaczeniu. To jest istota waszych rządów.

5 lat, podczas których sprawowana władza nie stała się narzędziem do uczynienia z Polski silniejszego, sprawniejszego bogatszego państwa, które rzeczywiście radziłoby sobie z problemami. Dlatego Konfederacja będzie głosowała za jego odwołaniem.

Resztę czasu wykorzysta pan poseł Krzysztof Bosak, koło Konfederacji. Panie Premierze! Panie Ministrze! Zrobiliście cyrk z kwarantanny. Zakazaliście ludziom pracować przy 100 zachorowaniach. Odmrażacie gospodarkę przy 400. Wykorzystaliście kryzys, żeby zaproponować kilka nowych podatków, nowe uprawnienia dla służb, żeby zamknąć Sejm. Ostatnio widzieliśmy nawet, że marszałek Sejmu ograniczyła Konfederacji miejsca z dwóch do jednego. To w ramach odmrażania. On ograniczył Konfederacji miejsca do zera i jeszcze został nagrodzony stanowiskiem. Być może gdyby pan marszałek wziął przykład, również dostałby jakieś dodatkowe stanowisko. Ale na razie jedyne, czego możemy tu doświadczyć, to kary za mówienie prawdy. Gdyby przez każde 12 miesięcy karać każdego z 11 posłów Konfederacji, to zaledwie po 343 latach uzbierałoby się brakujące 68 mln zł [[Oklaski]] wydane na wybory, których nie zorganizowaliście. Korzystajcie z pomysłów Konfederacji, tak jak robicie to na każdym posiedzeniu Sejmu.

Wysoka Izbo!

To jest logika, która mówi, że te wybory nie miały podstawy prawnej, podczas kiedy podstawę prawną daje konstytucja, wyraźnie mówiąc w swoim art. 128, kiedy wybory mają się odbyć.

Dzisiaj, kiedy słyszę zarzuty, że wybory nie odbyły się właśnie z tego powodu, że nie zostały przez nas, przez rząd należycie przygotowane, to przypominam sobie wypowiedź pana posła Budki, pana przewodniczącego, z 7 maja tego roku, kiedy demaskował, kto tak naprawdę do wyborów nie dopuścił. Mówił: Dzięki determinacji i stanowczości pani marszałek Kidawy-Błońskiej, determinacji senatorów opozycji i ciężkiej pracy parlamentarzystów, i stanowczej postawie samorządowców udało się doprowadzić do tego, że plan Kaczyńskiego przeprowadzenia wyborów 10 maja legł w gruzach. To są ci odpowiedzialni, Wysoka Izbo, za niedopuszczenie do wyborów i za straty, które z tego wynikają. A żeby pokazać tę logikę, to już 20 dni później, tylko tyle panu Budce wystarczyło, żeby całkowicie zmienić zdanie i powiedzieć, że całkowitą odpowiedzialność za to, że wyborów nie było, ponoszą rządzący. Tak wygląda, szanowni państwo, wasza logika i tym się kierowaliście, pisząc ten wniosek. A więc nie warto zagłębiać się w niego. Może warto powiedzieć, co jest prawdziwym powodem, dla którego chcecie odwołać mnie z funkcji ministra aktywów państwowych. To są działania, które od pół roku, bo tyle istnieje ministerstwo, którym mam zaszczyt kierować, podejmujemy i podejmuje rząd Zjednoczonej Prawicy. To jest całkowita zmiana filozofii, jeśli chodzi o majątek Skarbu Państwa. My repolonizujemy dzisiaj ten majątek, który rozsprzedaliście, pozyskując do Skarbu Państwa firmy, które zostały sprzedane, jak Pekao SA. My konsolidujemy, mądrze konsolidujemy spółki Skarbu Państwa, tak żeby dawać im szansę skutecznego działania i skutecznej konkurencji na europejskim rynku i dawać im również możliwości inwestycji. Dlatego doprowadziliśmy do fuzji Orlenu i Energi, dlatego chcemy i dyskutujemy dzisiaj z Komisją Europejską na temat fuzji Orlenu z Lotosem, dlatego również tworzymy holding spożywczy, po to żeby rzeczywiście to były mocne podmioty na polskim rynku. Tylko w tym krótkim, półrocznym okresie udało się uruchomić, podpisać umowę na budowę elektrowni Dolna Odra. To inwestycja za ponad 4 mld zł. Udało się stworzyć cały system finansowania, wielki, strategiczny dla polskich inwestycji, jakimi są Polimery w Policach - 7,5 mld zł. Przygotowujemy, Wysoka Izbo, również odpowiedzi na te wyzwania, które stanęły przed energetyką i przed górnictwem, te wyzwania, które są wynikiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dobrze by było, żebyście, szanowni państwo z opozycji, z Platformy Obywatelskiej, zamiast tak dzisiaj wylewać krokodyle łzy nad górnictwem i nad energetyką, przekonali swoich partnerów politycznych w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, że ta polityka dzisiaj jest dla nas bardzo trudna do zaakceptowania, bardzo trudna do wprowadzenia przy naszym modelu energetyki i górnictwa. Wolicie krytykować. Powołana została w Ministerstwie Aktywów Państwowych specjalna Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. W tym krótkim, półrocznym okresie przygotowaliśmy już projekty ustaw dotyczące prawa koncernowego, ustawę umożliwiającą przekazywanie przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom czy też ustawę, która zwiększa kompetencje rad nadzorczych. Mieliśmy również swój wkład w kolejne tarcze antykryzysowe, chociażby tworzyliśmy przepisy dotyczące uniemożliwienia przejmowania akcji polskich spółek w czasie kryzysu. Teraz, szanowni państwo, dodatkowo sukcesy międzynarodowe. Wspominał o tym pan poseł Zubowski, któremu za to dziękuję. Rzeczywiście wielki sukces, jeśli chodzi o nasze relacje z Gazpromem.

To jest ten rachunek, szanowni państwo posłowie i posłanki z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u, który powinien być wam wystawiony. 6,2 mld zł, które przepłaciliśmy przez ostatnie lata za rosyjski gaz, bo takie zawieraliście kontrakty z Gazpromem, tak nie dbaliście o polski interes narodowy. Wreszcie w tym krótkim okresie udało nam się uzyskać również bardzo korzystną decyzję niemieckiego regulatora rynku dotyczącą Nord Stream 2, który to regulator uznał, iż ta inwestycja, która nie jest korzystna dla Polski, zagraża polskim interesom, musi być poddana prawu europejskiemu, nie może być spod tego prawa wyłączona. To bardzo utrudnia dzisiaj realizację tej inwestycji, stawia ją być może nawet pod znakiem zapytania.

Państwo, zdaje się, nie zauważacie, że znajdujemy się w okresie kryzysu, który dotyka nie tylko Polskę, ale również cały świat. Chciałbym pokazać państwu ten ciekawy wykres. On pokazuje rzeczywiście notowania spółek Skarbu Państwa w czasach kryzysu obecnie i za czasów rządów Donalda Tuska.

Na drugim końcu tego wykresu - spadek, który mamy dzisiaj.

Dzisiaj, w czasach kryzysów związanych z koronawirusem - 23%. Jeśli chodzi o realne sumy, które wtedy straciliście na majątku państwowym, to same tylko udziały Skarbu Państwa w spółkach staniały wówczas o ponad 39 mld zł, a dodatkowo w czasie swoich rządów wyprzedaliście majątek narodowy o wartości 52 mld zł.

Takie są fakty, to nie demagogia, szanowni państwo. I wreszcie, co niezwykle ważne, udało nam się również doprowadzić do tego, że spółki Skarbu Państwa służą obywatelom.

Dlatego włączyliśmy się - Ministerstwo Aktywów Państwowych i spółki, które są przez ministerstwo nadzorowane - bardzo mocno w akcję wsparcia walki z koronawirusem.

Chodzi o cały zestaw działań, które w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie dały nam realne narzędzia do tego, żeby skutecznie walczyć z koronawirusem. Gdybyśmy tych spółek nie mieli, gdybyśmy posłuchali was i waszych ideologów ekonomicznych, szanowni państwo z opozycji, którzy mówili, że majątek państwowy w gospodarce należy wyrugować, że kapitał nie ma narodowości, że to nie ma znaczenia, czy mamy w Polsce polski kapitał, tobyśmy takich narzędzi nie mieli.

Wysoka Izbo!

Proszę zapamiętać tę sumę.

Tak zarządzaliście, szanowni państwo, spółkami.

Ale można powiedzieć: to abstrakcyjne liczby. Jak one się przekładają na sytuację Polaków? Otóż przekładają się, to bardzo proste. Chodzi o ceny benzyny, które Polacy musieli płacić na stacjach Orlenu w maju 2014 r. Kto wtedy rządził? Tak, szanowni państwo, koalicja PO i PSL, ci państwo, którzy dzisiaj chcą odwołania ministra aktywów państwowych.

Maj 2020 r., teraz, w realnej rzeczywistości, cena paliwa na stacjach benzynowych Orlenu to 4 zł, a na niektórych stacjach nawet mniej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wasz wniosek o wotum nieufności jest wielkim waszym przyznaniem się do błędu, wielkim przyznaniem się do winy. Jest rzeczą jasną dla Polaków, że stosowaliście całą paletę uników po to, żeby do tych wyborów nie doprowadzić. Najpierw obwieściliście światu, że są śmiercionośne koperty, zabójcze koperty. Pamiętamy wszyscy, jakie to miało być niebezpieczne. Pamiętamy doskonale obstrukcję Senatu, chociaż oczywiście już w trakcie pandemii marszałek Senatu wyjechał na narty do Włoch, więc chyba tam się nauczył strajku włoskiego. Z tego względu rozumiem, że ten strajk włoski stosował wtedy i stosuje go dzisiaj. Dzisiaj jednak Polacy już coraz mniej rozumieją, skąd bierze się taka potrzeba obstrukcji. Te wszystkie uniki, które stosujecie, już dzisiaj z całą pewnością przekładają się na to, że dla Polaków stało się jasne, że trzeba było wtedy działać w takich warunkach, w jakich się znajdowaliśmy. Wasz wniosek o odwołanie pana premiera Sasina jest kuriozalny, ponieważ znajduje się tam zarzut, Wysoka Izbo, że pan premier Sasin działał. Otóż działał po to, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. Tak, konstytucja. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak pan marszałek Senatu po 2 tygodniach podjąłby decyzję o tym, żeby ta ustawa jednak mogła wejść w życie na czas. Wtedy jak by wyglądał wniosek Koalicji Obywatelskiej? Otóż zapewne tak, że pan premier Sasin nie działał. Jak wiemy doskonale z praktyki, zawsze znajdzie się jakiś powód do tego, żeby wysunąć absurdalne zarzuty. Absurdalność tego zarzutu polega właśnie na tym, że do wykonania obowiązków konstytucyjnych potrzebne było działanie pana premiera Sasina. że podejmowane były działania w Ministerstwie Aktywów Państwowych i w innych miejscach po to, żeby wybory przeprowadzić. Natomiast to wasz strach ogromny przed gigantyczną porażką doprowadził do tego, że wasz marszałek Senatu przetrzymywał rzeczywiście. A więc my w konstruktywny sposób zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie. Dzisiaj znowu. Senat i marszałek Senatu zamrażają ustawę po to tylko, żeby opóźnić cały proces wyborczy, po to, żeby wybory nie mogły się odbyć w normalny sposób.

Dlatego najpierw, kiedy epidemia była w najtrudniejszym stadium rozwoju, i wszyscy doskonale o tym wiedzą, że w takim stadium była, zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne. Wasza obstrukcja doprowadziła do tego, że one były operacyjnie niemożliwe do przeprowadzenia. Dzisiaj proponujemy wybory w trybie tradycyjnym i jednocześnie też korespondencyjnym. To jest miara dobrej woli oraz miara tego, w jaki sposób, jak konstruktywnie staramy się podejść do tego tematu. Dodatkowo chcę podkreślić rolę pana premiera Sasina i podziękować mu, panu premierowi, za znakomite działania podczas tej pandemii koronawirusa. Pan premier Jacek Sasin był i jest członkiem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. PC. ...i specjalnego zespołu do zarządzania kryzysem gospodarczym. Ha, ha, ha! ...doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy z dumą zaprezentować pewien wykres. Ja bardzo lubię wykresy, jak wiadomo. A więc, szanowni państwo, tutaj jest pewien bardzo ciekawy wykres jednego z instytutów hiszpańskich, tak żeby... ...Santandera? Bo chwaliła nas ostatnio prasa francuska, „Le Figaro”, możecie sobie poczytać natomiast tutaj jest instytut hiszpański. I otóż tutaj są państwa Europy. Na jednej osi jest ochrona przed COVID-19, skuteczność tej ochrony mierzona liczbą zgonów na milion mieszkańców - to jedna z najbardziej ważkich miar, jakimi możemy potraktować sukces w walce z koronawirusem. Na osi poziomej jest wpływ na gospodarkę.

I to jest również zasługa pana premiera Sasina.

Tu warto podkreślić, szanowni rodacy, drodzy rodacy, pewną taką zależność. Otóż kiedy Senat Koalicji Obywatelskiej i sojuszników z Lewicy i z PSL przez miesiąc zastanawiał się, co zrobić z ustawą, my w 2 tygodnie przygotowaliśmy tarczę, która pobiera dane ze wszystkich możliwych systemów. ZUS, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Krajowa Administracja Skarbowa, środki europejskie i wszystkie inne, po to, żeby wiedzieć, czy dana instytucja, która potrzebuje wsparcia, jest rzeczywiście instytucją godną zaufania. I w ciągu 2 tygodni przygotowaliśmy tarczę, która działa od miesiąca. Ja mam do pana premiera Sasina nie tylko pełne zaufanie, ale mam pełne przekonanie, że pan premier Sasin jest najlepszą osobą stojącą na straży polskiego kapitału, polskich spółek Skarbu Państwa, polskiej własności.

Mówiliście: wybory są bezprawne, ale z drugiej strony, jak już sami doprowadziliście do tego, że one nie mogły się odbyć.

Ale one odbędą się w tym terminie konstytucyjnym, również dlatego że mamy ludzi godnych zaufania, pełnych determinacji, odwagi, odwagi podejmowania decyzji w trudnym czasie, w krytycznym czasie pandemii koronawirusa. I taką osobą jest właśnie pan premier Jacek Sasin.

To, że pomagaliśmy przedsiębiorcom i pomagamy, po to żeby ratować miejsca pracy, to skutek pracy również pana premiera Jacka Sasina w naszych zespołach gospodarczych, w rządowych zespołach zarządzania kryzysowego. Nie macie pojęcia, w jakim trybie podejmowane były tam decyzje. Tam pracowaliśmy 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Tymczasem nasze działania, działania dotyczące obrony miejsc pracy, szanowni państwo, drodzy rodacy, doprowadziły do tego, że dzisiaj przyrosty bezrobotnych, ale boli nas każdy bezrobotny, są jedne z najniższych w Europie. Jedne z najniższych w Europie. Tymczasem we Francji, w jednym z najbogatszych krajów świata, bezrobocie zaczyna sięgać 5 mln. Kilkaset tysięcy więcej osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. W Stanach Zjednoczonych liczba osób pobierających zasiłek przekroczyła 40 mln. To dla tych gospodarek są dane apokaliptyczne. Dla gospodarki hiszpańskiej to gwałtowny przyrost bezrobocia o blisko 1 mln osób.

O 1 mln osób wzrosło bezrobocie, a więc tak szybko trzeba było wtedy działać. Tarcza w Hiszpanii do dzisiaj jest nieobecna, tarczy w Hiszpanii do dzisiaj nie ma, tarczy w takim wymiarze, jaką my skonstruowaliśmy, takiej, o jakiej pan przewodniczący Budka z panem przewodniczącym Kosiniakiem tu po cichu rozmawiali, chwaląc tę naszą tarczę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Światowy kryzys o nieznanych do tej pory proporcjach. A co robi w tym czasie opozycja? To już jest zmysł destrukcji, który wkradł się w wasze szeregi. I apeluję, żebyście tego nie robili. Teraz potrzebna jest Polsce jedność, jedność rządu, Sejmu, prezydenta. I w związku z tym, podkreślając bardzo dużo tutaj wątków, o których była mowa w wystąpieniu pana premiera Sasina, chcę raz jeszcze podkreślić jedną rzecz, o której pan premier wspomniał. I ona jest bardzo ważna, ponieważ wystarczy podsumować okres waszych rządów i nadzór nad Skarbem Państwa, kiedy z liczby spółek nadzorowanych 1400 spadła ta liczba spółek do 400, a więc nastąpiła wielka wyprzedaż majątku, również spółek wielkich, takich, które dzisiaj są perłami w polskiej koronie, w koronie polskiej gospodarki. My repolonizujemy, my dokonujemy repatriacji polskiego kapitału do Polski z eksportu. To jest jedyna mądra polityka, która odwraca te wasze błędy gospodarcze 25 lat, blisko 25 lat, które doprowadziły do tego, że dzisiaj nasze zadłużenie względem zagranicy cały czas jest za wysokie. Ale chcę powiedzieć szanownym państwu, Wysokiej Izbie i drogim rodakom, że ono się zmniejsza i zmniejsza się właśnie dzięki polityce gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, polityce gospodarczej, której współtwórcą jest pan premier Jacek Sasin.

Gdyby nie to, moglibyśmy dzisiaj mieć lepszy współczynnik produkcji krajowej leków, bezpieczeństwa medycznego, również na czasy epidemii. Dzisiaj siedem na dziesięć leków jest niestety zagranicznych, ale to jest prosta konsekwencja tej wyprzedaży. Premier Jacek Sasin stoi na straży własności polskiej, własności Skarbu Państwa i robi to dobrze w tych bardzo trudnych czasach, do których można porównywać się tylko na zasadzie takiej właśnie, jak zostało to tutaj pokazane. Premier Jacek Sasin bardzo dobrze dba o polską gospodarkę, o polskie spółki Skarbu Państwa, a jego działania w okresie pandemii zmierzające do tego, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny, są godne pochwały.

Bardzo dziękuję, panie premierze. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy za chwilę. Ogłaszam przerwę do

Wznawiam obrady. Po przerwie, proszę państwa, przed głosowaniami mamy kilka. Sprawdzimy jeszcze raz kworum, w związku z czym bardzo państwa proszę o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu sprawdzenia kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Proszę bardzo, pan Robert Winnicki, Konfederacja.

Wysoka Izbo! Dzisiaj jest ważna rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego pod przewodnictwem pana prof. Andrzeja Zolla, szanowanego przez wielu w tej Izbie, zwłaszcza po tej stronie Izby. W uzasadnieniu tego wyroku czytamy: Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. Wysoka Izbo!

Porządek obrad został ustalony. Proszę bardzo, pan Borys Budka, Koalicja Obywatelska, wniosek formalny.

Kupowaliście Pekao SA - 123 zł za akcję. I jeszcze będziecie chcieli tworzyć jakąś narodową sieć sklepów spożywczych. Jesteście większymi socjalistami niż Marks, Engels, wszyscy razem wzięci. Naprawdę nie nadajecie się do zarządzania polską gospodarką. Nie nadajecie się do niczego. Pan broni Sasina? 30 mld mniej są warte aktywa spółek Skarbu Państwa po 6 miesiącach nadzoru przez pana Sasina. Pan poseł złożył wniosek o przerwę. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy?

Proszę nie dyskutować, panie pośle.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 386. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 386, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 392-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych wpłynęło osiem poprawek. Komisja rozpatrzyła poprawki i rekomenduje wszystkie poprawki odrzucić. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 392. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują tytułowi ustawy nadać brzmienie: o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania.